Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

W dniu dzisiejszym odbędą się również posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych: - Parlamentarnego Zespołu ds. Cyfryzacji - godz. 11, - Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki - godz. 11, - Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego - godz. 13. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw: - o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, - o zmianie ustawy o sporcie. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1605 i 1604. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Posłowie Barbara Dziuk, Andrzej Gawron i Ewa Malik z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chcą zadać pytanie w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 131 i nr 182 łączącej Katowice przez Tarnowskie Góry z lotniskiem GTL Katowice - do ministra infrastruktury.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W minionych dniach podpisano umowę na projekt modernizacji linii kolejowej nr 131, odcinek Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Herby Nowe pomiędzy PKP PLK a firmą Systra. Opracowanie dokumentacji projektowej to pierwszy etap inwestycji, której efektem będą lepsze podróże i przewóz towarów między Nakłem Śląskim a Herbami Nowymi na linii nr 131 z południa na północ Polski. Przygotowana inwestycja jest ważna dla poprawy przewozów towarowych w stronę Lublińca i Kluczborka, Inowrocławia, Bydgoszczy oraz Gdańska i Gdyni. Realizacja projektu zwiększy możliwości przyjaznego środowisku transportu kolejowego zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Również, panie ministrze, są już prowadzone czynności związane z rewitalizacją linii nr 182, która będzie łączyć cały region: z Katowic przez Tarnowskie Góry, lotnisko GTL Katowice znajdujące się w powiecie tarnogórskim przez Zawiercie do Katowic. Jest to jedna z największych inwestycji w województwie śląskim. W związku z powyższym zwracam się do pana ministra z następującym zagadnieniem: w jakim czasie jest przewidywane uruchomienie trasy, która jest potrzebna zarówno dla taboru pasażerskiego, jak i towarowego? Wiemy doskonale, że to działanie było podjęte przez rząd z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i za to chciałam bardzo podziękować. Panie Ministrze! Dodam tylko, że te inwestycje, o których mówiła pani posłanka, rzeczywiście bardzo mocno rozwijają kolej, jeżeli chodzi o Śląsk, o ruch pasażerski i towarowy.

Dziękuję bardzo. Dziękuję za zadanie pytania. Panie ministrze, proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście to są ważne pytania, ważne sprawy. Można powiedzieć, że linia nr 131 Śląsk - porty jest niezwykle istotna z punktu widzenia interesów nie tylko województwa śląskiego, ale i naszych portów w Gdańsku i w Gdyni.

Jeśliby doliczyć to, co planujemy w kolejnej perspektywie w ramach LOT-u B, łącznie daje to grubo ponad 4 mld zł inwestycji w ramach linii nr 131.

Tutaj bardzo wiele działań związanych jest właśnie z infrastrukturą pasażerską, z modernizacją przystanków, dobudową nowych przystanków. Mamy tutaj do czynienia z wieloma działaniami związanymi też z poprawą bezpieczeństwa, przebudową przejazdów kolejowych, budową dwupoziomowych skrzyżowań, m.in. z autostradą A1 czy drogą wojewódzką 913.

Zakładam, że marszałek śląski ułoży najlepszą z możliwych ofert dla przewozów regionalno-aglomeracyjnych.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Chciałam poruszyć temat trasy Sosnowiec - Pyrzowice, ponieważ od kilku tygodni trwa tam bardzo duży remont obwodnicy wschodniej. Stąd też bardzo trudno dostać się na lotnisko. Mieszkańcy Zagłębia pokładają nadzieję w tym, że w niedalekiej przyszłości drogę na lotnisko będą mogli odbyć pociągiem, w szczególności właśnie linią nr 182 Zawiercie - Pyrzowice. Mam pytanie do pana ministra: Jaka jest to perspektywa czasowa? Jaki jest stan zaawansowania budowy stacji kolejowej w Pyrzowicach i peronu trzeciego w Zawierciu, który jest budowany pod tę linię kolejową? I pytanie od mieszkańców: Czy jest zaplanowany przystanek w Porębie na tej linii? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo.

Oczywiście stacja Zawiercie będzie podlegała modernizacji, stacja Siewierz, stacja Miasteczko Śląskie Żyglin. Zostaną zmodernizowane perony na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba - czyli to, o co pani poseł teraz pytała. Nowe przystanki to Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów oraz stacja Pyrzowice Lotnisko.

Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu, dziękuję panu ministrowi. Proszę państwa, przechodzimy do pytania drugiego w sprawie drastycznych podwyżek opłat lotniskowych oraz ich skutków dla portów lotniczych. To pytanie będzie w pierwszej turze zadawał pan poseł Piotr Adamowicz, a w drugiej pan poseł Tadeusz Aziewicz z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Odpowiadał będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Marcin Horała. Bardzo proszę pana posła Piotra Adamowicza o zadanie pytania. Panie i Panowie! Wraz z posłem Aziewiczem zabieramy głos nie tylko w imieniu własnym i w obronie lotniska w Gdańsku, mówimy także, co chcę wyraźnie podkreślić, w imieniu wielu innych posłów z polskich miast i w obronie innych polskich lotnisk. Na skutek COVID cała branża lotnicza w 2020 r. poniosła dotkliwe straty finansowe.

Oczywiście straty poniosła także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Żeby przetrwać kryzys PAŻP, w agendzie rządowej proponuje się drastyczną podwyżkę opłat lotniskowych, szczególnie terminalowej, dla polskich lotnisk regionalnych aż o 70%. Tak o 70%. Przewidywane skutki: ceny biletów w górę, ograniczenie siatki połączeń, spadek rentowności lotnisk, obniżenie ich konkurencyjności itd., itd.

Należy mówić też o odłożonych w czasie negatywnych skutkach dla szeregu gałęzi gospodarki, zwłaszcza turystyki. W związku z tym pytanie: Dlaczego zamiast podwyżek opłat, czyli przerzucania problemów PAŻP na pasażera, przewoźników i lotniska, państwo nie obejmie pomocą finansową Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej? Należy przypomnieć, że odpowiednie instrumenty jednak potrafiono znaleźć np. w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, w Czechach czy w Estonii. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, panie pośle. Panie ministrze, zapraszam uprzejmie. Wysoka Izbo! Państwo posłowie, bo tu duża grupa posłów jest, pytają o podwyżki opłat lotniskowych. Opłaty lotniskowe są to opłaty, które nakładają zarządzający lotniskami na linie, w większości są to lotniska samorządowe, i ministerstwo, szczerze mówiąc, nie ma jakiejś wiedzy na temat planów zarządzających tymi lotniskami. Domniemywam, że nie chodzi o opłaty lotniskowe, tylko o opłaty nawigacyjne, trasowe i terminalowe. Te opłaty ustalane są w procedurze, która jest jednolita dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, której generalnym założeniem jest to, jeżeli chodzi o koszty kontroli przestrzeni powietrznej, czyli pewną usługę, która jest wykonywana na rzecz przewoźników, która dla ich biznesu jest niezbędna, żeby oni mogli swój biznes prowadzić, przewoźnicy muszą zarabiać i muszą taką usługę kontroli przestrzeni powietrznej mieć, ale z drugiej strony nie da się kontroli przestrzeni powietrznej inaczej zorganizować niż przez jedną państwową instytucję. Nie sposób sobie wyobrazić tego w formie jakichś prywatnych usług, gdzie byłoby kilku konkurencyjnych kontrolerów w tej samej przestrzeni powietrznej. A więc przewoźnicy generują pewien koszt, prowadząc swój biznes, i ten koszt powinien być przez nich pokrywany. Z powodu kryzysu na rynku lotniczym po-COVID-owym liczba operacji lotniczych się zmniejszyła. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wykonała cały szereg działań ograniczających koszty po jej stronie, dzięki którym w tej kilkuletniej perspektywie oszczędzony zostanie 1 mld zł. Ale te działania mają swoją naturalną barierę, tzn. kontrola przestrzeni powietrznej musi być zapewniona i to generuje pewne koszty, poniżej których zejść się nie da. Siłą rzeczy efektem matematycznym jest to, że jeżeli pewien koszt jest dzielony na mniejszą liczbę operacji, to koszt operacji wychodzi większy i stąd proponowane w ramach negocjacji dotyczących aktualizacji planu skutecznego działania podwyżki opłat terminalowych i trasowych. Chciałbym zaznaczyć, że takie podwyżki mają miejsce w całej Europie.

To jest taka instytucja afiliowana przez Komisję Europejską, która właśnie zbada, czy faktycznie jest tak, czy dochowano tych zasad, czy to są rzeczywiste koszty, czy ich nie zaniżono, czy nie dokonano tu jakiegoś ukrytego subsydiowania. W związku z tym, serdecznie ubolewając nad tym, że takie podwyżki są, musimy też mieć świadomość ich skali. Jeżeli mówimy o podwyżce o 70% dla portów regionalnych, to to jest podwyżka jednocześnie o kilkaset złotych na operację, czyli w przeliczeniu na jeden fotel, na jeden bilet trochę to będzie się różniło w zależności od samolotu, bo różne są samoloty, różną mają liczbę foteli, będzie to między 3 zł a maksymalnie 5 zł, pewnie najczęściej ok. 4 zł, przy założeniu, że przewoźnik będzie chciał na cenę biletu te koszty przerzucić. Tak jak mówię, jest to ubolewania godne i chcielibyśmy tego uniknąć, ale niestety realia są takie, jakie są i matematyka jest, jaka jest, koszty kontroli przestrzeni powietrznej są, jakie są. Proponowana przez państwa posłów bezpośrednia dotacja do PAŻP jest oczywiście prawnie możliwa, aczkolwiek niezwykle rzadko stosowana. Eurocontrol rekomenduje rozwiązania kredytowe.

W Polsce udało się z Banku Gospodarstwa Krajowego z gwarancją Skarbu Państwa zapewnić Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej kredyt na lepszych warunkach niż ten proponowany przez Eurocontrol.

Gdyby te podwyżki były zawyżone, one nie są zawyżone, ale gdyby były zawyżone, to po kolejnym okresie rozliczeniowym PAŻP musiałby po prostu zwrócić środki, musiałby tak obniżyć na następny okres rozliczeniowy opłaty, żeby to skompensować.

Te koszty są względnie wysokie, choć nie najwyższe w Europie i nie najwyższe w Europie Środkowo-Wschodniej, a skala podwyżek, opłat trasowych jest nawet poniżej średniej europejskiej. Wynika z tego, że mamy w Polsce bardzo rozproszony model transportu lotniczego, infrastruktury lotniczej. Wiemy, o co tu chodziło, o to, żeby wspierać penetrację polskiego rynku przez huby niemieckie, przez linie lowcostowe, a obniżać wartość polskiego, narodowego przewoźnika, żeby LOT pewnie gdzieś tam w planie na końcu sprywatyzować za ułamek jego potencjalnej wartości.

Niemniej nawet w tej strefie Polska 2, strefie lotnisk regionalnych, opłaty terminalowe będą mniejsze niż np. w Rumunii czy na Węgrzech, o Niemczech nie wspominając, gdzie będą znacznie większe.

Wśród tych państw są Niemcy, które i tak podniosły opłaty znacznie bardziej niż w Polsce, bo o 150%. Zdecydowanie nie przywoływałbym przypadku hiszpańskiego, bo w Hiszpanii agencja kontroli przestrzeni powietrznej faktycznie (Dzwonek) otrzymała wsparcie, ale nie od rządu, tylko od lotnisk. Myślę, że w Polsce lotniska nie chciałyby tak dokładać jak w Hiszpanii. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę pana posła Tadeusza Aziewicza o zabranie głosu. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Problemy finansowe służb żeglugi powietrznej wynikają z mniejszego ruchu - jak słusznie powiedział pan minister Horała - który jest skutkiem pandemii. Wysoka podwyżka opłat osłabi porty lotnicze oraz przewoźników i może skutkować dalszym zmniejszeniem liczby lotów, szczególnie że skończył się sezon i wchodzimy w kolejną fazę pandemii. Podmioty funkcjonujące na rynku lotniczym walczą o przetrwanie, nie mogą już liczyć na kolejne tarcze.

Porty lotnicze generują dużą ilość pozytywnych efektów zewnętrznych, dlatego że działają nie tylko dla pasażerów, ale także dla podmiotów, które żyją z turystyki: hotelarzy, gastronomików, taksówkarzy i wielu innych, którzy płacą podatki.

Nie do końca rozumiem, skąd ta obstrukcja, panie ministrze. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo! Mamy tutaj do czynienia z pewną. Oczywiście zgadzam się, że branża lotnicza jest w trudnej sytuacji i chcemy jej pomagać. Stąd decyzja o specjalnej dodatkowej dotacji poza innymi mechanizmami tarcz, 142 mln zł w zeszłym roku, stąd wsparcie dla narodowego przewoźnika, który dzięki temu działa, funkcjonuje, lata i ponosi różne opłaty, chociażby te na rzecz lotnisk.

Jest zagraniczny przewoźnik, prowadzi biznes na polskim rynku i ten biznes wiąże się z określonymi kosztami.

Opowieści o tym, że polscy pasażerowie w związku z tym uciekną i przeniosą się gdzieś za granicę, też włożyłbym między bajki, ponieważ np. właśnie we wspomnianych Niemczech jest znacznie większa podwyżka. Gdyby te podwyżki miały spowodować ucieczki i przenosiny pasażerów, to raczej możemy się spodziewać dużej liczby dodatkowych pasażerów, które przeniosą się do Polski z Niemiec, gdzie opłaty terminalowe są - przypominam - podwyższane o 150%, a w Polsce tylko o 70%.

Ale cieszy mnie ta deklaracja o wspieraniu sektora lotniczego. Zabrakło tego wsparcia, kiedy np. procedowaliśmy nad ustawą, która zapobiegała nadmiernemu obciążaniu portów lotniczych ze względu na podatek od nieruchomości, bo część samorządów wchodziła w pewną lukę prawną i naliczała podatek. To milionowe koszty dla portów lotniczych, które udało się ograniczyć, a opozycja wtedy była przeciw. Liczę też na wsparcie, kiedy będziemy procedować nad ustawą Prawo lotnicze, która m.in. ukróci pewną patologię w naliczaniu nienależnych odszkodowań hałasowych, co bardzo obciąża polskie porty regionalne, nieraz kwotami kilkudziesięciu, kilkuset milionów złotych. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do następnego pytania. Pan poseł Robert Obaz z klubu parlamentarnego Lewica zada pytanie w sprawie rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem kopalni węgla kamiennego Turów w Bogatyni i aktualnego stanu negocjacji ze stroną czeską. Pytanie to jest skierowanego do prezesa Rady Ministrów, w którego imieniu odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Piotr Dziadzio. Bardzo proszę pana posła Obaza o zadanie pytania. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie ulega wątpliwości, że rząd PiS zapomniał o mieszkańcach Bogatyni. Otwarcie mówią o tym mieszkańcy tzw. worka turoszowskiego. Gdyby nie sprawa kopalni, nikt z PiS nie wiedziałby nawet, gdzie Bogatynia leży, co uwiarygodnił jeden z ministrów spraw zagranicznych na posiedzeniu Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej. Nikt w rządzie nie pomyślał także, by Bogatynię zwolnić z płacenia podatku janosikowego. Skoro nie ma pieniędzy na transformację, to chociaż w ten sposób można by było przygotować grunty pod inwestycje, wyremontować drogi w regionie i dać nadzieję 22 tys. mieszkańców i ich rodzinom, których byt zależy od przemysłu wydobywczego. Czy więc rząd zwolni Bogatynię z płacenia tego podatku? Mieszkańcom należy się także rzetelna informacja odnośnie do stanu negocjacji ze stroną czeską. Biorąc pod uwagę, że od 25 maja opinia publiczna nie posiada żadnych oficjalnych informacji o stanie negocjacji z naszymi sąsiadami, a o ich przebiegu dowiadujemy się jedynie z przecieków medialnych, chcielibyśmy usłyszeć, na jakim etapie znajdują się obecnie negocjacje ze stroną czeską i czy to prawda, że pańska dyplomacja doprowadziła do impasu w rozmowach. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, zapraszam.

Szanowni Państwo! Panie Pośle! W zasadzie to dziękuję za to pytanie, które zostało zadane, bo wydaje mi się, że opinia publiczna dość dobrze jest informowana o sytuacji, która ma miejsce w Bogatyni, a związana jest z eksploatacją węgla brunatnego, a nie kamiennego, tak jak państwo piszecie tutaj w zapytaniu. Tak wiele błędów jest popełnianych w komunikacji przez niekompetentne osoby, które się wypowiadają w tym zakresie, i przekazywanych mnóstwo dziwnych, niesprawdzonych informacji, które uderzają tak naprawdę w Rzeczpospolitą, chociażby nawet ten błąd, który jest błędem merytorycznym z mojego punktu widzenia i wszystkich nas, bo mamy do czynienia nie z kopalnią węgla kamiennego, tylko z kopalnią odkrywkową węgla brunatnego. Proszę sobie to też wziąć pod uwagę. Kolejna sprawa, na którą chciałem państwu zwrócić uwagę, to to, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej przywiązuje najwyższą wagę do znalezienia możliwości polubownego zakończenia sporu z Republiką Czeską odnośnie do potencjalnych skutków działalności kopalni w Turowie. Na przestrzeni ostatnich lat utrzymywane były stałe kontakty na poziomie roboczym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w zakresie współpracy dotyczącej transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale równocześnie odbywały się regularne spotkania bilateralne ze stroną czeską. Wielokrotnie takie spotkania się odbywały, były to spotkania negocjacyjne, rozmowy, w których również brałem udział. O tym już państwa informowaliśmy tutaj, na forum Sejmu. Szanowni Państwo! To, że opinia publiczna nie posiada informacji, jest nieprawdziwa, dlatego że staramy się na bieżąco informować o wszystkich sprawach związanych z sytuacją w Turowie. Niemniej jednak jest ona sytuacją wrażliwą, bo trwają negocjacje.

Oczywiście mogę przybliżyć całą historię sytuacji związanych z Turowem, niemniej jednak chyba to nie jest miejsce ani czas, bo ten czas jest ograniczony, ale chciałbym państwu powiedzieć, że od wczoraj, od 29 września, pod przewodnictwem pana ministra Michała Kurtyki trwają rozmowy negocjacyjne. To jest 14. runda, tak jak już powiedziałem. Te rozmowy polegają na tym, że Polska przedstawiła bardzo konkretną propozycję, konkretną propozycję również finansową dla kraju libereckiego, czyli kraju sąsiadującego z Rzecząpospolitą.

Raczej czekajmy na rezultat, niż gdybajmy, co ewentualnie będzie, jaki rezultat może się pojawić. Dziękuję serdecznie. Żegnany na chwilę burzliwymi oklaskami pan minister siada i czeka na drugie pytanie. Bardzo proszę, panie pośle, drugie pytanie. Wysoka Izbo! Zupełnie nie odpowiedział pan na pierwszą część pytania dotyczącą rozwoju Bogatyni w przyszłości i możliwości zwolnienia z janosikowego. Druga rzecz. A swoją nieznajomość tematu podkreślił pan tym, że mówił pan dwukrotnie, że Kopalnia Węgla Brunatnego Turów leży w Turowie. Nie leży w Turowie, leży w Bogatyni w dzielnicy Turoszów, panie ministrze. O takich rzeczach chyba warto wiedzieć, zanim się odpowiada.

Co dalej, panie ministrze? Jakie plany przygotowaliście, żeby przygotować szkoły, samorząd, strefy ekonomiczne, żeby tam się mogło to znaleźć, żeby wybudować nowe drogi, trasy kolejowe? Co dalej z tym regionem? Dziękuję. Bardzo proszę.

Powiedziałem: Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Oczywiście, że jest w Bogatyni, to nie jest kwestionowane. Szanowni Państwo!

Koncesja, która jest obowiązującą koncesją, jest koncesją eksploatacyjną do 2044 r. Oczywiście cały obszar. Przedsiębiorca, który jest właściwy do zakończenia i zrekultywowania obszaru, jest odpowiedzialny za przygotowanie procesu zakończenia eksploatacji.

Ja o to pytałem.

Pytam, jakie pieniądze państwo przeznaczą jako rząd.

Czyli nie ma pomysłu. Pan poseł Andrzej Grzyb z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska zada pytanie w sprawie pilnej pomocy dla producentów trzody chlewnej w związku ze spadkiem cen i opłacalności produkcji spowodowanej rozszerzającym się obszarem występowania ASF. To pytanie jest skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a odpowie na nie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan minister Ryszard Bartosik. Panie pośle, bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze czy Panowie Ministrowie! Chciałbym zadać pytanie, które dotyczy sytuacji w produkcji trzody chlewnej, która jest sytuacją, jak rolnicy mówią, dramatyczną.

Bardzo wiele gospodarstw podejmuje decyzję o zamknięciu produkcji, jeżeli produkują w cyklu otwartym, a te, które produkują w cyklu zamkniętym, też redukują swoje stada mateczne.

Jakie mechanizmy zamierza uruchomić rząd, aby zatrzymać spadek produkcji oraz spadek cen? Czy rząd zamierza uruchomić interwencję na rynku, aby [[Dzwonek]] zatrzymać rujnujący gospodarstwa spadek cen i opłacalności w tych strefach?

Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam uprzejmie.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Kilka słów o działaniach pomocowych dla producentów świń. Pomoc w ramach programu obejmuje instrumenty zapewniające realizację działań związanych z bioasekuracją gospodarstw, eliminacją zjawiska najniższej ceny skupu żywca w strefach ASF, osłoną zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, odbudową pogłowia świń, wsparciem w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw. Aktualnie program jest skoncentrowany na inwestycjach w bioasekurację gospodarstw utrzymujących świnie. Trwa nabór wniosków w ramach działania 5.1.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji - do 80% - w przypadku np. utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekującej, modernizacji budynków albo formę standardowych stawek jednostkowych w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej wykonania ogrodzenia chlewni.

Producenci rolni prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF mogą ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Producenci świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, mogą również skorzystać z pomocy finansowej. Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony (Dzwonek) zakaz, i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Rząd zamierza również. Panie pośle, proszę bardzo, pytanie dodatkowe. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za tę część informacji, w której pan szeroko omówił kwestie redukcji populacji dzików, w tym monitoringu, barier i działań o charakterze prewencyjnym, ale również nowych instrumentów, które są uruchomione.

A tam są pełnowartościowe stada, które mogą być gospodarczo wykorzystane. Tam jest brak możliwości ruchu, są bardzo ograniczone możliwości sprzedaży, są ponoszone dodatkowe koszty, bo stada przerastają. Podobnie wyznaczenie stref niebieskich sprawia, że tam również występuje presja cenowa, presja na spadek cen ze strony podmiotów skupujących.

Panie ministrze, proszę bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zamierzamy uruchomić interwencję na rynku, aby zatrzymać rujnujący gospodarstwa spadek cen i opłacalności produkcji w obrębie stref niebieskich związanych z wystąpieniem ASF-u. Mechanizmy interwencyjne, które mają na celu poprawę opłacalności poprzez wzrost cen skupu, mogą być uruchamiane zgodnie z przepisami wspólnej organizacji rynków rolnych, które stosowane są jednolicie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami interwencja publiczna, jak wszyscy wiemy, w przypadku wieprzowiny nie obejmuje mechanizmów interwencyjnych. Mechanizmem rynkowym, jaki może być uruchomiony na rynku wieprzowiny, ale następuje on wyłącznie w drodze rozporządzenia Komisji Europejskiej, jest mechanizm dopłat to prywatnego przechowywania wieprzowiny. W chwili obecnej pomimo podnoszonej przez Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej dramatycznej sytuacji na rynku wieprzowiny Komisja Europejka stoi na stanowisku, że uruchomienie interwencji na rynku wieprzowiny jest niezasadne. Niestety taka jest sytuacja. Niezależnie od powyższego minister rolnictwa i rozwoju wsi wystąpił z pismem w trybie niejawnym do prezesa rady ministrów o uruchomienie zakupu mięsa wieprzowego lub wybranych wyrobów wieprzowiny na rezerwy strategiczne w ramach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Działanie będzie polegało na rekompensowaniu rolnikom kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt, zastosowaniem podwyższonych standardów. Tam są dwa warianty: dobrostan loch i dobrostan tuczników. Jeżeli chodzi o zamierzenia związane z zapowiadanym zwiększeniem dobrostanu w WPR, Komisja Europejska w strategii od pola do stołu wskazała na pilną potrzebę poprawy dobrostanu zwierząt.

Będziemy zwracać się na najbliższym posiedzeniu ministrów rolnictwa Unii Europejskiej z prośbą o uruchomienie interwencji, o której mówiłem wcześniej. Dziękuję bardzo. Czy ja mógłbym tylko poprosić pana ministra o przekazanie informacji pisemnej ze względu na obszerność tego materiału? Posłanki Barbara Bartuś oraz Joanna Borowiak zadadzą pytanie w sprawie rodzaju wsparcia udzielonego polskim hodowcom pszczół oraz planowanych działań, w tym przewidzianych środków finansowych na wspieranie ochrony pszczół i rozwoju polskiego pszczelarstwa. To pytanie jest skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a odpowie na nie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan minister Ryszard Bartosik. Bardzo proszę przedstawicielki Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o zabranie głosu. Dziękuję. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Na terenie Kancelarii Sejmu mamy pasiekę. Polski Sejm jest drugim na świecie parlamentem, który posiada własną pasiekę. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo pszczoły są potrzebne, a nawet nieodzowne w gospodarce człowieka.

Wiele gatunków roślin uprawnych do wydania plonu wymaga zapylenia przez owady. Obecnie jedynymi liczącymi się zapylaczami roślin są pszczoły utrzymywane w pasiekach. A współczesny świat stwarza tyle zagrożeń, że pszczoły pozbawione opieki człowieka nie przeżyłyby. Na szczęście w Polsce mamy wielu pszczelarzy, wielu pasjonatów, ludzi kochających pracować w pasiece.

Czasami ta pasieka przynosi zyski, czasami niestety do tej pasieki trzeba dołożyć, żeby ona przetrwała. Dlatego zwracamy się do pana ministra, bo wiemy, że jest wiele dotacji, z których mogą skorzystać pszczelarze. Są dotacje na założenie, na rozwój pasieki. Czy mogą to być tylko pszczelarze zrzeszeni w związku pszczelarskim, czy może to być każdy pszczelarz, który ma pszczoły?

Czy polski rząd będzie dalej promował pszczelarstwo? Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Budżet tegorocznego programu jest dwukrotnie wyższy w stosunku do 2015 r. i wynosi 45 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy kwota wynosiła 34 mln zł, wzrost budżetu wyniósł 32%. W ramach realizowanego aktualnie „Programu wsparcia pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022” refundowane są koszty organizacji szkoleń i konferencji pszczelarskich w wysokości 100%, zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego w wysokości 60%, zakupu środków leczniczych warrozobójczych w wysokości 90%, zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej oraz pakietów okładów pszczelich z takimi matkami w wysokości 70% oraz wykonywania analiz fizykochemicznych oraz analizy pyłkowej miodu w wysokości 100%. Po raz pierwszy uruchomiliśmy dodatkową krajową pomoc dla pszczelarzy. W roku bieżącym pszczelarze otrzymali pomoc finansową w wysokości 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Jest to pomoc o charakterze de minimis.

W tym roku ta pomoc została przez nas uruchomiona. W ramach krajowego „Planu strategicznego dla WPR na lata 2023-2027” planowana jest kontynuacja obecnie realizowanych działań w krajowym programie wsparcia pszczelarstwa oraz utrzymanie poziomu wsparcia finansowego dla sektora pszczelarstwa w wysokości 10 mln euro rocznie. Rodzaje interwencji rozszerzamy dodatkowo o wsparcie naukowo badawcze. Ponadto dopuszczamy możliwość, aby również pszczelarz mógł wnioskować o wsparcie w ramach modernizacji gospodarstw pasiecznych. Promujemy również, aby w pierwszej kolejności finansowane były wnioski o pomoc dla młodych pszczelarzy celem odmładzania sektora. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Dziękuję za udzieloną odpowiedź. Ja także, podobnie jak pani poseł Barbara Bartuś, wywodzę się z rodziny o głębokich tradycjach pszczelarskich, stąd ta tematyka jest mi niezwykle bliska. Polscy pszczelarze mogą uzyskiwać pomoc finansową na zakup pszczół i sprzętu pszczelarskiego. Pan minister mówił o tym szerokim spektrum wspierania. Natomiast chciałam zapytać pana ministra, jak przebiegają konsultacje, jakie wsparcie, jakie rozwiązania przewidziane są dla polskich pszczelarzy, dla gospodarek pasiecznych w planie strategicznym na lata 2023–2027. Ja bardzo cieszę się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pamiętają o polskich pszczelarzach. Odbieram takie sygnały, że pszczelarze doceniają to wsparcie rządu. Pamiętajmy, co (Dzwonek) powiedział Albert Einstein: Jeśli z Ziemi znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną tylko 4 lata życia. Nie ma pszczół, nie ma zapylania, nie ma roślin, nie ma zwierząt, nie ma ludzi. Poproszę, panie ministrze, o przybliżenie tego, jak przebiegają konsultacje i jakie są planowane rozwiązania. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cały czas jesteśmy w kontakcie ze środowiskiem pszczelarskim i przede wszystkim odpowiedzieliśmy na ten postulat dotyczący wsparcia, które zostało udzielone w ostatnim czasie, kiedy to pszczelarze otrzymali pomoc finansową w wysokości 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej i to było wprost odpowiedzią na postulaty pszczelarzy. Jeśli chodzi o krajowy plan strategiczny, to również jesteśmy w kontakcie z sektorem pszczelarskim. Pszczelarze zgłaszali i zgłaszają swoje uwagi i chcemy na to przeznaczyć 10 mln euro rocznie.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Joanna Jaśkowiak i Aleksander Miszalski z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska zadadzą pytanie w sprawie wysokiej inflacji oraz drastycznych podwyżek cen prądu i gazu. To pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów, w imieniu którego, i z jego upoważnienia, odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Piotr Dziadzio. Bardzo proszę panią poseł Joannę Jaśkowiak o zadanie pytania.

Trzeba włożyć legitymację i nacisnąć albo podejść tutaj. Zapraszamy. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Ostatnie pana publiczne wystąpienia przy okazji promowania Polskiego Ładu i podkreślanie, jak to bardzo dobrze żyje się Polkom i Polakom, nijak mają się do rzeczywistości. Lawinowo rosnące ceny prądu i gazu pokazują, że Polska za pana rządów staje się faktycznie państwem z tektury, jak to mawiała pana poprzedniczka. Skoro mamy tak wspaniałą koniunkturę, miliardy złotych w państwowej kasie, o których często pan mówi, to dlaczego za chwilę, gdy nadejdzie zima, Polki i Polacy będę sięgać jeszcze głębiej do portfeli, by nie musieć spędzać czasu przy zakręconych grzejnikach, by mogli kupić chleb, który drożeje na skutek wysokiej inflacji, podwyżek cen prądu, i by w końcu mogli ugotować na kuchence gazowej obiad dla rodziny. Rozhulana inflacja pozwala panu manipulować budżetem państwa. Stanowi natomiast wielkie zagrożenie dla stabilności ekonomicznej państwa. Panie Premierze! Co zamierza zrobić pana rząd, by Polki i Polacy nie odczuli wzrostu cen prądu i gazu? Kiedy w końcu zareaguje pan w sposób, który pozwoli spowolnić inflację?

Proszę państwa, tu zaszła zmiana i poprosimy o wypowiedź pana ministra Piotra Patkowskiego. Bardzo proszę. Miałem inną informację, panie ministrze, przepraszam za nieporozumienie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie dotyczące inflacji, oczywiście warto rozpocząć od takiego dość już oczywistego stwierdzenia, ale zawsze dobrze jest przypominać, że inflacja często ma w odczuciu powszechnym, społecznym o wiele silniejszy wymiar, niż na to wskazują czynniki makroekonomiczne. I oczywiście w pełni rząd musi te odczucia społeczne szanować i respektować. Natomiast też od pewnych porównań makroekonomicznych nie da się uciec i warto do nich przejść.

W tym momencie głównym zadaniem czy to banku centralnego, czy w zakresie polityki rządu, czy tak naprawdę wszystkich podmiotów sceny publicznej jest dość rzetelne i realne informowanie o rzeczywistych rozmiarach obecnej inflacji. Warto także zwrócić uwagę na przyczyny obecnych odczytów inflacyjnych.

To przez kilka ostatnich lat potęgowało czy stopowało wzrosty cen ropy.

Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żeby, po pierwsze, wskazać, że dużo czynników inflacyjnych jest poza kontrolą rządu i tak naprawdę są to czynniki światowe, po drugie, zwrócić uwagę na to, że to jest trend ogólnoświatowy związany także z pewnymi kwestiami, na które nie ma wpływu, natomiast warto zauważyć, że wiele z tych państw nie reaguje w sposób drastyczny, ograniczając tę inflację - Chiny, Stany Zjednoczone, Niemcy.

Warto także zwrócić uwagę na pewien kontekst historyczny.

Bardzo podobne do tych, które występują teraz: przede wszystkim wysokie ceny surowców rolnych i energetycznych na rynkach międzynarodowych, znaczna deprecjacja złotego związana głównie z istotnym pogorszeniem nastrojów na globalnych rynkach finansowych i - uwaga - znaczna podwyżka stawek VAT w roku 2011. Ta inflacja utrzymywała się przez kilkanaście miesięcy, natomiast w ciągu 4 lat przerodziła się w deflację, która jest długookresowo o wiele gorszym stanem dla gospodarki niż inflacja. Dlaczego o tym mówię?

Warto zwrócić uwagę, że obecna inflacja nie ma znamion stagflacji, która jest chyba najgorszym możliwym zjawiskiem, jakie może wystąpić, a potwierdza to obecny niski odczyt dotyczący wskaźnika bezrobocia, a także realny wzrost pensji, który przewyższa inflację. Zostało mi pół minuty. Jakie można podjąć działania w tym celu?

Trzecim działaniem są pewne osłonowe rozwiązania dla grup najuboższych, m.in. najuboższych energetycznie, ale o tym być może powie pan minister Dziadzio w drugiej części. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Eksperci prognozują, że nawet może być paręnaście procent w 2022 r.

Manipulowanie prognozami w tym wypadku nic nie da, ponieważ wzrost cen ludzie odczuwają i on wywołuje presję (Dzwonek) na wzrost wynagrodzeń. Pytam konkretnie: Co chcecie zrobić, żeby zatrzymać ten trend? W jaki sposób chcecie walczyć z inflacją, jeżeli nie znacie nawet dynamiki wzrostu tych cen? Panie ministrze, bardzo proszę o odpowiedź. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie jest to moja kompetencja, a każda wypowiedź w tym zakresie mogłaby być bardzo nerwowo odczytana przez rynki finansowe.

On mieści się w średniookresowych prognozach międzynarodowych instytucji finansowych. Na przyszły rok jest to 3,3%. To również mieści się w widełkach prognoz instytucji finansowych, bo wszystkie instytucje wskazują, że ta inflacja rok do roku będzie spadała. Jeśli chodzi o działania rządu - pewnie nie wystarczy na to czasu - to pan Dziadzio razem z panem ministrem Kurtyką przygotowują rozwiązania osłonowe dla grup ubogich energetycznie, bo jak wspomniałem, w tym momencie to ceny energii są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost inflacji. Warto też zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, mechanizm luzowania ilościowego w jakimś stopniu, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, przyczynia się do wzrostu odczytów inflacyjnych. Stąd Polska nie zapowiada wprowadzenia taperingu, ale od 9 miesięcy go stosuje jako jedno z pierwszych państw Unii Europejskiej czy w ogóle tych, którzy stosowali mechanizm luzowania ilościowego. Jako pierwsi zastosowaliśmy mechanizm taperingu.

Natomiast jak odpowiadałem przy pierwszej części pytania, obecna luka produktowa nie wynika ze strukturalnych niedomagań podażowych gospodarki, tylko z chwilowo zaburzonych łańcuchów dostaw i czynników geopolitycznych. Uzależnianie (Dzwonek) ograniczenia działalności inwestycyjnej państwa od chwilowych czynników wywołujących lukę produktową byłoby najgorszą rzeczą, jaką można zrobić dla gospodarki wychodzącej z kryzysu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Lidia Burzyńska oraz Mariusz Trepka będą zadawali pytanie w sprawie ogólnej kwoty dofinansowania przekazanej w tym roku w ramach programów „Senior+” oraz „Aktywni+” w skali całego kraju. Pytanie to jest skierowane do ministra rodziny i polityki społecznej, w którego imieniu odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pan minister Stanisław Szwed. Bardzo proszę panią poseł Lidię Burzyńską z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o zadanie pytania. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Najważniejsze w działaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości jest to, że jesteśmy po prostu wiarygodni, że nie rozkładamy rąk, mówiąc: pieniędzy nie ma i nie będzie, tylko wprowadzamy rozwiązania prowadzące do tego, żeby osoby na jesieni swego życia były piękną częścią naszego społeczeństwa, nie tylko ze względu na ich wiedzę, doświadczenie, ale również ze względu na zaopiekowanie się nimi nie tylko przez osoby bliskie, ale również przez państwo. Programów skierowanych do seniorów rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje wiele - to m.in. trzynasta emerytura, w tym roku czternasta, „Opieka 75+”, „Leki 75+” - ale filarami tej polityki są takie programy jak „Senior+”, „Aktywni+”

W związku z prowadzeniem takiej polityki, nakierowanej na wielopokoleniową łączność, która jest najpiękniejszym sposobem realizowania polityki rodzinnej, bardzo proszę o odpowiedź, jaka była ogólna kwota dofinansowania przekazana w tym roku w ramach programów „Senior+” oraz „Aktywni+” w skali całego kraju. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, panie ministrze.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie dotyczące wsparcia dla naszych seniorów. Oczywiście to wsparcie jest bardzo szerokie, o czym mówiła też pani poseł. Przecież mówimy o wsparciu materialnym, o już wspominanej trzynastej emeryturze, w tym roku czternastej emeryturze, ale też o waloryzacji, która była waloryzacją kwotową, procentową, była wsparciem dla naszych seniorów.

To jest program skierowany do samorządów i dotyczy tworzenia dziennych domów seniora i klubów seniora.

Program „Aktywni+”, który jest skierowany do organizacji pozarządowych, też się cieszy dużym uznaniem, dużą popularnością.

I to są te jednostki, które funkcjonują.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ten program skierujemy do samorządów.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie ministrze, bardzo dziękuję za te programy, które rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi, bo to świadczy właśnie o docenieniu naszych seniorów za to, że po prostu pracowali całe życie dla Polski, o tym, że w tej chwili pamiętamy o nich.

Bardzo dziękuję. Zapraszam pana ministra. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję za te dodatkowe pytania.

W województwie łódzkim utworzono dziewięć nowych placówek, a 19 placówek otrzymało dofinansowane na kwotę ponad 2400 tys. zł. W województwie kujawsko-pomorskim utworzonych zostało 14 nowych placówek oraz 17 placówek otrzymało dofinansowanie na kwotę ponad 4200 tys. zł.

Jeśli chodzi o dwa dodatkowe pytania.

W tej chwili ponad 71 tys. kobiet i ponad 200 ojców z tego programu korzysta na łączną kwotę ponad 880 mln zł. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ono zapewnia właśnie tym osobom, które nie były w stanie wypracować sobie odpowiedniego stażu ze względu na wychowanie dzieci, pozostawanie w domu, to, że mają dzisiaj możliwość otrzymywania minimalnej emerytury. Ponad 71 tys. osób ma w tej chwili minimalną emeryturę z tego tytułu, czyli z programu „Mama 4+”

Dzisiaj granica, która dopuszcza otrzymanie świadczenia, to jest kwota 1772 zł.

Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska zadadzą pytanie w sprawie nepotyzmu i kumoterstwa związanego z kształtowaniem składów zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych oraz braku działań naprawczych mających zatrzymać masową skalę tego patologicznego zjawiska. Pytanie to zostało skierowane do prezesa Rady Ministrów, który upoważnił podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana ministra Andrzeja Śliwkę do odpowiedzi. Zapraszam pana posła Michała Szczerbę. Proszę bardzo, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam wrażenie, że przed tym pytaniem pan marszałek Czarzasty powinien puścić muzykę Ennio Morricone z „Ojca chrzestnego”, bo będziemy, szanowni państwo, pytać o mafię, o polityczną mafię, którą mogliśmy dostrzec po wielkim dziennikarskim śledztwie trzech redakcji, 50 dziennikarzy, którzy ujawnili 900 tłustych kotów w spółkach Skarbu Państwa, ściśle powiązanych albo rodzinnie, albo poprzez związki z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Dziwię się, że jest pan wiceminister, dziwię się, że nie ma premiera, który jest ojcem chrzestnym tej ekipy. To, co się dzieje w państwie PiS, to jest niebywały skandal. To już nie jest nepotyzm ani klientelizm. Klientelizm, używam tego słowa, bo wiedzieliśmy również z maili ścisłą korelację między nazwiskami osób wpłacających na kampanię szefa KPRM-u a później ich awansami w spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych. To już nie jest nepotyzm ani klientelizm, państwo po prostu ukradliście państwo. To polityczny kolonializm, tak to trzeba dzisiaj nazwać. Ta skala, można powiedzieć w putinowskim stylu, z której już się nie daje zawrócić. Pan dostał konkretne zadanie od premiera, od prezesa Kaczyńskiego. Jak ta uchwała kongresu PiS jest realizowana? Ile tłustych kotów panu się udało ustalić, bo dziennikarze ustalili ich 900? Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W praktyce to wygląda tak: premier Morawiecki powołuje prezesa (Dzwonek) LOT-u. W czasie pandemii przekazuje nawet 3 mld na ratowanie LOT-u, więc już na pensje zarządu jest, a dostają niemało, bo prawie ponad 2,5 mln, a zwykłe stewardesy, piloci są wyrzucani na bruk. Dzisiaj trzeba brać załogę z Węgier. Tak wygląda patologia państwa PiS. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo!

Postaram się systemowo wyjaśnić, jak ten proces wygląda.

Jeśli przedmiotowa legislacja nie została zauważona, to służę wyjaśnieniem. Zacznijmy od rad nadzorczych. Kandydatem Skarbu Państwa do tego organu może być jedynie osoba, która posiada pozytywną opinię rady do spraw spółek. W skład rady wchodzą osoby z ugruntowanym dorobkiem zawodowym, urzędniczym, jak i naukowym z różnych dziedzin, są to specjaliści z zakresu prawa, finansów, ekonomii. Przed reformą decyzje o doborze kandydatów do rady nadzorczej podejmował minister skarbu. Kandydat musi spełniać również szereg ustawowych wymogów. Musi mieć odpowiednią wiedzę, doświadczenie, wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letni staż pracy.

Poza wymogami formalnymi Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa weryfikuje również merytoryczne przygotowanie kandydata na członka rady nadzorczej. Dlatego dobór kandydatów dokonywany jest spośród osób, które posiadają wysokie kwalifikacje oraz merytoryczną wiedzę potrzebną w danej radzie nadzorczej konkretnej spółki. Jednak to nie jest koniec procesu. Ostateczna decyzja dotycząca powołania danej osoby do rady nadzorczej zapada w zdecydowanej większości przypadków na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy danej spółki. Zwracam uwagę, że w wielu spółkach, szczególnie tych najważniejszych, tych największych, Skarb Państwa posiada udział mniejszy niż 50%. Często jest to pułap wynikający z ustawy o ofercie publicznej, czyli mówię o pułapie do 33%. Oznacza to, że na walnym zgromadzeniu znaczenie ma również głos akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa, którzy mogą nie zgodzić się na przedstawioną kandydaturę do rady nadzorczej. Wyjątkiem są oczywiście uprawnienia statutowe Skarbu Państwa w niektórych spółkach, które często wpisywane były podczas ich prywatyzacji, przed 2016 r. W takich sytuacjach powołanie może nastąpić oświadczeniem reprezentanta Skarbu Państwa, w niektórych sytuacjach także bez uchwały walnego zgromadzenia. Co do zarządów. Zgodnie z przywołaną już przeze mnie ustawą o zasadach zarządzania mieniem z 2016 r. ta kwestia została uporządkowana. Członkowie zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa powoływani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Takie postępowanie prowadzi rada nadzorcza, która sprawdza i ocenia kwalifikacje kandydatów oraz wyłania najlepszego z nich. Dodatkowo w sektorze finansowym część członków zarządu musi uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego. Ex ante chodzi o prezesa i wiceprezesa do spraw ryzyka. Jeżeli mówimy o procedurze ex post, ona dotyczy wszystkich pozostałych członków zarządu. Warto także wskazać, że zgodnie z przepisami ani do rady nadzorczej, ani do zarządu nie można wybrać osób, które są asystentami posłów czy senatorów albo wchodzą w skład organów partyjnych lub pracują dla partii politycznych. Na samym końcu chciałbym również zwrócić uwagę, że wykaz wszystkich członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa w nadzorze ministra aktywów państwowych jest dostępny publicznie. Mamy zatem pełną transparentność i merytoryczny dobór kadr. Takie standardy funkcjonują teraz. Ale mogę powiedzieć, że nie spoczywamy na laurach, ponieważ do Sejmu właśnie wpłynął projekt opracowany w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zawierający kompleksową, największą od 20 lat reformę prawa handlowego. Jednym z dwóch filarów proponowanych zmian jest zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze. Nie dotyczy to rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, ale wszystkich podmiotów. Dajemy tym radom nowe kompetencje, ale idzie za nimi również większa odpowiedzialność. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Dariusz Joński. Chciałem panu posłowi Michałowi Szczerbie powiedzieć, że zafascynowała mnie informacja, że Ennio Morricone napisał muzykę do „Ojca chrzestnego” Bardzo proszę, panie pośle. Tak? Super. Człowiek się uczy całe życie. Wysoka Izbo! Otóż jestem rozczarowany. Pytanie było proste, panie ministrze: Ile pan ustalił, ile pan wytropił tłustych kotów, krótko mówiąc, tych wszystkich nazwisk polityków, działaczy Prawa i Sprawiedliwości, członków ich rodzin? Tymczasem mamy do czynienia z ośmiornicą, której macki dotykają każdej instytucji, każdego miejsca, gdzie rządzi PiS. A tam działacze, często bez wykształcenia, doświadczenia, z pensjami wielomilionowymi - kosztem fachowców. Podam teraz panu drugi przykład, Poczty Polskiej. Akurat prezes jest teraz z namaszczenia ministra Błaszczaka. Ale czy pan wie, że połowa pracowników Poczty Polskiej jest na minimalnym wynagrodzeniu, [[Dzwonek]] bo nie ma pieniędzy, bo wydaliście 70 mln w piach i zabraliście tym ludziom nawet pieniądze na premie? Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie pośle, jeśli chciałbym być złośliwy, a nie jestem, to przypomniałbym kazus pewnego posła, który w 2015 r. przegrał elekcję i bez żadnego doświadczenia i wiedzy został wiceprezesem miejskiego aquaparku. Rozumiem, że wtedy to był przykład fachowości i kompetencji. Być może państwo życzylibyście sobie, żeby w radach nadzorczych i zarządach zasiadali ludzie o poglądach zbliżonych do poglądów pana premiera Rostowskiego czy pana ministra Sienkiewicza, którzy cały państwowy majątek chcieliby sprywatyzować. Jednak nasza filozofia - Ministerstwa Aktywów Państwowych, rządu jest zgoła inna. Zamiast sprzedawać aktywa państwowe, wolimy je pomnażać. Do pracy angażujemy menedżerów, którzy to potrafią. Od momentu powołania Ministerstwa Aktywów Państwowych, mówię o czasie od listopada 2019 r. do września br., wartość notowanych na giełdzie spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa wzrosła o prawie 30 mld. Udziały samego Skarbu Państwa zyskały w tym okresie na wartości ponad 11,5 mld. Dla porównania WIG wzrósł w tym czasie o 5,4%. Ogółem blisko 70% spółek Skarbu Państwa notowanych na warszawskim parkiecie poprawiło notowania w omawianym okresie. To jest właśnie dobre zarządzanie i umiejętne reagowanie na różne czynniki makroekonomiczne, takie jak chociażby kryzys spowodowany pandemią koronawirusa.

Tu warto wskazać, że od 2017 r. nakłady inwestycyjne spółek notowanych na giełdzie będących pod kontrolą Skarbu Państwa systematycznie rosły. W pandemicznym roku 2020 inwestycje tych spółek wzrosły do rekordowego poziomu 45 mld. To jest wzrost, panie pośle, blisko o 20%, podczas gdy nakłady pozostałych przedsiębiorstw, głównie prywatnych, dotknął spadek o 13%. Spółki Skarbu Państwa były zatem motorem napędowym polskiej gospodarki w tym trudnym czasie. Jeżeli aktualne wyniki, rekordowe wydatki CAPEX, ale przede wszystkim zaufanie inwestorów - bo proszę mieć świadomość tego, że ci inwestorzy alokują swoje prywatne środki w akcje Skarbu Państwa, przepraszam, w akcje spółek Skarbu Państwa - nie są wystarczającym dowodem, że podmioty z domeny Skarbu Państwa są dobrze zarządzane przez kompetentnych menedżerów, merytorycznych i sumiennych członków rad nadzorczych, to znaczy to tyle, że merytoryczne argumenty do pytających nie trafiają. A szkoda. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, przechodzimy do następnego pytania.

Panowie posłowie Waldemar Andzel, Marek Polak i Jarosław Krajewski zadadzą pytanie w sprawie systemu dozoru elektronicznego. To pytanie jest skierowane do ministra sprawiedliwości. Odpowiadać będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan minister Michał Woś. Panu ministrowi Andrzejowi Śliwce serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości polski system dozoru elektronicznego jest najnowocześniejszy w Europie i stale się rozwija. Proszę o przedstawienie najistotniejszych zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu systemu dozoru elektronicznego, a także wskazanie ilości odbytych kar w tym systemie przez osadzonych. Jaka jest efektywność kary w systemie dozoru elektronicznego, ilu skazanych zostaje osadzonych w zakładach penitencjarnych. Czy planowane są jakieś dalsze zmiany w przepisach dotyczących systemu dozoru elektronicznego? Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Marek Polak. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Otóż obecnie decyzji o odbyciu kary w systemie dozoru elektronicznego nie podejmuje sąd karny wymierzający karę, a podejmuje ją sąd penitencjarny już na etapie wykonywania orzeczenia. Chciałbym zapytać, z czego to wynika i czy nie byłoby lepiej, a być może nawet sprawniej i szybciej, gdyby robił to sąd wydający wyrok, który od początku do końca zna już całą sprawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, zapraszam. Szybkie pytania. Pan minister Michał Woś. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Polskie e-więzienie konkuruje w różnych miesiącach z Francją, ale można powiedzieć, że jest największym elektronicznym więzieniem w Europie, a być może także na świecie.

Kiedy objęliśmy władzę, już 11 marca 2016 r. nastąpiła nowelizacja Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, gdzie przywróciliśmy szeroką możliwość stosowania systemu dozoru elektronicznego, który ma bardzo wiele pożytecznych, pozytywnych cech. Pozwala skazanym za łagodniejsze przestępstwa odbywać karę właśnie w dozorze elektronicznym, podejmować dalej pracę, realizować chociażby swoje zobowiązania alimentacyjne, nie być oderwanym jednoznacznie od tego środowiska czy czasem nie powodować tego, że trafiają oni do zakładów karnych czy aresztów śledczych, skąd, bywa i tak, wychodzą bardziej zdemoralizowani. Oczywiście każdy taki przypadek odbieramy jako państwo jako porażkę i robimy wszystko, żeby tak nie było. Żeby trafić do systemu dozoru elektronicznego, rzeczywiście jest potrzebna decyzja sądu penitencjarnego, po - i to jest niezwykle istotne - nie tylko zbadaniu warunków technicznych, co oczywiste, ale przede wszystkim po zbadaniu warunków rodzinnych, lokalowych, tego, czy rodzina się na to godzi i czy miejsce do objęcia systemem dozoru elektronicznego jest odpowiednie. Szanowni Państwo! Po tym przywróceniu w 2016 r. możliwości odbywania kary, a nie tylko ograniczenia wolności, w systemie - czyli już po tych złych zmianach z lipca 2015 r. i po załamaniu systemu - kolejna reforma została przeprowadzona ustawą, która weszła w życie 1 czerwca 2018 r. Wówczas usprawniliśmy działanie systemu dozoru elektronicznego w ten sposób, że obowiązków związanych z realizacją tej kary nie wykonuje prywatna firma, ale są one nałożone na państwo. To Służba Więzienna, mając specjalne Biuro Dozoru Elektronicznego pod bardzo sprawnym dowództwem pana gen. Nasiłowskiego, któremu serdecznie dziękuję za te lata poświęcone rozwojowi tego systemu, i całemu zespołowi oczywiście, doprowadziła do tego przede wszystkim - statystyki statystykami, ale wszystkie statystyki okazały się lepsze - że ci ludzie, którzy trafiają do systemu dozoru elektronicznego, odbywając swoją karę, nie powracają do przestępczości. Jednoznacznie statystyki pokazują, że w ramach systemu dozoru elektronicznego powrotność do przestępczości jest dużo, dużo niższa niż przy wykonywaniu zbliżonego wymiaru kary w zakładach karnych. Kolejne rozszerzenie systemu dozoru elektronicznego nastąpiło przy ustawach COVID-owych w marcu 2020 r. Wówczas zdecydowaliśmy się rozszerzyć możliwość stosowania SDE - stosować go nie tylko w przypadkach kar do roku pozbawienia wolności, ale do roku i 6 miesięcy, do półtora roku pozbawienia wolności. I, szanowni państwo, teraz konkretne dane.

Obecnie najnowsze dane pokazują, że mamy w nim ok. 7 tys. osób, w zależności od dnia, bo oczywiście codziennie są instalacje i deinstalacje. Czyli tylko w ciągu ostatniego roku nastąpił wzrost wykorzystania systemu dozoru elektronicznego o 49% i to jest rzeczywiście duży sukces, z którego resort sprawiedliwości jest dumny. Mianowicie system dozoru elektronicznego jest po prostu tańszy, 5-krotnie tańszy niż wykonywanie kary pozbawienia wolności w tradycyjnym modelu.

Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Pan poseł Jarosław Krajewski, pytanie dodatkowe. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, system dozoru elektronicznego to najnowocześniejszy, nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności, ale również najtańszy sposób odbywania kary.

W związku z powyższym mam dodatkowe pytanie do pana ministra: Ile osób objętych systemem dozoru elektronicznego w 2021 r. naruszyło warunki odbywania kary i ile przeprowadzono profilaktycznych wizyt kontrolnych w miejscu pobytu skazanych w 2021 r. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo! Rzeczywiście jest to dużo lepszy, skuteczniejszy system niż model tradycyjny. Ale też chcę powiedzieć, dlaczego mówimy o tym, że jest to największe więzienie w Europie.

To pokazuje, że rzeczywiście działania wdrożone przez rząd Zjednoczonej Prawicy przynoszą odpowiednie efekty, odpowiednie skutki. Planujemy też dalsze reformy i dalsze zmiany, rozszerzenie systemu dozoru elektronicznego. Chodzi o to, żeby tym modelem, tym skutecznym sposobem wykonywania, odbywania kary objąć jeszcze większą liczbę osób z korzyścią dla państwa. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Jarosław Gonciarz, Wojciech Szarama i Jerzy Bielecki z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadadzą pytanie w sprawie dostępności napojów energetycznych. A ja panu ministrowi Wosiowi serdecznie dziękuję za przybycie. Proszę bardzo, głos zabierze pan poseł Jarosław Gonciarz. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Z roku na rok coraz bardziej zauważalne jest spożycie napojów energetyzujących niestety wśród dzieci i młodzieży. Substancje zawarte w takich napojach mogą być bardzo szkodliwe w przypadku przyswojenia większych ilości. Jednymi z najczęściej pojawiających się problemów są nadmierne pobudzenie skutkujące brakiem skupienia, bezsenność oraz bóle głowy. Jednak zdecydowanie gorszymi powikłaniami wywołanymi zawartymi substancjami są zaburzenia rytmu serca, martwica wątroby, zaburzenia neurologiczne. Zwracam się zatem do pana ministra z pytaniem: Czy rozważa się wprowadzenie ograniczeń wiekowych związanych ze sprzedażą omówionych produktów na wzór innych państw europejskich, aby zadbać o zdrowie dzieci? Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ja chciałbym zapytać, czy ministerstwo monitoruje, co znajduje się w napojach energetycznych, czy monitoruje, które energetyki uzależniają najbardziej, jakie są objawy uzależnień od napojów energetycznych i jakie są skutki picia napojów energetycznych. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam uprzejmie.

Będziecie panowie zadawali dodatkowe pytanie? Proszę bardzo, panie ministrze. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Spożywanie napojów energetycznych oczywiście jest dużym problemem, zaczyna się robić dużym problemem, bo widzimy, że młodzież coraz chętniej po te napoje sięga.

Badanie wskazuje na możliwe niekorzystne tendencje w przyszłości, ponieważ spożycie tych napojów u coraz młodszych respondentów zdecydowanie rośnie. Wspomaganie się napojami energetyzującymi w czasie nauki jest coraz powszechniejsze, a to ze względu na skład, głównie ze względu na zawartość kofeiny i tauryny, a nie są to przecież produkty obojętne dla zdrowia. Kofeina oraz tauryna stanowią najczęstsze dodatki do napojów energetyzujących.

To m.in. liście krzewu herbacianego, ostrokrzewu paragwajskiego mate, nasiona kawy, kakao i wielu innych roślin. W napojach energetyzujących najczęściej stosowana jest kofeina razem z tauryną jako składnik, który ma korzystny wpływ na wytrzymałość, koncentrację, czas reakcji, szybkość i samopoczucie. Kwestie legislacyjne. Zgodnie z normami, które są przekazane przez prawo europejskie dotyczące prawa żywnościowego, żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka. Warto podkreślić, że zgodnie z tymi aktami europejskimi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji ponosi właściciel zakładu będący podmiotem działającym na rynku spożywczym. W przepisach prawa żywnościowego nie ma definicji napojów energetyzujących.

Wysoka zawartość kofeiny w tych produktach działa niekorzystnie właśnie na młodzież, na dzieci, na kobiety w ciąży, także na matki karmiące, dlatego na tych napojach takie hasła, takie ostrzeżenia na etykiecie są umieszczane. Także minister zdrowia podejmuje szereg działań, aby ograniczyć spożycie napojów energetyzujących u dzieci i młodzieży.

Ale nie tylko to. W ubiegłym roku wprowadziliśmy także tzw. opłatę cukrową. To opłata, która dotyczy napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących, ale także kofeiny oraz tauryny.

Tak, oczywiście. Są pewne normy, które nie mogą być przekraczane, i to jest pod stałym monitoringiem.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Jarosław Gonciarz. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dużą rolę w uświadamianiu nieletnim szkodliwości energetyków odgrywa najbliższe środowisko, w tym oczywiście rodzice, opiekunowie. Pragnę zapytać, czy ministerstwo zamierza zachęcać szkoły, placówki oświatowe do podjęcia wspólnych starań w uświadamianiu najmłodszym i ich opiekunom skali szkodliwości tego zjawiska. Dziękuję. Proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!

Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do ostatniego pytania. Posłowie Józefa Szczurek-Żelazko, Anna Pieczarka oraz Urszula Rusecka z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadadzą pytanie w sprawie programu budowy domów bez zbędnych procedur administracyjnych i innych programów wspierających rodziny w uzyskaniu własnego mieszkania lub domu. To pytanie jest skierowane do ministra rozwoju i technologii, a odpowie na nie sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pan minister Piotr Uściński, którego witamy razem z ekipą. Zaczynamy od pytania. Bardzo proszę, pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko. Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 r. konsekwentnie realizuje strategię wspierania polskich rodzin. Na dowód można podać wiele ustaw, które zostały wprowadzone i które mają na celu wspieranie rodzin pod względem finansowym.

Tutaj chciałabym podać przykład samorządu gminy Zakliczyn w województwie małopolskim, która z dużym powodzeniem realizuje wielorodzinne budownictwo.

Mam pytanie do pana ministra. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwaliliśmy ustawę, która daje możliwość budowy domów jednorodzinnych bez zbędnych formalności.

Bardzo proszę, druga część pytania, pani poseł Anna Pieczarka. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje dodatkowe pytanie spowodowane jest bardzo dużym zainteresowaniem, które osobiście odbieram, mieszkańców południowej Polski, skąd pochodzę.

Stąd moje pytania, panie ministrze. Kiedy wejdzie w życie możliwość budowy domów bez zezwolenia? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana ministra. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie.

Gmina Zakliczyn buduje już 30 mieszkań komunalnych, korzysta przy tym z bezzwrotnego wsparcia dla gmin z Funduszu Dopłat. Następna inicjatywa, w której gmina bierze udział, to przystąpienie w sierpniu do założonego niedawno SIM Małopolska. Dostała w tym zakresie wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł i wraz z 16 innymi gminami będzie budowała w ramach SIM. Chodzi o budownictwo społeczne, czyli budownictwo, w którym będzie po prostu tani czynsz i rodziny z Zakliczyna znajdą swoje miejsce do życia. Druga część pytania dotyczyła ustawy o domkach 70-metrowych. Chodzi o takie domy, które będą miały w podstawie 70 m zabudowy, maksymalnie dwie kondygnacje. Muszą być zaprojektowane tak, aby nie oddziaływały na działki sąsiednie, czyli wszelkie przepisy muszą być tak spełnione, żeby tam nie było oddziaływania, żeby sąsiedzi nie musieli być stronami w postępowaniu, żeby to była po prostu łatwiejsza procedura. Muszą być zaprojektowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania. Jeśli miejscowego planu zagospodarowania nie ma, to muszą być badane warunki zabudowy, tak jak do tej pory w każdym innym przypadku.

Taki termin wpisaliśmy do ustawy.

Do starostwa będzie składany oczywiście projekt architektoniczno-budowlany. Ten projekt będzie można pobrać za darmo ze strony GUNB-u.

Wystarczy go zaadaptować, wrysować w plan zagospodarowania działki, to zrobi projektant, i taki projekt będzie można zgłaszać.

Senat ma kilka tygodni. Myślę, że na przełomie roku ta ustawa wejdzie w życie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zapewnienie mieszkania jest jednym z bardzo ważnych elementów stabilizacji rodziny. Niewątpliwie ta ustawa wpisuje się w szeroką politykę prorodzinną realizowaną przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Moje pytanie do pana ministra. Żeby ten program się udał, muszą być plany zagospodarowania w gminach, musi być współpraca z samorządami. Co w przypadku nieposiadania przez gminy planów zagospodarowania przestrzennego? Bardzo dziękuję. Zapraszam, panie ministrze. Wysoka Izbo! Jeśli plan miejscowy jest, to oczywiście budowa musi być zgodna z planem. W tych warunkach zabudowy analizują obszar dookoła inwestycji, sprawdzają, jaka zabudowa jest w pobliżu. Obecne przepisy mówią, że w odległości nie mniejszej niż 50 m od terenu inwestycji bądź trzy długości działki wzdłuż drogi, przy której znajduje się ta działka inwestycyjna.

Jeśli w tym obszarze jest jakaś zabudowa, to do tej zabudowy będą dostosowane te warunki techniczne, które będą wydane. Jeśli nie będzie zabudowy, nie będzie możliwości budowy takiego budynku. Nie możemy dopuszczać do nieładu architektonicznego. To ograniczenie do 200 m spowoduje, że nie będzie można budować tych budynków w szczerym polu, tylko będą mogły być realizowane w pobliżu zabudowy, jeśli nie ma miejscowego planu, tak jak podkreślam. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie poziomu realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w oparciu o rozwiązania zaproponowane w Polskim Ładzie, o której przedstawienie wnosi Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. I tego na pewno będziemy się trzymać. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Wojciecha Zuborowskiego. Pana posła Zubowskiego. Przejęzyczyłem się, przykro mi. Przepraszam serdecznie. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Art. 75 konstytucji mówi, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania, i że ochronę praw lokatorów określa ustawa. Warto dowiedzieć się, jak realizacja tego zadania przebiegała w ostatnich latach i czego w sprawie zaspokojenia jednej z najważniejszych potrzeb obywateli mogą spodziewać się Polacy. Posiadanie mieszkania nie tylko jest jednym z warunków potrzebnych do założenia rodziny, wychowywania dzieci. Sytuacja na rynku mieszkaniowym pokazuje też stopień zamożności społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Pozwolę sobie przytoczyć kilka danych, które pozwolą porównać lata rządów naszych poprzedników, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, z rządami Zjednoczonej Prawicy. Nie został uruchomiony żaden program budownictwa społecznego.

Zadań tych nie da się zrealizować bez współpracy z samorządami.

O 15 punktów procentowych zwiększyło się wsparcie na tworzenie lokali na wynajem realizowanych przez inwestora innego niż gmina. Pomoc dla kredytobiorców czy środki przekazywane samorządom w ramach Polskiego Ładu na rozwój infrastruktury i konieczną przebudowę mieszkań to działania, których efekty widać chociażby we wskaźnikach.

Co bardzo ważne, regularnie zmniejsza się udział wydatków na utrzymanie mieszkania w wydatkach gospodarstw domowych, wskaźnik deprywacji mieszkaniowej, tj. liczba mieszkań, które tak delikatnie mówiąc, wymagają remontu - dotyczy to najczęściej osób najgorzej sytuowanych - i współczynnik przeludnienia. Widać więc wyraźnie, że prowadzona w ostatnich latach polityka nastawiona na mieszkańców, a nie na banki i deweloperów, daje efekty. Nie znaczy to jednak, że potrzeb już nie ma.

Dziękuję serdecznie panu posłowi. Proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pana Piotra Uścińskiego. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Mam przyjemność przedstawić dzisiaj informację rządu w sprawie poziomu realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w oparciu o rozwiązania zaproponowane w Polskim Ładzie. Po pierwsze, jakie były te cele Narodowego Programu Mieszkaniowego, o które państwo pytacie?

Instrumenty tej polityki na bieżąco dostosowywane są do sytuacji rynkowej, jednak cele programu wyznaczone w perspektywie do 2030 r. pozostają niezmienne i wyznaczają ramy makroekonomiczne polityki społecznej, polityki mieszkaniowej w Polsce. Główne cele określone w Narodowym Programie Mieszkaniowym są trzy. Pierwszy to zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Drugi cel określony w 2016 r. to zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową. Trzeci cel to poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa i stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Jak te cele są realizowane? W zakresie celu pierwszego Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada osiągnięcie wskaźnika liczby mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców. Taki cel został zapowiedziany w Narodowym Programie Mieszkaniowym. W 2015 r. były to 363 mieszkania na 1000 mieszkańców. W tej chwili to 392 mieszkania na 1000 mieszkańców, czyli przez tych pierwszych kilka lat osiągnęliśmy ponad 40% tego celu, co sugeruje, łatwo to wywnioskować, że w 2030 r. z pewnością uda się ten cel określony w Narodowym Programie Mieszkaniowym zrealizować. Oczywiście do wzrostu tego wskaźnika przyczynia się cała polityka rządu.

Mamy w 2020 r. wybudowanych ponad 220 tys. mieszkań, z czego duża część to mieszkania oparte na rozwiązaniach, które proponuje rząd Zjednoczonej Prawicy. O tym później. Drugi cel. W 2020 r. na możliwość najmu mieszkania gminnego oczekiwało 136 tys. gospodarstw domowych. To jest realizacja tego drugiego celu. O 17% zmniejszyła się kolejka osób oczekujących na mieszkanie komunalne i będzie nadal się zmniejszała, bo nasze programy są realizowane. Dzięki samorządom we współpracy z rządem. Bo my wspieramy te inicjatywy. Nigdy nie mieliśmy mniej osób oczekujących na mieszkanie gminne niż w tej chwili.

Przyczynia się do tego realizacja programów, według których na koniec sierpnia wybudowaliśmy ponad 14 tys. mieszkań, a ponad 20 tys. znajduje się w budowie.

Przewidywania na najbliższe lata są bardzo optymistyczne, gdyż będziemy mieli do czynienia z pozytywnymi efektami tego, co w tej chwili się dzieje, tych działań legislacyjnych, które również teraz podejmujemy.

W tym roku już. co powinno przełożyć się na coraz wyższe statystyki w kolejnych latach i dalsze zmniejszanie kolejek osób oczekujących na najem mieszkania gminnego. W ostatnich latach zanotowaliśmy ogromny przełom, jeśli chodzi o programy wsparcia, poprawy stanu technicznego, programy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych.

Ponadto od 2019 r. wprowadziliśmy tzw. ulgę termomodernizacyjną. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z odliczenia od podatku kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Szanowni państwo, skorzystało z tego ponad 650 tys. podatników, a kwota wynosi ponad 10 mld zł. Stworzyliśmy dwa instrumenty, które już są w Sejmie, kolejne trafią do Sejmu. Natomiast jeden wyszedł już z Sejmu, przepraszam. Jeden z priorytetów Polskiego Ładu to instrumenty wspierające rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych.

Wszyscy państwo, również z opozycji, go przyjęli i bardzo za to dziękuję.

Osoby, które z tego skorzystają, nie będą musiały mieć swoich pieniędzy na budowę budynku bądź na zakup mieszkania w banku. Będą mogły w 100% sfinansować swoją nieruchomość, swój dach nad głową. Polskie młode rodziny oczekują tego, bo sytuacja gospodarcza jest dobra, ludzie zarabiają więcej, mają pieniądze z 500+, z innych programów rządowych, stać ich na spłacanie rat kredytu. Ale często nie mają tego wkładu własnego. Nie chcą latami czekać, odkładać na ten wkład własny, bo chcą już zakładać rodzinę, chcą mieć dzieci. Nie ograniczajmy im tego, pozwólmy im na to.

To bardzo pozytywna polityka prorodzinna. Łączymy politykę mieszkaniową z polityką prorodzinną. Szanowni Państwo! Ludzie często chcieliby wybudować własny dom. Chcieliby wybudować - niekoniecznie w centrum miasta, może gdzieś w mniejszej miejscowości, może gdzieś w rodzinnej wsi - swój własny dom.

Nie chcemy zabraniać kupować kawalerek, ale jeżeli chcą wybudować 100-metrowy dom i tam wychowywać swoje dzieci, niech skorzystają z tej możliwości. Szanowni Państwo! Do zadania pytań zgłosiło się bardzo wielu posłów, więc proponuję, jeżeli państwo się zgodzą, żeby skrócić czas zadawania pytań, tak by wszyscy mogli wziąć udział w dyskusji. Oczywiście pozwolę dokończyć, ale tak, żeby to trwało krócej, dobrze? Jako pierwsza pani poseł Gabriela Masłowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, pani marszałek. Rzeczywiście Sejm nad tym pracuje, myślę, że to jest rewelacyjne rozwiązanie dla osób, które mają zdolność kredytową i nie mają pieniędzy na wkład własny, wobec tego będą mogły w rezultacie kredytem sfinansować zakup w całości mieszkania, domu lub budowę domu, łącznie z gruntem. Chciałam zapytać, dlaczego ta forma, ten program w ramach Polskiego Ładu z taką konsekwencją realizowany przez rząd ma być lepszym rozwiązaniem niż program „Mieszkanie dla młodych” Bardzo proszę, pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tej ustawy o budowie domów bez pozwolenia na budowę prezydent Lech Kaczyński by nie podpisał. Podobne rozwiązanie zostało przez pana prezydenta skierowane do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny przyznał prezydentowi rację. Wy szargacie pamięć Lecha Kaczyńskiego. I jeszcze jedno. 2018 r. O czym mówił premier Morawiecki? Obiecał 100 tys. mieszkań. Pytamy: Gdzie jest 100 tys. mieszkań? Pan premier Morawiecki okłamał Polaków. Rozpoczęliście budowę ok. 30 tys., z czego tylko kilka tysięcy zostało do tej pory ukończone. Byłyby te obiecane mieszkania, [[Dzwonek]] gdybyście nie wygasili programu „Mieszkanie dla młodych”

Zagłuszał. Pani poseł, bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proponowane w Polskim Ładzie rozwiązania mają przede wszystkim formę popytową i dotykają problemów, których rządzący nie potrafili rozwiązać przez ostatnich 5 lat.

I czy rzeczywiście uważacie, że gwarancje wkładu własnego udzielane przez Skarb Państwa i państwo polskie nie wpędzą młodych ludzi w tzw. pułapkę kredytową? Bardzo dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska. Należałoby rozliczyć to stare, co było. Mieszkanie 500+, dlaczego o tym się nie mówi? Ani razu nie padło tutaj to sformułowanie. Gdzie jest Mieszkanie 500+? Ile wybudowano? Obciążaliście samorządy, że nie chcą pomagać, nie chcą wspierać. Ale tak naprawdę ile tych mieszkań jest wybudowanych?

Pięknie ten program zaczynał działać. Zablokowaliście, bo chcieliście mieć plusa. To gdzie ten plus jest dzisiaj? Gdzie jest ten plus? Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska też proponuje. Mamy projekty: ziemia za złotówkę. Dać ludziom ze skarbu państwa ziemię za złotówkę, jeżeli chcą się budować. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na początku, bo czasu mamy mało, chcę sprostować to, co padło na tej sali, że polityka rządu jakoby skierowana jest na ludzi, mieszkańców, a nie na banki i deweloperów.

Pan poseł Szymon Pogoda, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Stanowi jeden z elementów rozwoju polityki mieszkaniowej. Opozycja krytykuje tę ustawę, argumentując m.in., że kosztami dodatkowymi zostaną obciążone samorządy, które będą musiały budować drogi czy doprowadzić media do tych domów.

Rozumiem, że dbanie o zrównoważony rozwój to dla opozycji pewnego rodzaju nowość, ale tam też żyją ludzie i trzeba to w końcu zrozumieć. Mówicie państwo również, że ustawa spowoduje chaos architektoniczny i rozlewanie się zabudowy. Chciałbym więc zapytać pana ministra, czy, jak twierdzi opozycja (Dzwonek), grozi nam jakikolwiek chaos. Dziękuję bardzo panu posłowi. Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Sibińska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Pan minister raczył powiedzieć, że macie dobry trend w polityce mieszkaniowej. Nie wiem, czy pan minister skonsultował tę wypowiedź z panem premierem, który przyznał publicznie, że program mieszkaniowy jest wielką klęską PiS. Mieszkanie+” nie wyszło, mieszkań nie ma i miejmy nadzieję, że propozycje, które popieramy.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W związku z tym mam konkretne pytania.

W jakim zakresie nastąpiło wsparcie finansowe mniej zamożnych gospodarstw domowych, jeśli chodzi o zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych? Poproszę o podanie konkretnych liczb. Czy rząd ma świadomość, że wymyślony przez rząd sposób udzielania gwarancji kredytowych na wkład własny w przypadku kredytów hipotecznych dla młodych Polaków może skończyć się dla nich taką samą pułapką kredytową jak kredyty we frankach? Czy rząd chce w ten sposób wspomóc zaprzyjaźnione banki, czy też są jakieś inne cele wprowadzania tych rozwiązań? Uprzejmie proszę o odpowiedź na piśmie. Pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Szanowni Państwo! Pytam konkretnie: Ile tysięcy zapowiadanych domów powstało do dziś? Ile do tej pory kosztowała nas obsługa tej spółki? Które z czterech strategicznych inwestycji, które miały rozpocząć się do końca 2020 r., się rozpoczęły, szanowni państwo?

Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Polska, przepraszam, Polska 2050. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oczywiście polityka mieszkaniowa dotyczy jednego z najbardziej wrażliwych obszarów dla obywateli.

Już chyba każdy w Polsce o tym słyszał, natomiast nikt nigdy w życiu na oczy tego nie widział. Nawet rządowi eksperci, oceniając pomysły rządu, z rozbrajającą szczerością pisali, że pomysły mieszkaniowe Prawa i Sprawiedliwości nie działają i nie miały prawa zadziałać. PiS zmarnował Polakom 6 lat życia, obiecując gruszki na wierzbie i kłamiąc w żywe oczy, szanowni państwo. Teraz rząd przyznaje się do porażki i będzie rozdawał pieniądze na mieszkania za urodzenie dziecka. Problem w tym, że te pomysły rządu spowodują dalszy wzrost cen mieszkań. To oznacza, że PiS szkodzi ludziom tak naprawdę, a nabija kasę (Dzwonek) nieuczciwym w gruncie rzeczy deweloperom. Mam jedno pytanie: Dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości, posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, aby ceny mieszkań rosły, co w sposób oczywisty uniemożliwi zakup mieszkań na własność zwłaszcza młodym rodzinom? Bardzo bym prosił pana ministra o odpowiedź na to kluczowe pytanie. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Od początku, kiedy moje ugrupowanie wzięło odpowiedzialność za rozwiązanie problemów mieszkaniowych polskich rodzin, stało się to dla nas ważnym zadaniem. W ostatnich latach uruchomiono naprawdę sporo różnorakich narzędzi, które są ukierunkowane na wsparcie rodzin w zakupie mieszkania, ale, co warte podkreślenia, również w jego utrzymaniu. Form wsparcia rodziny przy pomocy różnych mechanizmów jest naprawdę dużo i, co ważne, nie są to, jak za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, mechanizmy, które wspierają przede wszystkim monopol deweloperów. Stąd moje pytanie do pana ministra i prośba o przypomnienie opozycji, jakie programy już dziś służą wsparciu rodzin w pozyskiwaniu własnego mieszkania. Co więcej, wiemy, że rząd poszukuje nowych form. Dlatego proszę pana ministra o przypomnienie, jakie programy wspierające rozwój mieszkalnictwa (Dzwonek) zostaną uruchomione w ramach Polskiego Ładu. Pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Z polityki mieszkaniowej PiS na siłę chce zrobić sukces. Na razie go nie ma. Jeżeli będzie, to dopiero jesteście przed. Być może będzie, ale nie wiemy tego. Ile mieszkań zawdzięczamy polityce rządu? Ile mieszkań zostało zbudowanych dzięki rządowi PiS przez 6 lat albo przez rok ostatni? Co zrobiliście, by nie rosła cena mieszkań? Skrzętnie ominięto ten temat. Za waszych rządów o kilkadziesiąt procent, może nawet o 50% wzrosła cena mieszkań, a w ostatnim roku, w tym roku - już o kilkanaście procent. Co zrobiliście, żeby tak się nie działo? Co proponujecie, by senior mógł się przebazować na starość, na jesień życia? Jakie wsparcie finansowe? Gdzie są struktury senioralne tak popularne na zachodzie Europy? Proszę powiedzieć, proszę napisać to w odpowiedzi pisemnej. To jest jedna z ważniejszych kwestii, na które rząd PiS w ogóle nie reaguje i w ogóle nie odpowiada seniorom, co mogą zrobić, jeżeli są przykładowo więźniami czwartego piętra albo ich mieszkanie po prostu jest za duże na ich potrzeby mieszkaniowe w danym momencie, albo po prostu nie są w stanie go utrzymać. To jest gigantyczny zasób, który mógłby służyć również młodym ludziom. Bardzo proszę, pani poseł Magdalena Biejat, Lewica. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W grudniu 2020 r. Sejm uchwalił przygotowany przez minister Jadwigę Emilewicz pakiet mieszkaniowy. W ramach projektu stworzono mechanizmy zachęcające samorządy gminne do zakładania społecznych inicjatyw mieszkaniowych, tzw. SIM-ów, lub przekształcania TBS-ów w SIM-y. Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępu Polek i Polaków do mieszkań i zakłada również wspieranie społecznego budownictwa. Mam zatem konkretne pytania. Ile gmin skorzystało z tych zachęt finansowych i założyło nową społeczną inicjatywę mieszkaniową lub przekształciło istniejący TBS w SIM? Ile lokali chcą zrealizować nowo powstałe SIM-y? Na jaką liczbę mieszkań SIM-y złożyły wnioski o dofinansowanie budowy z funduszu SBC lub rządowego funduszu mieszkaniowego? Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nowe propozycje programów mieszkaniowych to jest jednoczesne przyznanie się PiS-u, że program „Mieszkanie+” to całkowita lipa. Dzisiaj nawet nie chcecie posługiwać się sformułowaniem „Mieszkanie+”, ponieważ ono jednoznacznie kojarzy się z klapą waszego programu. Natomiast mam konkretne pytania. Dlaczego, formułując nowy program mieszkaniowy w Polskim Ładzie, jednocześnie chcecie zaszkodzić osobom wynajmującym mieszkania? Wy myślicie, że na tym zaoszczędzicie, na braku odliczenia amortyzacji, ale przecież na tym stracą na początku polscy budowlańcy, a później w konsekwencji polski budżet. Czy zdajecie sobie sprawę (Dzwonek), że idziecie w kierunku budowy brazylijskich faweli w Polsce? Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Wysoka Izbo! Wszyscy mówią, łącznie z panem premierem, że wasz program „Mieszkanie+” poniósł spektakularną porażkę. Prawdopodobnie nie uda się również zapisana w tym najnowszym planie 5-letnim koncepcja spontanicznej budowy małych domków, bo to ani uporządkowane, ani ekologiczne, a wymagające zapewnienia infrastruktury i poniesienia w tym celu bardzo, bardzo dużych nakładów. Nie zmieni to zatem sytuacji ekonomicznej polskich rodzin, nie zmieni rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że dzisiejsze ceny mieszkań wykluczają i będą wykluczać z rynku setki tysięcy rodzin. Ofertę mogłyby stanowić mieszkania na wynajem, np. te budowane w systemie budownictwa społecznego, ale niezmiennie od lat, niezależnie od opcji politycznej, nie ma wyraźnego wsparcia finansowego z budżetu państwa dla TBS-ów. Dla porównania w Niemczech - 54%. No i pytanie: Jak zamierzają państwo wspierać system budownictwa społecznego?

Bardzo proszę, pan poseł Marek Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.

A przewidziane są one zarówno dla rodzin, tych o mniejszych dochodach, gorzej sytuowanych i tych wielodzietnych, jak i dla małżeństw bezdzietnych, a także osób samotnych. To m.in. gwarantowanie przez państwo wkładu własnego na zakup mieszkania, a także budowy domu, w przypadku którego formalności zostaną maksymalnie uproszczone. Istotny jest też fakt, że rodziny rozwojowe, w których przybędzie kolejne dziecko, będą mogły dodatkowo liczyć na znaczne umorzenie kredytu, i tak aż do piątego dziecka, a także na bony mieszkaniowe dla dużych rodzin. Nietrudno zatem dostrzec, że przewidziane w Polskim Ładzie rozwiązania i środki finansowe szeroko otwierają drogę polskim rodzinom do własnego lokum. Chciałbym zapytać: Jak program: mieszkanie bez wkładu własnego wpłynie na rynek mieszkaniowy i w jakim stopniu pomoże zaspokoić potrzeby mieszkaniowe młodych Polaków? Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wasz program „Mieszkanie+” to niestety fiasko. Do dziś powinniście wybudować 1 mln mieszkań.

Na kredyty, które nie mają zagwarantowanej stałej stopy oprocentowania przez cały czas kredytowania. Wy obiecywaliście oddłużenie frankowiczów, to są wasze postulaty wyborcze. Proszę o uciszenie tych pań. A dziś, w momencie kiedy są najdroższe mieszkania, namawiacie ludzi na kredyty. Tyle są warte wasze obietnice, tyle jest warta wasza rzetelność, która jest właśnie oceniana przez Najwyższa Izbę Kontroli. Dziękuję bardzo, pani poseł. Szanowne panie, bardzo proszę o spokój na sali. Szanowne panie. Bardzo proszę, pan poseł Maciej Konieczny, Lewica. Wysoka Izbo! Premier Morawiecki solennie obiecywał te 100 tys. mieszkań, a okazuje się, że wybudowano 15 tys., w budowie jest 20 tys., będzie 35 tys. i wiadomo, że nie będzie więcej. Nie da się, normalnie nie da się. Nie da się jak za Tuska, można powiedzieć. Zamiast tego co mamy? Mamy dopłaty do banków i deweloperów, żeby ceny mieszkań dalej rosły, jak za Tuska. Czy w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zupełnie porzuciło już plan wspierania publicznego, społecznego mieszkalnictwa? Czy w pełni skapitulowaliście przed deweloperami? Czy Polacy i Polki będą już skazani na ciągle rosnące ceny mieszkań wobec braku społecznej publicznej alternatywy? Wszystkie wasze obietnice w tym zakresie złamaliście. Wasze najnowsze rozwiązania związane z Nowym Ładem to jest powtórka tego, co robiła Platforma Obywatelska. To jest rzucanie pieniędzmi w banki, rzucanie pieniędzmi w deweloperów, a ceny mieszkań będą od tego tylko rosły. Pełna kapitulacja. Pani poseł Ewa Kozanecka, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Przypomnę: za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie uruchomiono żadnego programu budownictwa społecznego. Wspierano monopol deweloperów. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchomił wiele programów mieszkaniowych. Samorządy, podmioty rynku mieszkaniowego, w tym towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminne spółki mogą skorzystać z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego. Roczny budżet to 450 mln zł. Do 2009 r. wsparcie odbywało się ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zlikwidowanego przez rząd Donalda Tuska. Obecnie SIM-y mogą liczyć na państwowe grunty od Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz pokrycie do 45% kosztów budowy, a lokatorzy dostaną bon na partycypację. SIM-om czy TBS-om wystarczy nieduży kredyt na realizację inwestycji. Przypomnę, że chociażby (Dzwonek) w regionie bydgoskim wiele jest gmin, które przystępują do tych programów. Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Michał Szczerba, Koalacja Obywatelska. Nie ma pana posła. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Dzisiaj jest głód mieszkań w szczególności wśród ludzi młodych, osób o niskich dochodach. Dla nich receptą były mieszkania na wynajem. Narodowy Program Mieszkaniowy, ale też stanowisko klubu Lewicy w sprawie negocjacji Krajowego Planu Odbudowy i finansowania tych przedsięwzięć z Funduszu Odbudowy spowodowały, że wpisano tam również ewentualne finansowanie z tych środków inwestycji w zielone budownictwo wielorodzinne. Chciałbym, żeby pan minister zechciał rozszyfrować ten zapis, który znajduje się w Krajowym Planie Obudowy. Inwestycje w zielone budownictwo wielorodzinne - to jest istotne i ważne.

Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na początek bardzo chcę podziękować panu posłowi Wojciechowi Zubowskiemu za przygotowanie tematu informacji bieżącej na to posiedzenie. Przypomnę wszystkim państwu, że dzisiaj rozmawiamy o problemie mieszkalnictwa z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość wie, jak to jest ważny temat dla młodych Polaków. Natomiast totalna opozycja jak zwykle, jak wszystko, co dotyczy szczególnie Polskiego Ładu czy programów realizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, po prostu totalnie krytykuje, a szczególnie te dwa kluby, które rządziły poprzednio przez 8 lat. Ale nie ma się co dziwić, bo jeżeli samemu się nie ma programu, samemu się przez 8 lat Polskę niszczyło, to dzisiaj, tak jak to powiedział pan Donald Tusk, nieważne są programy, bo przecież kto to czyta, po co pisać programy, najważniejsze jest wygrać wybory. nie musicie go czytać, to przynajmniej przeczytajcie, nad czym dyskutujemy, o czym mówimy. Program, który teraz jest zaproponowany, jest programem bardzo ważnym. Nie powtarzajcie, że nic się nie udało, bo za rządów Prawa i Sprawiedliwości wiele się udało. Ale udało się tam, gdzie była założona współpraca z samorządami. Wszędzie tam, gdzie samorządy chciały współpracować z rządem przy realizacji „Mieszkania+”, to się udawało. Niech będzie przykładem chociażby mała miejscowość Zakliczyn, gdzie mieszkania są budowane, będą budowane. Natomiast tam, gdzie jest totalna opozycja, to samorządy robiły wszystko. żeby to nie wyszło.

Panie Posłanki! Pani Marszałek! Proszę państwa, właściwie to powinniśmy zacząć od minuty ciszy nad wszystkimi programami mieszkaniowymi Prawa i Sprawiedliwości, bo jasno mówiąc, tak naprawdę to ogłosiliście w Nowym Polskim Ładzie dezercję z zajmowania się sprawami mieszkaniowymi. Po pierwsze, ciekawą sprawą jest to, że w 2018 r. zlikwidowaliście program „Mieszkanie dla młodych”, żeby teraz wrócić do podobnego, tylko trochę gorszego. Po drugie, wasze „Mieszkanie+” okazało się kompletną porażką. Tu wiele już o tym mówiono. Kwestia drewnianych domów też nie wyszła. Ogólnie rzecz biorąc, co ma zrobić młody człowiek, którego nie stać na kredyt nie dlatego, że nie ma wkładu własnego, tylko dlatego, że nie ma stabilnej pracy, a poza tym nie chce on się na stałe wiązać z danym miastem, żeby mieć gdziekolwiek mieszkać? Nie ma żadnych rozwiązań, które pozwoliłyby młodym ludziom zakładać rodziny. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Karolina Pawliczak, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! We wrześniu 2016 r. rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy. Był to program adresowany do Polaków mających problem z najmem lub kupnem mieszkania. Miało być 100 tys. mieszkań, a jest ich tylko procent tej liczby. Z szumnych planów dotyczących rządowego programu „Mieszkanie+” udało się zrealizować niewiele. Nim budowa ruszyła na dobre pod koniec 2018 r., wiadomo było, że program będzie potężną klapą obozu rządzącego. W realizacji programu „Mieszkanie+” popełniono liczne błędy. Częste zmiany koncepcji programu, źle przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa akty prawne sprawiły, że pierwsze 2 lata jego funkcjonowania należy uznać za stracone. Kolejny projekt, który funduje nam ten rząd, w założeniach programowych może i jest słuszny, ale spóźniony o kilka lat, bo dziś, nawet z poręczeniem wkładu własnego, ceny nieruchomości są tak wysokie, że wiele osób nie ma już zdolności kredytowej, jeśli chodzi o dostępne mieszkania, a kwestia spłaty kredytu (Dzwonek) przy wzroście liczby dzieci również wydaje się chybiona. Proszę zatem powiedzieć: Czy zamierzacie państwo w tym aspekcie wesprzeć w jakimkolwiek nowym programie budownictwo komunalne, w szczególności socjalne, w ramach współpracy z samorządami? Bardzo proszę, pani poseł Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Własne cztery kąty to dla każdej rodziny poczucie stabilizacji i fundament dalszego rozwoju. No ale cóż, przyzwyczailiśmy się już do tego, że posłowie Platformy krytykują programy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale zapewniam: wasze wrzaski z sejmowej mównicy czy wygrażanie palcem nie zatrzymają realizacji naszych programów dla dobra polskich rodzin. Trzy spektakularne sukcesy: po pierwsze, podwyższenie wieku emerytalnego Polkom i Polakom, po drugie, grabież środków z OFE. a po trzecie, likwidacja Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w 2009 r. To wam się udało. Chwalicie samorządy? Ale mówcie prawdę. Mówcie, że gdyby nie wsparcie finansowe rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie byłoby budowy mieszkań. Tu konkretny przykład mojego miasta Włocławka: 58 mln zł z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego na 288 mieszkań. Panie ministrze, jest ogromne zainteresowanie programem mieszkanie bez wkładu własnego, wiele osób, szczególnie młodych osób, pyta mnie o szczegóły tego programu i z tym programem wiąże ogromne nadzieje. Od kiedy on wejdzie w życie? Kto będzie mógł do tego programu się zgłosić i z niego i z niego skorzystać, aby mieć swoje własne cztery kąty? Nie wynajęte, a własne. I jeszcze jedno króciutkie zdanie. To sformułowanie, którego użył dzisiaj pan poseł z Platformy, jest po prostu karygodne. Chcemy polskim seniorom zapewnić właśnie godne i dogodne warunki, tak by nie musieli się w jesieni życia przenosić w inne miejsce. Dziękuję bardzo. Proszę o spokój na sali. I bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Bardzo proszę o spokój. No tak, od zawsze Prawu i Sprawiedliwości bardzo dobrze wychodziły programy, propaganda, slajdy. Natomiast co z tego wynika, to widzimy cały czas od 2005 r. Panie Ministrze! Od 2015 r. zlikwidowaliście 17 kopalń. Uwolniliście zasoby nieruchomości. Chciałem pana zapytać, ile przejęliście do Krajowego Zasobu Nieruchomości tych terenów. Ile na tych terenach wybudowano mieszkań? Zlikwidowaliście miejsca pracy, ile zostało tam stworzonych miejsc pracy? My przed 2015 r. wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i ministerstwem rozwoju budowaliśmy programy budownictwa na wynajem oraz wsparcie dla budownictwa społecznego. Pytanie do pana ministra, które programy (Dzwonek) przygotowane właśnie przez Platformę Obywatelską wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostały przejęte do realizacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r. Bardzo proszę, pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tutaj z tej mównicy padło takie słowo „przebazowanie” w odniesieniu do seniorów. Chciałam tylko przypomnieć, że faktycznie, można się pokusić o takie stwierdzenie, że państwo mieliście sukces z przebazowaniem 40 tys. mieszkańców Warszawy na bruk, niestety. W tym znalazły się nawet osoby, które były kombatantami i które walczyły w powstaniu warszawskim. Ale wracając w tej chwili do tego, o czym dyskutujemy, chciałabym spytać pana ministra o kwestie związane ze spółdzielniami mieszkaniowymi. To jest ważna instytucja, ważna organizacja w życiu Polek i Polaków.

Bardzo proszę, pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Posłowie! Nie wyszło, ale mnie to nie dziwi, bo nie wiem właściwie, co panu premierowi wyszło. Ale mam dość dobrą pamięć i sobie przypominam, jak pan prezes Jarosław Kaczyński obiecał 3 mln mieszkań. No to ja was pytam, gdzie są te 3 mln mieszkań? Naprawdę, wchodzić na tę mównicę i mówić, że macie programy i że dla was sprawy mieszkańców i rodzin są takie ważne i ten własny kąt.

Już nie będę mówiła, co to zrobi z naszym zagospodarowaniem przestrzennym, krajobrazem, miastami i podmiejskimi terenami. Ale jak wy mówicie o tych domach, to mi się przypomina ten polski dom drewniany i pan minister Kowalczyk, który mówił, że w roku (Dzwonek) 5 tys. tych domów powstanie. I w ogóle jak to będzie świetnie i jak to będzie znakomicie. Spółka, a potem agencja. Tak jak powstał Narodowy Program Mieszkaniowy. Bo wy myślicie, że jak coś nazwiecie „narodowe”, to już macie załatwione. Pan poseł Patryk Wicher, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Powiem na początku coś, co jest najważniejsze. Polacy oczekują właśnie na te mieszkania. Drodzy państwo, walczmy o Polaków, walczmy o te mieszkania, walczmy, żeby ten program był jak najlepszy, a nie bawmy się we wspominki, które nikomu nic nie dadzą.

Czy trzeba zakładać dziennik budowy? Jeśli tak, to czy w pełnym wymiarze, czy w jakimś okrojonym? Czy ewentualnie trzeba zatrudniać kierownika budowy? Jeśli nie, kto będzie pełnił funkcje nadzorcze w kontekście budowy tych domów? A więc to są takie niby techniczne, ale bardzo ważne (Dzwonek) dla mieszkańców pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Gdzie te niskie czynsze z Mieszkania+?

Sukces TBS-ów poprzednich rządów zawłaszczacie, zmieniając tylko nazwę na SIM.

Szkoda, że to taki bubel+.

Proszę przeczytać. Po drugie, chwalicie się wprowadzeniem określenia decyzji o warunkach zabudowy. To właśnie jest dokładnie tak określone, od 18 lat to obowiązuje, tylko w rozporządzeniu do ustawy. To jest zakłamanie, hipokryzja, okłamywanie ludzie. Zwyczajnie kopiujecie zapisy już istniejące, manipulując, że to są wasze nowe pomysły. Wstyd! Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W naszych biurach poselskich, a także na różnych spotkaniach rozmawiamy z mieszkańcami o ich potrzebach i trudnościach.

Własne mieszkanie jest marzeniem wielu osób. Jego posiadanie nie jest w dzisiejszym świecie czymś niezwykłym. Jest podstawowym dobrem, by móc funkcjonować w sposób spokojny, planować swoje dalsze życie. Stąd moje pytanie brzmi: Jak zmieniają się wskaźniki dostępności mieszkań dla obywateli? Pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W 2016 r. deklarowaliście, że Narodowy Program Mieszkaniowy będzie służył rozwijaniu sektora mieszkań na wynajem, tak żeby stały się tańsze i bardziej dostępne. Obiecywaliście 100 tys. mieszkań, a ile powstało? Niespełna 12 tys. Jednak najbardziej martwi mnie to, że w Polskim Ładzie wycofaliście się z tego, o czym sami wcześniej mówiliście.

Wróciliście także do dopłat do kredytów. W związku z tym mam pytanie: Któremu rządowi powinniśmy wierzyć? Temu sprzed 5 lat, który chociaż deklarował dobre pomysły, czy temu, który chce wspierać banki i patodeweloperów? Możecie się na coś zdecydować? Panie Ministrze! Dziękuję bardzo. Pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rządowy program powstał, by wspierać wszystkich, którzy z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie. Dzięki realizacji programów w Polsce pojawiają się kolejne mieszkania i będą się pojawiać. Są to bardzo dobre kierunki rozwojowe. Proszę, panie ministrze, udzielić mi informacji, bo tutaj nam totalna opozycja zarzuca, że coś robimy po nich, że w ogóle nic nie robimy, proszę, żeby pan minister udzielił informacji, jakie były dotacje finansowe w latach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, a jak jest obecnie, od 2015 r. do czasów obecnych. Totalna opozycja miała program, który nie został zrealizowany, a wszystkie dobre decyzje, które obecnie rząd podejmuje, są torpedowane. Pamiętamy słowa: państwo teoretyczne. Bardzo proszę, pani poseł Mirosława Nykiel, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Wszystko, co obiecują rządy PiS, opiera się na trzech zasadach. Pierwsza: obiecać nic nie kosztuje, bo jak nie wyjdzie, to się jakoś wytłumaczy albo zminusuje. Druga: wszystko musi być plus, bo jest dobrze kojarzone, bo ludzie myślą, że im coś dodajemy. I trzecia zasada: poprzednicy nic nie zrobili, a my jesteśmy najlepsi. Do tej pory z tych obietnic oprócz rozdawnictwa pieniędzy nic wam nie wyszło. Ogłoszony wielki projekt SOR - klapa, główny wskaźnik inwestycji, stopy inwestycji legł w gruzach. Czy tak też będzie z wielkim planem Polski Ład? W dziedzinie mieszkalnictwa - już to wiele razy mówiono - też wam nic nie wyszło. A ceny mieszkań szaleją, inflacja też.

Chodzi o to, czy będzie stosowana zasada ochrony inwestycji w toku? Czy ta zasada będzie stosowana?

Wysoki Sejmie! Od roku 2016 systematycznie wzrasta liczba budowanych i oddawanych do użytku mieszkań. Lata 2019 i 2020 jak do tej pory były pod tym względem rekordowe. Nawet tytuły prasowe informowały o tym, że tak dużo mieszkań nie zbudowano w Polsce od prawie 40 lat.

Raport firmy Deloitte za rok 2021 podaje, że było to 5,79 mieszkania na 1 tys. obywateli i jest to najwyższy wynik w Europie. Jednak to nie oznacza, że potrzeby mieszkaniowe naszych obywateli zostały zaspokojone, stąd m.in. w Polskim Ładzie znalazły się domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m budowane (Dzwonek) bez pozwolenia. W związku z tym mam pytanie do pana ministra: Jak przedstawia się sytuacja budownictwa mieszkaniowego i jego różnych form po roku 2016 w porównaniu właśnie z poprzednimi latami przed 2016 r. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Niedługo, jak mówił klasyk, nie będzie niczego. Natomiast w sytuacji, w której deweloperzy wypowiadają umowy, bo nie są w stanie zrealizować nieruchomości za wcześniej ustalone kwoty, w sytuacji, w której tysiące Polaków posiadających kredyty hipoteczne mają problem z rozliczeniem kolejnej transzy, bo materiały budowlane z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc drożeją o 100–200%, co państwo proponujecie? Kredyty hipoteczne. Mam pytanie: Czy państwo weźmiecie odpowiedzialność za dramaty tysięcy ludzi, jakie pojawią się w przyszłości, kiedy stopa procentowa będzie na właściwym poziomie, a nie tak jak dzisiaj, zaniżonym, kiedy ludzie będą tracić te nieruchomości, kiedy komornicy zapukają do ich drzwi? Jeszcze jedno zdanie, pani marszałek, bo panie podważają sformułowania dotyczące polityki senioralnej w zakresie mieszkalnictwa. Proszę państwa, jeżeli państwo nie widzicie problemów (Dzwonek) milionów polskich seniorów, którzy mieszkają w za dużych mieszkaniach na trzecim, czwartym piętrze, nie są w stanie ponieść kosztów utrzymania tego mieszkania, nie są w stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chcę zdementować, że ludzie nie chcą mieszkań plus. W Radomiu o 124 bodajże lokale ubiega się 1100 obywateli. Chcę powiedzieć też o Witnicy, z mojego lubuskiego, pani poseł mówiła również o klapie programu „Mieszkanie+” Nieprawda, „Mieszkanie+” jest realizowane przy ogromnym oporze radnych z opozycji. krzyczycie państwo przy programie mieszkaniowym, a przez 8 lat działalności PO-PSL na mieszkalnictwo przeznaczono 560 mln, natomiast już (Dzwonek) w roku 2019 500 mln. Pytanie o najbiedniejszych, najmniej zasobnych, panie ministrze. Jaki jest program mieszkaniowy dla tych ludzi?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Opozycja mówi coś o chaosie. Ja się zgadzam z tym, tyle tylko, że ten chaos jest spowodowany przede wszystkim dobrymi rozwiązaniami proponowanymi przez polski rząd w ramach Polskiego Ładu dla naszych rodzin. A teraz do rzeczy. Posiadanie własnego mieszkania jest jednym z podstawowych dóbr, o których marzą Polacy, tym bardziej jest nim posiadanie choćby małego domku. Kto budował jakąkolwiek budowlę, kto budował dom, wie, jak długa i mozolna jest procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę. Dlatego każde uproszczenie, panie ministrze, tej procedury jest przyjmowane z dużym zadowoleniem. Ale pytanie, panie ministrze, do pana jest takie: (Dzwonek) Chodzi mi o dokumenty, które będzie musiał złożyć wnioskodawca do tego zgłoszenia.

Pani Marszałek! Panie Ministrze!

To wskazuje, że było zapotrzebowanie na takie mieszkania dla osób, które mają za niskie dochody, żeby sięgnąć po kredyt hipoteczny, a za wysokie, żeby się starać o mieszkanie komunalne. W ramach tego programu jest w trakcie budowy lub zbudowano 35 tys. mieszkań, szanowni państwo. Czy wy tego nie widzicie, nie słyszycie? Natomiast jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to w tej chwili, w ubiegłym roku oddano 221 tys. mieszkań. To tylko za Gierka, panie ministrze Grabarczyk, było więcej, ale wtedy były niskiej jakości, teraz są (Dzwonek) mieszkania o większej powierzchni. Panie ministrze, moje pytanie: Czy ten program będzie kontynuowany? A jeśli nie, to dlaczego?

A państwo tego nie widzicie. I na koniec powiem tak: jeśli państwo chcecie być jeszcze w opozycji, kontynuujcie takie rozmowy jak w tej chwili w Sejmie. Bardzo proszę, pani poseł Anna Ewa Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rząd Zjednoczonej Prawicy wychodzi naprzeciw polskim rodzinom, naprzeciw tym, którzy z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania. Dzięki programom wspierającym budownictwo mieszkaniowe z każdym rokiem powstają nowe mieszkania. Szanowni państwo, tutaj nie zabrakło miejsca na budownictwo, na wsparcie budownictwa. Panie Ministrze!

Chcą budować te nasze piękne małe ojczyzny, tam inwestować, tam pozostać.

Panie Ministrze! Z badań wynika, że synonimem indywidualnego szczęścia Polaków jest szczęście rodzinne. Młodzi ludzie deklarują, że chcą mieć dwoje lub troje dzieci. Wydawałoby się, że zapaść demograficzna nam nie grozi. Na ten kryzys demograficzny, który mamy teraz, pracowaliśmy przez 30 lat.

Mam pytanie do pana ministra.

Bardzo proszę, pan poseł Aleksander Mrówczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tylko krytyka. My czynimy tyle dobra, a wy mówicie, że tyle zła.

Te 3 mln mieszkań też wybudujemy, bo chcemy długo rządzić. A teraz konkretnie. Nowy pakiet mieszkaniowy daje nadzieję, że budownictwo komunalne złapie wiatr w żagle, że powstanie więcej mieszkań i kolejki oczekujących w końcu się skrócą. Jedną z najważniejszych zmian jest znaczący wzrost wysokości dofinansowania dla gmin, którego udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wiem, że dzisiaj mnóstwo samorządów wchodzi do tego programu, bo przecież mówimy o mieszkaniach, na które bardzo często ludzi nie stać. Czy w ramach tego programu, panie ministrze, można uzyskać środki na dofinansowanie remontów istniejących zasobów komunalnych? Czy w krajowym programie odbudowy uwzględniono problematykę mieszkaniową? Dziękuję bardzo. Pani poseł Beata Strzałka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Posiadanie mieszkania to nie tylko status czy komfort. To przede wszystkim podstawa bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. Rozwiązania finansowe zaproponowane w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym to dla wielu młodych ludzi, dla rodzin marzących o własnym kącie jedyny sposób na zdobycie środków na wymagany wkład własny przy kredycie hipotecznym. Ten czynnik bywa główną barierą zaporową w ubieganiu się o kredyt. Niestety banki zaostrzają kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Dziś wkład własny to średnio 20% wnioskowanej kwoty, a bywa również, przy zwiększonym ryzyku kredytowym, że jest to powyżej tej granicy procentowej. Niestety bardzo często młodzi ludzie nie mogą zgromadzić wymaganej kwoty, 80 tys. zł czy 100 tys. zł, na wkład własny. Panie Ministrze! Ile do wkładu własnego dopłaci rząd i na jakich warunkach? Co jest istotą rozwiązań przedstawionych przez rząd w ramach gwarantowanego kredytu mieszkaniowego? Pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Bardzo proszę, pan poseł Piotr Uruski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Droga Opozycjo! Tak, to była klapa. 8 lat rządów Platformy i PSL-u to była jedna wielka klapa. Potrzeby mieszkaniowe w Polsce są ogromne. Mieszkań potrzeba tak jak. Potrzeby mieszkaniowe to tak jak w biblijnym psalmie.

Pan poseł Grzegorz Adam Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł Agnieszka Górska, Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dla budownictwa społecznego nie zrobiliście nic albo prawie nic, ale obietnic jak zwykle przy każdej okazji było bardzo dużo. Exposé premiera Donalda Tuska z 2007 r.: stworzymy takie warunki, aby Polacy mogli budować na tańszych gruntach. Exposé premiera z 2011 r.: myślimy o tym, żeby tym razem skuteczniej niż do tej pory zbudować przepisy prawa, np. kiedy mówimy o pozwoleniu na budowę. Exposé premier Ewy Kopacz z 2014 r.: Polacy czekają od wielu lat na Kodeks budowlany, który uprości procedury związane z budową m.in. domów jednorodzinnych. I dziś macie czelność mówić, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nic nie zrobił w tej sprawie. A wy? To obłuda z waszych ust. Może właśnie wspieraliście monopol deweloperów.

Jest pan poseł? Ostatnie pytanie zadaje pani poseł Daria Gosek-Popiołek, Lewica. Wysoka Izbo! 35 tys. mieszkań zamiast 100 tys. i pani poseł, która chwali się tym, że w Radomiu na 100 wybudowanych przez was mieszkań jest 1000 czekających rodzin. Myślę że obydwie strony powinny ze sobą poważnie porozmawiać na temat tego, jak nie robi się polityki mieszkaniowej. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze, czekajcie państwo na naszą, bo my dokładnie wiemy, czego potrzebujemy. Nie potrzebujemy dotować deweloperów, bo oni sobie poradzą. Teraz pytanie.

Tego właśnie potrzebujemy. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Wojciecha Zubowskiego. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Z informacji uzyskiwanych podczas dyżurów poselskich wynika, że rozwiązań jest tak dużo, że problemem może być wręcz momentami niewiedza obywateli o już funkcjonujących lub wprowadzanych rozwiązaniach. Nie wszyscy wiedzą o pożyczce z Funduszu Dostępności pozwalającej osobom ze szczególnymi potrzebami na likwidację barier architektonicznych, która może być częściowo umorzona lub połączona z dotacją ze środków PFRON-u. Mamy też Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pozwalający na otrzymanie do 2 tys. zł miesięcznie na okres do 36 miesięcy na spłatę kredytu mieszkaniowego. Są programy, które już funkcjonują albo wkrótce zaczną funkcjonować, a nie zawsze ich potencjalni beneficjenci mają wiedzę, że mogą z nich skorzystać. Warto więc zastanowić się, czy polityka informacyjna nie wymaga sprawdzenia, bo na takie wykluczenie informacyjne najczęściej narażeni są mieszkańcy mniejszych miejscowości. A przecież to dla nich tworzone są społeczne inicjatywy mieszkaniowe, dzięki którym można liczyć na państwowe grunty od Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz na pokrycie do 45% kosztów budowy.

Mieszkańcy na to czekają. Jest też pomoc dla kredytobiorców, którzy zdecydują się na dzieci, czy też bon mieszkaniowy. Szkoda, proszę państwa, że część opozycji zamiast konstruktywnej dyskusji wolała przy tak ważnym temacie robić z sali plenarnej ring dla politycznych pyskówek. Mało tego, wskaźniki, które przedstawiłem w swoim pierwszym wystąpieniu, nie pozostawiają wątpliwości, że sytuacja na rynku mieszkaniowym się polepsza, i bez względu na zaklęcia opozycji obywatele to widzą. Na politykę mieszkaniową, na mieszkania socjalne czy komunalne przeznacza się więcej środków. Pojawiły się programy wcześniej niedostępne, mało tego, są programy kierowane do posiadaczy mieszkań czy domów, programy umożliwiające sfinansowanie nowego lokum lub tego już posiadanego. Liczby nie kłamią, więc przypomnę raz jeszcze: rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczył więcej środków na politykę mieszkaniową niż rządy PO i PSL. Przypomnę dane z roku 2020: rekordowa ilość mieszkań, dwa razy więcej środków w dwa razy krótszym czasie na budownictwo społeczne i wiele innych. Buduje się rekordową ilość mieszkań i owszem, są to też mieszkania budowane przez samorządy, ale dzięki wsparciu rządowych programów, których kiedyś nie było. Przypomnę taki cytat: Dobry rząd jest od tego, żeby stworzyć warunki i ramy prawne, szczególnie dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Myślę tu także o szeroko zakrojonej debiurokratyzacji tej dziedziny życia, jaką jest indywidualne inwestowanie we własne mieszkanie, we własny dom. To jest fragment exposé Donalda Tuska, proszę państwa. Ewa Kopacz mówiła przecież: Polacy czekają od wielu lat na kodeks budowlany, który uprości procedury związane z budową m.in. domów jednorodzinnych. Bo to jest program Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy? Bo to program dla ludzi? Bo się cieszy poparciem społecznym? Bo jest oczekiwany? Zapewniam opozycję, że nie chcemy budować, jak to określiliście, brazylijskich faweli. My chcemy, by Polacy mogli godnie żyć we własnych mieszkaniach. Wy woleliście głosować przeciw. Skoro więc nie chcecie poprzeć dobrych dla Polaków rozwiązań, to choć nie przeszkadzajcie nam w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych naszych rodaków. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pana Piotra Uścińskiego.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Tak jak dzisiaj powiedziano, Polacy chcą budować własne domy, chcą mieszkać na przedmieściach, chcą mieszkać w małych miejscowościach, w rodzinnych miejscowościach, a my taką szansę chcemy im dać.

Zrobi to taniej, trzeba dać mu tylko szansę.

Planowanie przestrzenne to jest kompetencja samorządu i my tej kompetencji w żaden sposób nie odbieramy.

Były pytania o kierownika budowy i dziennik budowy.

Z tego rozwiązania będą korzystali ci, którzy znają się sami na budowie i są w stanie sami tę budowę nadzorować, kierować procesem budowlanym, ci, którzy podpiszą oświadczenie, że biorą na siebie całą odpowiedzialność spoczywającą na kierowniku budowy.

Szanowni Państwo!

Teraz komisja dodała: przy nadbudowie czy rozbudowie skutkującej powstaniem nowego lokalu mieszkalnego. My te pieniądze gwarantujemy, ale to nie jest wielki koszt dla państwa. Kosztem będzie. Nawet nie kosztem, źle mówię. To będzie inwestycja w młode pokolenie, bo pieniądze z budżetu państwa będą wydawane w tym programie wtedy, kiedy będą rodziły się dzieci: 20 tys. na drugie dziecko, po 60 tys. na kolejne dzieci. To będą te miliardy. I niech te miliardy będą wydawane. Niech te dzieci się rodzą. Ten program uzupełnia nasz program prorodzinny i prodemograficzny.

Jak ma podejmować decyzję o trzecim czy czwartym dziecku?

My w tej ustawie wprowadzamy mechanizm ograniczający wpływ tej ustawy na wzrost cen nieruchomości. Jest limit ceny, do tego jest elastycznie zarządzany, regulowany, w zależności od sytuacji na rynku, tak żeby ta ustawa nie wpływała, i nie będzie wpływała, na wzrost cen na rynku nieruchomości. Były z państwa strony pytania dotyczące tego, ile rocznie w Polsce się buduje. Szanowni państwo, chciałem państwu pokazać.

Te granatowe, niebieskie słupki to są mieszkania społeczne, mieszkania rynkowe realizowane przez PFRN, te czerwone to są mieszkania komunalne. Budujemy również te mieszkania społeczne. Mam tutaj listę inwestycji. Każda pozycja na tej liście to jest konkretna gmina, konkretny blok, konkretne kilkadziesiąt mieszkań, w których zamieszkają polskie rodziny. Nie będę tego wszystkiego opowiadał. To te 35 tys. mieszkań, które faktycznie powstają. Wasz program MdM dawał tylko pieniądze na zakup mieszkania u dewelopera. My te mieszkania realnie budujemy i wspieramy polskie rodziny w tym, żeby mogły zamieszkać we własnym lokalu, nawet jeśli nie mają wkładu własnego.

Pytaliście, ile się w Polsce rocznie buduje. 220 tys., ponad 220 tys. mieszkań rocznie. To jest polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, ostatnich kilku lat. Za waszych rządów, mimo programu MdM, w którym dawaliście pieniądze deweloperom, ci deweloperzy nie budowali tyle, ile teraz budują. Teraz budują dużo więcej. 2021 r., ten obecny, to będzie kilka procent wzrostu w stosunku do poprzedniego roku.

Było też pytanie o SIM-y, czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe, ile ich jest.

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, 844 mln na 317 wniosków dotyczących SIM-ów i TBS-ów. Szanowni Państwo!

Natomiast ci, których nie stać, którzy nie mają teraz zdolności kredytowej, ci, którzy będą chcieli skorzystać z budownictwa czynszowego, z TBS-ów, SIM-u, ze spółdzielni mieszkaniowych, będą mogli skorzystać z bonu mieszkaniowego, który wesprze ich w zapewnieniu wkładu własnego. To też pomoże po tej stronie podażowej w lepszym przygotowywaniu, w szybszym przygotowywaniu inwestycji, tak jak zrobiliśmy i przygotowaliśmy cyfryzację (Dzwonek) map geodezyjnych, cyfryzację procesów związanych z pozwoleniami budowlanymi, z Prawem budowlanym. To wszystko działa i cyfryzacja w Polsce różnych procesów, tych właśnie, jest na najwyższym poziomie. W Unii Europejskiej mało jest krajów, które mają mapy geodezyjne tak dostępne, jak te, które w tej chwili udostępniliśmy. Szanowni Państwo! Uważam, że polityka mieszkaniowa rządu Zjednoczonej Prawicy to jest sukces. My ten sukces będziemy kontynuować i te projekty, nad którymi dzisiaj procedujemy w Sejmie i w Senacie, są tego dobrą kontynuacją. Polski Ład jest dla Polaków i zapewni Polakom mieszkania, dach nad głową polskim rodzinom. Dziękuję. Wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego.

Proszę panią poseł Mirosławę Stachowiak-Różecką o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, druk nr 1582. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 16 września 2021 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania. Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Pani Marszałek! Kilka zdań. Myślę, że mogłabym ten projekt odczytać, jeśli pani wyraża zgodę. Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Art. 2. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest świętem państwowym. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jeśli państwo pozwolicie, chciałabym powiedzieć z dumą jeszcze jedno zdanie. Jest dla mnie szczególnym zaszczytem, że mogłam reprezentować komisję kultury i sprawozdawać przed państwem ten projekt. Sama jestem prawnuczką powstańca wielkopolskiego. Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni i będziemy bardzo dobrze, wzorowo dbać o to, żeby rzeczywiście to święto, które uchwalimy, przynosiło chlubę, oddawało hołd uczestnikom, powstańcom wielkopolskim. Będziemy takim pierwszym frontem i przykładem.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Pierwszy pan poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Mam zaszczyt przemawiać w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za podjęcie tej inicjatywy. Do tej wdzięczności naszego klubu dołączam moją osobistą wdzięczność jako poznaniak i jako Wielkopolanin. Trzeba docenić, że to kolejna ważna inicjatywa naszego prezydenta związana z powstaniem wielkopolskim. Pamiętamy jego piękne słowa w Poznaniu 27 grudnia 2018 r. w dniu stulecia wybuchu powstania wielkopolskiego, jego słowa o męstwie Wielkopolan, a także świadomość tego, że powstanie wielkopolskie jest osadzone w długiej, historycznej tradycji. Tego dnia prezydent odwiedził także Mosinę, żeby pokazać, że powstanie wielkopolskie to nie tylko moje miasto, Poznań, ale także aglomeracja poznańska, cała Wielkopolska, historyczna Wielkopolska, a więc także niektóre z terenów, które leżą dzisiaj w sąsiednich województwach. Trzeba też przy tej okazji przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda jest tą głową państwa, która po 25 latach starań Wielkopolan podjęła sprawę uhonorowania dwóch dowódców powstania wielkopolskiego: gen. Stanisława Taczaka i gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Z różnych powodów one nigdy nie kończyły się sukcesem. W listopadzie 2018 r. spotkałem się z panem prezydentem Andrzejem Dudą i raz jeszcze przedstawiłem wszystkie racje, które przemawiają za tym, aby naszych dowódców odznaczyć. Czułem się w obowiązku jako członek korporacji akademickiej Lechia, której obaj dowódcy byli honorowymi członkami. Jesteśmy wdzięczni prezydentowi za działania, które konsekwentnie podejmuje w sprawach powstania wielkopolskiego. Wielkopolska, drogie panie i panowie posłowie, ma dwie wielkie tradycje: tradycję organicznikowską i tradycję insurekcyjną. Wysoka Izba w ostatnich latach kilkakrotnie przypominała o tradycji organicznikowskiej. Temu służyły uchwały upamiętniające powstanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Międzynarodowe Targi Poznańskie czy zupełnie niedawno pierwszego prezydenta Poznania po odzyskaniu niepodległości Jarogniewa Drwęskiego. Ale nie mniej istotna, choć nie kojarząca się z Wielkopolską, jest także tradycja insurekcyjna. To w Wielkopolsce miały miejsce dwa zwycięskie powstania: w roku 1806, które Wysoka Izba w 2016 r. przypomniała i upamiętniła - miałem wtedy zaszczyt zaproponować tekst tej uchwały - oraz oczywiście wielkie powstanie z 1918 i 1919 r. Powstanie wielkopolskie, mimo że zwycięskie, tak bardzo i tak mocno nie wryło się w naszą historyczną świadomość jak powstania listopadowe czy styczniowe. Częściej mówimy gloria victis, rzadziej gloria victoribus. Dzięki m.in. tej inicjatywie prezydenta, w związku z tym, że staje się to świętem państwowym, wszyscy w kraju będziemy mogli pamiętać, przypominać, oddawać hołd powstańcom wielkopolskim. Tak że bardzo dobrze, że prezydent z tą inicjatywą wystąpił, a właściwie przychylił się do szerokiej inicjatywy samorządowców, społeczników z Wielkopolski, także często bezimiennych, którzy ideę, aby dzień wybuchu powstania wielkopolskiego był świętem ogólnonarodowym, od lat propagowali. Przypominam jego nazwisko, ale myślę, że takich osób było dużo, dużo więcej na terenie całej Wielkopolski. Ustawa, którą mamy uchwalić, przypomina powstanie wielkopolskie, ale ma też szersze znaczenie, bo pamiętamy (Dzwonek), że powstańcy wielkopolscy walczyli także w powstaniach śląskich, bronili Lwowa, walczyli dzielnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Raz jeszcze bardzo dziękuję prezydentowi. Proszę Wysoką Izbę - myślę, że będzie to decyzja podjęta wspólnie, ponad podziałami - o to, żeby możliwie szybko były kontynuowane prace w parlamencie i abyśmy już w tym roku mogli cieszyć się świętem zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Rafał Grupiński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To rzeczywiście niezwykle ważny czas dla wszystkich Wielkopolan, czas upamiętnienia we właściwy sposób czynu, zrywu Wielkopolan tuż po zakończeniu I wojny światowej. To jest historia insurekcji zwycięskiej. Kiedy wchodzi się w Internet i wpisuje się słowo „powstanie”, to powstanie wielkopolskie pokazuje się jako ostatnie, po wszystkich przegranych powstaniach narodowych.

Po pierwsze, z powodu właśnie XIX-wiecznej pracy organicznej Wielkopolan, pracy u podstaw, budowania społeczeństwa świadomego swoich celów, patriotycznego i jednocześnie edukowanego ku przyszłej, niepodległej Rzeczypospolitej. Wszelkie towarzystwa, takie jak czytelnie ludowe, banki spółdzielcze, spółdzielnie rolne, ba, towarzystwa gimnastyczne, towarzystwa śpiewacze - wszystko to tworzyło tkankę ludzi, którzy po prostu chcieli wolnej Wielkopolski i wolnej Rzeczypospolitej. O tym naprawdę warto pamiętać.

O czym chcę powiedzieć?

Od 2008 r., czyli od 90. rocznicy powstania wielkopolskiego, dzień po rocznicy wybuchu powstania organizowane są obchody w Warszawie, w stolicy państwa, żeby w ten sposób propagować powstanie. Jest to bez wątpienia osobista zasługa marszałka Marka Woźniaka. Dzisiaj ustanowienie tego święta jest oczywiście czymś dla nas szczególnie istotnym.

Cieszymy się, że pan prezydent podjął tę lokalną inicjatywę i postanowił przekształcić to w święto państwowe.

Otóż mówię o moim małym miasteczku Wronki. Przeczytam fragment pamiętnika związany z tym miejscem. Otóż: przyjechał z Poznania do Wronek mój przyjaciel z lat młodości i ławy szkolnej dr Stanisław Krzyżankiewicz, mianowany w Poznaniu wiceprezydentem Policji, a zarazem członkiem Rady Ludowej. Przyjechał do rodzinnego miasta, by zorganizować władzę na miasto i pod jego nadzorem dokonano zburzenia pomnika Wilhelma II i ścięcia lipy Friedenslinde, drzewa pokoju, posadzonego na pamiątkę zwycięstwa armii pruskiej nad Francuzami.

Następnie poszczególne urzędy zostały przez Polaków zajęte, zaś dalszych urzędników niemieckich usuwano w miarę odpowiedniego dokształcania naszych, a we Wronkach powstała komora celna i przepustkowa. Wybudowano barak dla przyjezdnych do rewizji bagażu oraz podróżnych udających się za granicę. Oddział wojska zajął więzienia centralne i władza wojskowa wspólnie z cywilną działała na dworcu przy kontroli i obsłudze pociągów. Było to konieczne, ponieważ kolejarze niektórzy zaczęli wyłamywać się spod obowiązków. Zajechał maszynista do Rokietnicy i dalej ani rusz. Trzeba było postawić żołnierza z karabinem, aby go zniewolić do wykonania rozkazu. Wojsko uczciwie i sumiennie spełniało swoje rozkazy, natomiast inni funkcjonariusze, zwłaszcza przy badaniach przepustkowych, nie zawsze okazywali się służbowi, a gdy została zorganizowana Policja z komendantem Skąpskim na czele, to ja powołany przez wiceprezydenta Krzyżankiewicza do nadzoru stałem się dla Policji bardzo niewygodny. Nie podobało się, że miałem na dworcu nadzór, że odbierałem skonfiskowane rzeczy, że przekazywałem je do Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Urzędowałem tam z ppor. Błażejewskim, a później wyjechałem najpierw do Bydgoszczy, potem do Chojnic, gdzie pozostałem do dnia odwołania ppor. Błażejewskiego, a po pewnym czasie poprosiłem w urzędzie wywiadowczym, przefirmowanym na Urząd Bezpieczeństwa, o zwolnienie ze służby. W tym czasie gen. Dowbor-Muśnicki przeprowadzał wzdłuż granicy inspekcje, gen. Haller dokonał zaślubin Bałtyku, a niemieccy kolejarze w Chojnicach ryczeli „Deutschland über alles”

Przemycano do Niemiec masło, zboże wbrew władzom powstańczym, ale daliśmy radę, patriotyzm zwyciężył nad tego rodzaju słabościami. Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Kretkowska, Lewica. Wysoka Izbo! Powstanie wielkopolskie było jednym z zaledwie pięciu zwycięskich polskich powstań.

Oprócz tej ogromnej zdobyczy terytorialnej powstanie przyniosło też największe w 1000-letniej historii oręża polskiego łupy wojenne. Zginęło w nim 2289 powstańców, ponad 6 tys. odniosło rany. Już 16 lutego 1919 r. nastąpiło formalne zakończenie walk na mocy pokoju w Trewirze. Powstańcy wielkopolscy odnieśli dyplomatyczne zwycięstwo, uwieńczone podpisanym 28 czerwca 1919 r. traktatem wersalskim, w wyniku którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. Fakt, że powstanie trwało krótko, niekiedy kwitowany jest żartobliwie, iż cały wysiłek powstańców ograniczał się do zakupy peronówek, by wejść na dworzec w Poznaniu i owacyjnie powitać przybywającego tu pociągiem, mimo zakazu, Ignacego Paderewskiego. To oczywiście nieprawda. Powstanie miało elementy spontanicznego zrywu, ale tak naprawdę było dobrze przemyślane, porządnie, po poznańsku przygotowane i obfitowało w genialne posunięcia taktyczne. Jego podwaliny to cały okres zaboru pruskiego i skutecznego oporu Wielkopolan przed naporem kulturkampfu, germanizacji, prób ekonomicznego podporządkowania niemieckiemu kapitałowi. Wielkopolanie wygrali tę najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy zarówno ofiarnymi zrywami zbrojnymi, często niesłusznie zapominanymi, jak i mozolną, upartą strategią samomodernizacji i wzmacniania gospodarczego, inwestowaniem w naukę, edukację, kulturę, w podnoszenie wielkopolskiego rolnictwa według najnowocześniejszych wzorców. Działały tu specyficzne cechy Wielkopolan: realizm, racjonalizm, trzeźwe liczenie się z rzeczywistością, dobra organizacja i porządek. Wbrew stereotypom owa wielkopolska odmienność nie była wynikiem przejęcia niektórych cech pruskiego zaborcy, lecz była zrodzona wcześniej, jeszcze w średniowieczu. I to te cechy Wielkopolan powodowały, że Wielkopolska od średniowiecza przez cały okres nowożytny była najsilniej zurbanizowanym, zorganizowanym w kraju regionem, jedynym, który mimo wojen wykazywał stały wzrost gospodarczy. Ów melanż zapobiegliwości, zdrowego rozsądku i umiłowania porządku wraz z głęboko zakorzenionym patriotyzmem przełożył się na charakter i przebieg powstania wielkopolskiego oraz na jego zwycięstwo. W XIX w. ów melanż zaowocował zarówno społeczno-ekonomiczną samomodernizacją, jak i dalekowzrocznym formowaniem przyszłych oddziałów zbrojnych w postaci konspiracyjnych drużyn skautów czy oddziałów „Sokoła”, które już na początku I wojny światowej przeszły z trybu pokojowego na bojowo-niepodległościowy. Walczyli na wszystkich frontach Europy, a nabyte doświadczenie wojskowe, znajomość języka niemieckiego, kontakty z żołnierzami i oficerami niemieckimi wykorzystali w czasie powstania wielkopolskiego. 15 lutego 1918 r. powołano Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Polscy żołnierze służący wcześniej w niemieckiej armii przejmowali kontrolę nad radiostacjami, łącznicami telegraficznymi, całymi koszarami i arsenałami. 25 grudnia w Buku przejęli np. cały pociąg z bronią zmierzający do Poznania. Koronkową operacją przeprowadzoną bezkrwawo był tzw. zamach na ratusz 13 listopada, gdy Polacy przerwali obrady niemieckiego Komitetu Wykonawczego Rady Żołnierzy w Poznaniu. Wkroczyli do ratusza i perswazją zastąpili czterech Niemców czterema Polakami, zyskując tym samym kontrolę nad komitetem. Płomienne przemówienie Ignacego Paderewskiego z balkonu hotelu Bazar było jedynie iskrą do lontu, który był dobrze przygotowany i gotowy do odpalenia. Powstanie obfitowało w taktyczne majstersztyki, jak zajęcie Cytadeli, największego fortu w Poznaniu obsadzonego przez 900 niemieckich żołnierzy i odbitego przez jednego polskiego telegrafistę, Stanisława Jóźwiaka, w drodze pertraktacji i negocjacji. W wyniku bitwy o Ławicę zdobyto lotnisko i stojące na nim gotowe do startu samoloty. A w wyniku walki o Halę Zeppelinów na Winiarach pozyskano 300 rozłożonych na części samolotów bojowych i balony. Ogółem zdobyto sprzęt lotniczy warty 200 mln marek niemieckich. Powstanie miało swoich bohaterów, ale także bohaterki.

15 sekund. Mimo iż ukazało się ponad 3 tys. publikacji dotyczących powstania wielkopolskiego, nie jest ono utrwalone w świadomości narodowej jak inne powstania i nie cieszy się takim odbiciem w naszych narodowych wyobrażeniach historycznych.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Z dużym wzruszeniem staję dzisiaj na tej trybunie, popierając w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów i Konserwatyści idee powołania i projekt, który to materializuje, przedstawione przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, tym bardziej że został on przyjęty przez aklamację, co jest rzadkie w naszej Wysokiej Izbie. Sądzę, że najpierw jestem zobowiązany, wspominając związki rodzinne z powstaniem, bowiem rodzeństwo moich rodziców to też byli powstańcy, czworo braci. Ale przed wszystkim chcę dziękować inicjatorom ustanowienia tego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, którymi są Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja Zakłady Kórnickie, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz sygnatariusze licznie podpisani pod tym apelem, który został skierowany do prezydenta Rzeczypospolitej, marszałków Sejmu i Senatu, do nas jako parlamentarzystów oraz premiera rządu Rzeczypospolitej.

I ona mówiła: Apeluję do ciebie, abyś w tej sprawie, jak tylko sprawa stanie na porządku, żebyś głosował za ustanowieniem tego dnia. Więc wtedy mogłem jej odpowiedzieć, że będę zabierał głos, bowiem wielokrotnie miałem okazję być i w Środzie, i w wielu innych miejscach w Wielkopolsce, łącznie z rodzinnym Ostrzeszowem, na obchodach dnia wybuchu powstania wielkopolskiego. Te daty są różne w różnych miejscach Wielkopolski. Bo w Poznaniu to 27 grudnia, ale w niektórych miejscach to był 6 stycznia, czyli dzień Trzech Króli i to jest też data wybuchu powstania, bo tak się rozwijało pod względem militarnym, ale również pod względem możliwości. Wiele odcinków jest z tego powstania wspominanych. Najbardziej znane są oczywiście te wydarzenia, które miały miejsce w centrum, w Poznaniu, i te, które miały miejsce na froncie kujawskim.

Ale też było wielu przedstawicieli z innych regionów, np. Ślązaków biorących udział w tym powstaniu.

Wszyscy oni zgromadzili się między 3 a 5 grudnia w sali kina Apollo w Poznaniu po uroczystej mszy świętej, aby niejako apelować do wszystkich tych, którzy mogą w tej materii pomóc, aby Wielkopolska i inne wymienione dzielnice stały się integralną częścią niepodległego państwa polskiego. To było ogromne wydarzenie. To jest mało znany fakt. W tym 129 kobiet było posłami tego Sejmu. To jest też ważny fakt. Chcę podkreślić ogromną rolę nie tylko żołnierzy, którzy brali udział w powstaniu, ale również kobiet wielkopolskich. Przecież te nie tylko baretki, ale mundury, ale również nakrycia głowy - to wszystko było szyte przez wielkopolskie kobiety. Jak to zrobili, że 40 prawie tys. ludzi zostało umundurowanych w tamtym czasie? To był wielki zbrojny czyn. Nie byłoby to możliwe z punktu widzenia wojskowego, powiedział to prof. Pilarczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, historyk wojskowości. Z militarnego punktu widzenia powstanie wielkopolskie nie miało szans, ale miało solidną podstawę społeczną, solidną podbudowę. Sukces zapewniła dobra organizacja zrywu, wysoka organizacja, samoorganizacja społeczeństwa. Każdy mógł się włączyć (Dzwonek), działając w czytelniach i bankach ludowych, kółkach rolniczych i kółkach włościańskich, towarzystwach śpiewaczych i gimnastycznych. Ale jednocześnie wiemy, że to przygotowanie trwało przez okres, który nazywamy najdłuższą wojną nowoczesnej Europy. To był wielki czyn pracy organicznej, który przerodził się później w czyn zbrojny Wielkopolan. Przypomnę chociażby, że w samym Ostrowie Wielkopolskim było 30 towarzystw śpiewaczych. Popatrzmy na współczesną geografię naszych inicjatyw kulturalnych w różnych miejscach. W Towarzystwie Czytelni Ludowych w mojej miejscowości w 13 r. na odczyt poświęcony twórczości Sienkiewicza przyszło 250 osób. To świadczyło o budowaniu ducha polskiego wśród wszystkich stanów, które wzięły udział w tym zwycięskim powstaniu. Dziękuję prezydentowi Rzeczypospolitej, że podjął tą inicjatywę, a my możemy w dniu dzisiejszym wypowiadać się w tej sprawie i głosować w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Koła nr 5 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Zielonej Górze jestem zaszczycony, że mogę w tej kwestii przemawiać. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. na ziemiach Prowincji Poznańskiej. Było to jedno z bardzo niewielu polskich powstań narodowych, które zakończyło się tak znaczącym sukcesem.

Miał rację Roman Dmowski, kiedy mówił: Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. Powstanie wielkopolskie wybuchło po wizycie Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Było wyrazem słusznego gniewu Polaków wobec niemieckich agresorów. Polacy z Poznańskiego zachowali w sobie tożsamość narodową mimo dekad germanizacji, kulturkampfu, hakatyzmu i prześladowań. Nie pozwolili na odarcie się z polskości, wynarodowienie, zniemczenie. Są przykładem tak bardzo potrzebnym także dzisiaj, gdyż niektórzy starają się tożsamość narodową rozmyć w tożsamości europejskiej, regionalnej czy jakiejkolwiek innej. Nie byłoby sukcesu powstania wielkopolskiego, gdyby nie niezłomny duch narodowy Wielkopolan. Duch ten powstał przy udziale Narodowej Demokracji, która była najsilniejszym obozem ideowym w Wielkopolsce. Roman Dmowski, który stał na czele Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, zapewniał stałe poparcie dyplomatyczne dla sprawy polskiej w Wielkopolsce. O endeckiej podbudowie powstania wielkopolskiego świadczą chociażby słowa jego dowódcy, gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, który w swych wspomnieniach napisał: uważam się za nacjonalistę i narodowca. Na terenie Wielkopolski 1 czerwca 1919 r. odbyły się wybory uzupełniające do Sejmu ustawodawczego. Wspólna lista Narodowej Demokracji i innych stronnictw prawicowych uzyskała 97% poparcia i wszystkie 42 mandaty w Sejmie przeznaczone dla Wielkopolski. Powstanie wielkopolskie jest przykładem niezłomnego ducha narodowego, przykładem cnoty wojskowej oraz jedną z najpiękniejszych kart w historii Polski. Konfederacja oczywiście popiera należyte upamiętnienie powstańców wielkopolskich. Proszę, pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Wielkopolanie dobrze znają historię wybuchu powstania - przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego, jego entuzjastyczne przyjęcie w Poznaniu, wywieszanie polskich flag, potem gniew Niemców i pierwsze strzały. Do końca roku Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski. Musimy podkreślić, że u podstaw sukcesu powstania wielkopolskiego leżała przede wszystkim ogromna praca wykonana przez całe polskie społeczeństwo jeszcze pod zaborami. To w Wielkopolsce mieliśmy wówczas do czynienia z naprawdę dobrze kształtującym się nowoczesnym, świadomym społeczeństwem, które, co najważniejsze, nie było skonfliktowane. Wypracowane przez Wielkopolan idee pracy organicznej stały się dobrym fundamentem do prowadzenia prac nad organizacją powstania, wpłynęły na sposób jego zorganizowania, a potem zagospodarowania niepodległości po jej odzyskaniu. Wielu moich przedmówców podkreślało to w swoich wystąpieniach, bo to faktycznie leży u podstaw sukcesu powstania wielkopolskiego.

Niejednokrotnie padało pytanie, dlaczego powstanie nie zyskało dotąd należytego miejsca w literaturze, sztuce, malarstwie czy filmie.

Zasługi powstańców wielkopolskich są ogromne i nie ograniczają się wyłącznie do czasów zwycięskiej insurekcji. Ich rola w odbudowie ojczyzny odradzającej się po czasach zaborów jest bezcenna.

Dlatego upowszechnianie wiedzy o nim wymaga intensywnej pracy, poszukiwania atrakcyjnych nowych form przekazu i sprzyjających temu okazji.

W imieniu Wielkopolan, ale także swoich przodków - jestem prawnuczką powstańca wielkopolskiego - proszę państwa o poparcie tej inicjatywy i szerzenie wiedzy i pamięci o powstańcach wielkopolskich. Pani poseł Iwona Michałek, Porozumienie. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Historia narodu polskiego to niespotykana sinusoida chwil podniosłych i smutnych, wzlotów i upadków. Moment utraty przez I Rzeczpospolitą niepodległości to wielka rana na naszej narodowej duszy, niemniej moment odzyskania niepodległości i powstanie II Rzeczypospolitej to już wydarzenie pełne szczęścia i dumy. A ta nie została nam dana na tacy.

Jednak jej kształt mimo końca Wielkiej Wojny dalej zależał od siły oręża i od Polaków. Nasza historia jest pełna insurekcji i powstań, które mimo szlachetnych pobudek i zaangażowania wielu miały dla nas gorzki smak porażki. Powstanie wielkopolskie zajmuje jednak szczególne miejsce w naszej historii. Jest to zryw, który był dobrze przeprowadzony, skutecznie dowodzony i zakończył się naszym pełnym sukcesem. Z tego względu powstanie wielkopolskie zasługuje na szczególne upamiętnienie.

Wielkie uznanie oczywiście należy się Ignacemu Janowi Paderewskiemu, wybitnemu kompozytorowi, który swoim przyjazdem do Wielkopolski dał impuls do

Bardzo dziękujemy panu prezydentowi za to, że podjął taką inicjatywę.

Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Pytanie pierwsze zadaje pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście inicjatywa ustawodawcza zgłoszona przez pana prezydenta, dotycząca ustanowienia święta państwowego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest jak najbardziej słuszna.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wielkopolanie od dziesiątków lat w trakcie zaborów przygotowywali się do tego zrywu. Skuteczne przeciwdziałanie germanizacji, obrona Kościoła katolickiego i wiary, które stanowiły ostoję polskości, przeciwstawianie się działaniom Hakaty i Kulturkampfu, kult pracy organicznej, pozytywistyczne podejście do gospodarki, tworzenie polskich banków, spółdzielni i stowarzyszeń i budowanie dobrych relacji między poszczególnymi stanami, mieszczanami, chłopami i duchowieństwem (Dzwonek) - to dało początek ukształtowaniu się nowoczesnego i świadomego społeczeństwa, co z kolei stanowiło solidne podstawy do przygotowania i przeprowadzenia powstania wielkopolskiego. Oddając hołd kolejnym pokoleniom Wielkopolan, jestem przekonany, że celebrowanie kolejnych rocznic wybuchu zwycięskiego powstania będzie także doskonałym momentem do podkreślenia właśnie tych cech: otwartości, pracowitości, pragmatyzmu i w końcu odwagi w miłości do małej i wielkiej ojczyzny. Pani poseł Maria Małgorzata Janyska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z ogromną radością pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy propagowali i propagują pamięć o zwycięskim powstaniu wielkopolskim, ale chciałabym tutaj wyróżnić parę osób.

Pragnę także wyrazić wdzięczność wszystkim samorządowcom, którzy podjęli uchwałę z wnioskiem do prezydenta o ustanowienie tego święta, na czele z Jackiem Gurszem, szefem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, burmistrzem Chodzieży.

Wykonały ogrom pracy, szukając informacji właśnie o kobietach, które były do tej pory historii nieznane. Cieszę się również, że mogłam wesprzeć tę inicjatywę w tamtym czasie. Oddaję hołd wszystkim powstańcom i ich rodzinom, które w każdym miejscu Wielkopolski dbają o to, aby ta pamięć cały czas trwała. I na koniec jeszcze, proszę państwa, trochę prywatnej wdzięczności. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Niewiele jest dni w polskim parlamencie, kiedy tak zgodnie rozmawiamy i z dumą wspominamy tak ważny moment, jakim było powstanie wielkopolskie, i tak wielki sukces. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy od wielu lat kultywują pamięć o tych osobach, o tych miejscach. Tak jak mój kolega Grupiński wspomniał - pochodzimy z jednego miasta, z Wronek w Wielkopolsce, też jestem rodowitym Wielkopolaninem. Szanowni państwo, to wydarzenie było bardzo ważne dla mnie również osobiście jako wnuka ostatniego powstańca wielkopolskiego, który dożył prawie 106 lat - por. Jana Rzepy.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Kurzawa, Koalicja Polska. Dziękuję serdecznie. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Grzybowi za to, że upomniał się również o bardzo ważny kujawski epizod powstania wielkopolskiego. To bardzo ważne epizody związane z wyzwoleniem Mogilna, Strzelna, Kruszwicy, Inowrocławia, bitwa pod Rynarzewem, bitwa o Szubin, Żnin, Barcin, Nakło. Powstańcy także podeszli pod Bydgoszcz, która była wtedy zbyt silna, aby ją zdobywać. Jestem z tego niezmiernie dumny, że dzisiaj ta ustawa jest procedowana w Sejmie. Ale chciałbym zapytać o jedną bardzo ważną sprawę: Jakie działania zostaną podjęte, aby utrwalić w świadomości Polaków, w świadomości także tych młodych, wszystkie wydarzenia związane z powstaniem wielkopolskim (Dzwonek), aby powstanie wielkopolskie na trwałe znalazło się w świadomości Polaków i było przedmiotem dumy Polaków? Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Historia nie musi dzielić. Powstanie wielkopolskie jest naszą dumą. Ostatnie 4 dni grudnia 1918 r. w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim to chwile, gdy powstańcy wyzwolili instytucje publiczne, zdobyli koszary przy ul. Wrzesińskiej, zorganizowali oddział powstańczy, wzmocniony powstańcami z Wrześni, z Kłecka, który uczestniczył w potyczce z Niemcami pod Zdziechową. Ta bitwa pod Zdziechową odbiła się szerokim echem również w Berlinie. To powstanie ma wielu bohaterów. Jednym z tych bohaterów jest kpt. Paweł Cyms, urodzony w Pawłowie, gmina Czerniejewo. To właśnie z Gniezna na Kujawy ten dowódca prowadził powstanie wielkopolskie.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Na wstępie wielkie podziękowania dla pana prezydenta Andrzeja Dudy za to, że zjednoczył jako głowa państwa tak wiele środowisk, o których słyszeliśmy, i wprowadził projekt tej ustawy pod obrady Sejmu. Nareszcie, chciałoby się powiedzieć, dobrze, że jest taki prezydent, który po 32 latach od przemian w 1989 r. taką ustawę wprowadza, bo Wielkopolska na to zasługuje, tradycje powstania wielkopolskiego jak najbardziej na to zasługują, aby być wzorem i inspiracją dla całej naszej ojczyzny. Szanowni państwo, to bardzo ważne, że walczymy o ogólnonarodowe obchody rocznicy i przebiegu powstania wielkopolskiego, pamięć o powstańcach. Pamiętajmy także, że cała idea powstania wielkopolskiego to okres zaborów (Dzwonek), pracy organicznej, pracy u podstaw, wychowania młodzieży, pracy gospodarczej i właśnie realizowania myśli narodowej, realizowania konsekwentnie wychowania młodzieży, dbania o kulturę zgodnie z polską myślą narodową. To zwycięskie powstanie - sama nazwa w ustawie podkreśla sformułowanie: zwycięskie - niech będzie lekcją i inspiracją dla nas wszystkich, dla Polaków w całym kraju. Wielkie podziękowania dla pana prezydenta Andrzeja Dudy.

Pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jako poznaniak bardzo się cieszę, że powstanie wielkopolskie nareszcie zostało dostrzeżone, a prezydent spełnił postulat wielu Wielkopolan i Wielkopolanek. Upamiętnianie naszej historii nie może być ciągłym powracaniem do porażek i martyrologii. Musimy pamiętać, że były też momenty, gdy praca organiczna i silne społeczeństwo obywatelskie przynosiły zwycięstwo. Ten sukces nie był zasługą tylko karabinów i bitew, ale też przede wszystkim silnej lokalnej tożsamości i współpracy. Wiele osiągnięto dzięki doskonałej organizacji i negocjacjom, które powstańcy prowadzili z Niemcami. W ten sposób zdobyto chociażby pierwszego dnia powstania komendy policji, a w kolejnych dniach wiele innych ważnych budynków w centrum Poznania. Warto zapamiętać tę lekcję z powstania wielkopolskiego. Praca u podstaw (Dzwonek), edukacja i współpraca długofalowo są skuteczniejsze niż jakakolwiek broń. Wysoka Izbo! Chciałbym tylko przypomnieć, że w wyniku powstania wielkopolskiego wolność uzyskały Mogilno, Strzelno, Kruszwica, Żnin, Barcin.

Przy współudziale mieszkańców zajęto Rynarzewo oraz Brzozę. W Bydgoszczy działał szpital powstańczy, którym kierował m.in. dr Jan Biziel.

Chciałbym z tego miejsca w imieniu mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz w imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu prezydentowi za podjęcie tej inicjatywy ustanowienia takiego dnia, natomiast apeluję, że gdyby to można nazwać świętem, byłoby chyba znacznie lepiej. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Piotr Nowak, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To piękny dzień, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Ileż w nas, Wielkopolanach, jest w tej chwili dumy i światła, które dało nam to zwycięstwo. Oto bardzo pragmatyczna, oto taka bardzo pozytywistyczna Wielkopolska nagle w końcu grudniowych dni 1918 r. nabrała bardzo romantycznego wymiaru, wymiaru tak charakterystycznego dla całej Polski, tej kongresowej Polski. Ale w tej kongresowej Polsce ten romantyzm wiązał się z klęską, a tu romantyzm stał się zwycięski i dał taką przepustkę właśnie dla tego pozytywizmu, dla tego racjonalnego działania, racjonalnego działania zwycięskiego, racjonalnego również w powstaniu. Chwała bohaterom! Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! My mamy to wpisane w nasze DNA. Ale myślę, że tego dnia by nie było, gdyby nie fantastyczna postawa wielu samorządowców. 27 grudnia praktycznie w każdym miejscu, w każdym mieście, nie tylko w miastach wielkopolskich, te obchody są realizowane w sposób naprawdę godny.

Gdyby nie Wielkopolanie, mogło być różnie. Bardzo proszę, pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jako Wielkopolanin z urodzenia i wnuk powstańca wielkopolskiego Stefana Wilczyńskiego, który spoczywa w Poznaniu na cmentarzu na Miłostowie, chciałbym ze wzruszeniem wyrazić radość z faktu, że dzień powstania wielkopolskiego staje się świętem państwowym. To spora radość i satysfakcja obywatelska dla nas wszystkich.

To pytanie stawiam panu prezydentowi: Czy zamierza pan również zadbać o status dnia 4 czerwca? Wysoka Izbo! Dziękuję wszystkim tym Wielkopolankom i Wielkopolanom, wszystkim ambasadorom czczenia tego dnia, upamiętniania tego dnia każdego roku.

Były dni powstania wielkopolskiego, dni Wielkopolski. Bardzo serdecznie dziękuję, panie marszałku.

Tam znajduje się grób gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, nad którym trzymaliśmy wielką pieczę. Tam zostały przeniesione prochy jego córki, która zginęła w Katyniu.

Wielce Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Święto powstania wielkopolskiego to chluba dla Polski. To chluba dla całej Polski. Dla nas wszystkich Polaków, nieważne, gdzie mieszkamy. Ustanawiając to święto, powinniśmy być razem. Takie okoliczności jak święto ważne dla Wielkopolski, ważne dla Polski powinno nas łączyć. Przyjmijmy wszyscy to postanowienie o ustanowieniu święta powstania wielkopolskiego jako wspólną ważną decyzję przed kolejnymi decyzjami, aby waśnie w narodzie nie istniały. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Chciałam powiedzieć, że od wielu lat prowadzę obrady w Sejmie i nie pamiętam tak spokojnej, tak ciekawej, tak merytorycznej i tak pozytywnej debaty, za którą chciałam wszystkim państwu bardzo podziękować. Chciałam także przypomnieć bardzo stary serial, który opracowywał pan Stefan Bratkowski, a reżyserował pan Sztwiertnia „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” Pokazano, jak należy wspólnie działać. Wszystkim państwu bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszą debatę dziękuję i mam nadzieję, że to taki nowy początek debat historycznych w Sejmie. Bardzo dziękuję.

Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1616 i 1615. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w łącznej dyskusji nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedłożył wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na przedłużenie na okres 60 dni stanu wyjątkowego obowiązującego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, druk nr 1617. W związku z tym, na podstawie art. 117a ust. 2 regulaminu Sejmu, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tym przypadku Sejm wysłuchał 7-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Uprzejmie proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, druk nr 1509, a sprawozdanie to druk nr 1601. Sejm na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Procedowana ustawa stanowi dopełnienie dotychczasowej polityki prorodzinnej i jest kolejnym elementem budowanego spójnego systemu wsparcia i rozwoju polskich rodzin, który od lat jest realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Celem projektu ustawy jest przede wszystkim łagodzenie niekorzystnych trendów demograficznych, redukcja wskaźnika ubóstwa rodzin z dziećmi na utrzymaniu, inwestycja w rodzinę, wzmacnianie społecznego kapitału ludzkiego, wzmocnienie instrumentów umożliwiających łączenie rodzicielstwa z zatrudnieniem i rozwój szeroko pojmowanych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Najważniejsze rozwiązania zawarte w przedkładanym projekcie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Zostaje wprowadzone nowe świadczenie kierowane do rodzin z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe, a środki nie będą opodatkowane. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc. Miesięczna wysokość wsparcia wyniesie 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł przez rok, w zależności od tego, jak będą chcieli rodzice, jaką złożą deklarację. Prawo do wsparcia będzie przysługiwać także rodzinom, które będą posiadały drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w dniu wejścia w życie ustawy.

Zadanie będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 r. ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 600 tys. dzieci. Dodatkowym elementem i rozwiązaniem w ustawie będzie wzmocnienie systemu opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Będzie wprowadzone dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Jednocześnie koło Polska 2050 zgłosiło dwa wnioski mniejszości. Wysoka Izbo! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu tego projektu ustawy wnosi do Wysokiej Izby o uchwalenie procedowanego projektu ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Teresa Wargocka. Zapraszam, pani poseł. Pani Minister! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym i sprawozdania dotyczącego tego projektu, druk nr 1601. Wysoka Izbo! W ostatnich 5 latach, co mogę stwierdzić z pełną satysfakcją, sytuacja materialna rodzin, status materialny rodziny uległ zdecydowanej poprawie.

Wielki pakiet, który realizujemy od 5 lat, czyli program 500+, program „Dobry start”, wsparł rodziny wychowujące dzieci. Jest to niekwestionowany sukces ze strony wysiłku finansowego państwa, ale przede wszystkim wielki sukces rodzin, dzieci, ponieważ to zdecydowanie wpłynęło na rozwój młodego pokolenia.

Otrzymali to wsparcie również młodzi ludzie, którzy podejmują przeważnie swoją pierwszą pracę bądź studiują i pracują na swoje własne utrzymanie. Zwolniliśmy tych młodych ludzi do 26. roku życia z podatku dochodowego. Dochód rozporządzalny w polskiej rodzinie w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł o kilkadziesiąt procent. Dzisiaj rozmawiamy o kolejnym segmencie wsparcia polskich rodzin. Widzimy lukę, która powstała w systemie wsparcia rodzin wychowujących dzieci pomiędzy ukończeniem 1. roku życia a tym wiekiem, kiedy dziecko może zostać przyjęte do przedszkola. To jest ogromnie ważny moment, ponieważ zazwyczaj w tym momencie, kiedy rodzą się pierwsze i kolejne dzieci, załamuje się również to, co jest ambicją i marzeniem wielu kobiet, czyli możliwość połączenia pracy zawodowej z wychowaniem dziecka. W strategii demograficznej opracowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej bardzo wyraźnie zobaczyliśmy te bariery, które powstrzymują młodych ludzi przed tym, żeby zdecydować się na pierwsze bądź kolejne dziecko.

Grozi nam wyludnienie. Grozi nam starzenie się społeczeństwa. To pułapka demograficzna, która może przynieść bardzo negatywne skutki.

Są wykształcone, ambitne. Można powiedzieć - w takim potocznym znaczeniu - nowoczesne i ten kapitał opiekuńczy daje im takie możliwości. Kolejne bardzo duże pieniądze są na organizację opieki żłobkowej.

liczby posiadanych dzieci.

Ustaliliśmy w komisji, że jest zbieżność dwóch ustaw, nad którymi równolegle procedujemy w Sejmie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Projekty, które dotyczą wsparcia rodzin, szczególnie łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, są zawsze bardzo ważne.

Przedwczoraj na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny chcieliśmy zadać pytania dotyczące poszczególnych artykułów, ale niestety nie było to do końca możliwe, więc dzisiaj wykorzystam drugie czytanie do zadania konkretnych pytań czy też wyjaśnienia poprawek.

7 lutego 2018 r. na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zamieszczona została informacja, że program „Rodzina 500+” jest sprawnie realizowany przy dobrej współpracy z samorządami.

Przecież państwo, podejmując decyzję, żeby płatnikiem był samorząd, również dokonaliście pewnych inwestycji, nakładów finansowych.

Inwestujecie najpierw w samorząd, później przenosicie to do ZUS-u, dlatego składamy taką poprawkę, aby płatnikiem był ZUS. Druga poprawka dotyczy rodzin dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Mam mało czasu, więc niestety muszę iść dalej. Kolejna, trzecia poprawka. Chodzi o to, żeby pieniądze przysługiwały również na pierwsze dziecko. Tak było w przypadku 500+, tak jest teraz.

Kolejna poprawka, czwarta.

Nie rozumiem, po co zabraliście, a teraz dajecie. Jeszcze jedna poprawka, piąta. Chodzi o sposób, w jaki zlecacie to zadanie: bez przetargu, bez respektowania ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przynajmniej moglibyście państwo posłuchać legislatora, który na posiedzeniu komisji powiedział tak: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2014 r. w sprawie zamówień publicznych określa zamknięty katalog wyłączeń. Stosowanie jej przepisów i tym samym każdy przypadek wyłączenia stosowania przepisów wprowadzany w polskim systemie prawa powinny być oceniane pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej. I tu trzeba mieć na względzie taką uwagę, takie zastrzeżenie, że to może być naruszenie przepisów prawa unijnego. Skoro Polski Ład i to rozwiązanie, bardzo dobre, były ogłoszone w maju, to trzeba było nad tym projektem procedować wcześniej, a nie we wrześniu. I ostatnia poprawka - myślę, że zdążę, pani marszałek - poprawka szósta. To fajnie, że dążymy wszyscy do cyfryzacji, do automatyzacji, do elektronizacji. Wszystko dobrze, ale jednak nie możecie (Dzwonek) państwo nie widzieć 4,5 mln ludzi, którzy nigdy nie korzystali z Internetu. Chociaż przez rok dajcie możliwość tym wykluczonym cyfrowo złożenia wniosków w formie papierowej. Sześć poprawek.

Dotyczą one przede wszystkim tego, żeby dzieci w pieczy zastępczej też mogły otrzymywać rodzinny kapitał opiekuńczy, ale także abyśmy zastanowili się nad tym, żeby w rodzinach, w których jest dziecko z niepełnosprawnością, ten rodzinny kapitał opiekuńczy przysługiwał na pierwsze dziecko od urodzenia. To jest oczywiście związane z tą sytuacją rodzinną, z sytuacją zdrowotną, ale tak naprawdę to dotyczy też sytuacji w ochronie zdrowia, tego, jak długo czeka się na specjalistów, jak bardzo kosztowne są wizyty u lekarzy, szczególnie w czasie kiedy poszukuje się jeszcze diagnozy bądź kiedy ta diagnoza zapada i potrzebna jest np. rehabilitacja.

Składam więc poprawki.

Chciałabym dzisiaj w ramach drugiego czytania przytoczyć uwagi do projektu opublikowane przez Katarzynę Roszewską, profesor z wydziału prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współtwórczynię Centrum Badań nad Niepełnosprawnością, głównie dlatego, że są one zgodne z tym, o czym mówiłam podczas pierwszego czytania, a także z tymi uwagami, które prezentowałam w czasie posiedzenia komisji. Przede wszystkim piszecie, w projekcie wskazuje się, iż celem kapitału jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wiemy, że jest to pewnego rodzaju określenie, które wprowadza w błąd, ponieważ dotyczy tylko sytuacji, gdy w rodzinie jest drugie i kolejne dziecko, a głównym celem nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych każdego dziecka, lecz pewnego rodzaju premia za urodzenie lub wychowanie kolejnego dziecka, co potwierdzacie na str. 12 uzasadnienia projektu ustawy. Jest to do pewnego stopnia powielanie też pierwotnej koncepcji świadczenia wychowawczego, które przysługiwało na kolejne dziecko. Na pierwsze tylko po spełnieniu kryterium dochodowego, ale spotkało się to z krytyką i doprowadziło to faktycznie do zmiany. Na marginesie też warto wykazać, że świadczenie wychowawcze 500+, a nie kapitał, pełniej realizuje cel częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Problem dzietności, który w istocie jest celem ustawy, związany jest nie tylko z niższym wskaźnikiem dzietności, a jego poprawa nie jest uzależniona wyłącznie od transferów socjalnych. Niestety nie wystarczy dać, żeby rodziło się więcej dzieci. Wskaźnik dzietności wzrósł jeszcze przed wprowadzeniem świadczenia wychowawczego, co też pokazuje, że wasze świadczenie wychowawcze również nie było skuteczne, jeśli chodzi o problem demografii. Utrzymująca się jednak niska dzietność wynika przede wszystkim ze zmniejszenia się populacji kobiet w wieku adekwatnym do posiadania dzieci, to jest echo spadku urodzeń, począwszy od okresu transformacji ustrojowej, oraz z odraczania decyzji o urodzeniu pierwszego dziecku. Ciągle wzrasta ten średni wiek kobiet decydujących się na urodzenie pierwszego dziecka i strona społeczna w toku konsultacji projektów wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność oddziaływania właśnie na ten wskaźnik, czyli na decyzję o posiadaniu pierwszego, a nie kolejnego dziecka. Powinniście więc dążyć do skutecznego projektowania ustaw, do poprawy dzietności może nie poprzez nagradzanie tylko przez innego rodzaju działania, które skłaniałyby kobiety do tego, żeby wcześniej rodzić pierwsze dzieci. Przede wszystkim cieszy mnie oczywiście to, że dzisiaj odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i będziemy omawiać projekt dotyczący tzw. matek z EWK, bo o tym też mówiłam przy pierwszym czytaniu, punktując boleśnie niestety politykę społeczną Prawa i Sprawiedliwości. Na tym naprawdę nam bardzo zależy. Czyli dobra, skuteczna polityka społeczna, która ukierunkowana jest na osoby z niepełnosprawnościami, na ich rodziny, bo to pokazuje tak naprawdę siłę państwa. Dobra polityka społeczna nie zostawia nikogo poza marginesem i tak naprawdę dba o wszystkich. Wracam więc do tego jeszcze raz, odnosząc się do naszej poprawki, i proszę o zastanowienie się, czy nie byłoby dobrym pomysłem, żeby rodzinny kapitał opiekuńczy został poszerzony o rodziny osób z niepełnosprawnościami, gdzie często jest tylko jedno dziecko, tym bardziej że nie dajecie rodzicom prawa wyboru.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Jest tylko jeden problem: poprawka została złożona nieformalnie. Dziękuję bardzo. Może rozpocznę od tego, na czym zakończyła moja przedmówczyni pani posłanka Kotula. Rzeczywiście postanowiliśmy zgłosić poprawkę, która dotyczy rozszerzenia tego programu na pierwsze dziecko, jeśli jest to dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

Pani marszałek, przekazuję tę poprawkę. Dziękuję bardzo.

Polityka społeczna wymaga zupełnie innych narzędzi.

To są te najważniejsze rzeczy i ich cały czas brakuje.

Jeśli mówimy o usłudze publicznej najwyższej jakości, to mówimy o opiece wczesnodziecięcej, już w żłobku, w przedszkolu, na najwyższym poziomie.

Niestety mamy głębokie przekonanie, że ten przetarg jest już rozstrzygnięty, mimo że nie miał prawa być. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Ma to wypełnić lukę pomiędzy zakończeniem urlopu macierzyńskiego a objęciem dziecka opieką przedszkolną i wesprzeć finansowo rodziców w zakresie zorganizowania opieki nad dzieckiem.

Przede wszystkim bezpieczeństwo: bezpieczeństwo i pewność jutra, bezpieczeństwo pracy, ale także całego otoczenia, które jest związane z rodziną. Państwo mówicie o żłobkach, przedszkolach.

Niestety poprzez taką instytucję, jaką jest ZUS, która oczywiście pełni całkowicie inną funkcję. Tak, wiemy, jaką funkcję.

Dlatego też Polskie Stronnictwo Ludowe, szanowni państwo, wesprze tę inicjatywę, zagłosujemy za tym projektem.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Minister! Wysoka Izbo! Porozumienie zawsze będzie popierało wszystkie dobre rozwiązania, które będą służyć polskiej rodzinie i polskim dzieciom. Omawiany projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia. Przysługujące 12 tys. na dziecko ma być wypłacane w ratach miesięcznych. Chcę zwrócić uwagę na to, że projektodawcy postawili sobie bardzo ambitne cele.

Te cele są, jak już powiedziałam, ambitne i mam nadzieję, że zostaną spełnione.

Trzeba nad nią jeszcze pracować, ale Porozumienie wspiera i będzie popierało te rozwiązania prawne. Dziękuję bardzo. Pani poseł Agnieszka Ścigaj w imieniu koła Polskie Sprawy. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Chodzi tu też o pomoc w wychowaniu dzieci, w tym, żeby rzeczywiście polskie społeczeństwo nie podpadło pod te wskaźniki, o których mówiła pani poseł Wargocka. Jak najbardziej będziemy głosować za tą ustawą.

Szanowni państwo, zastanówmy się, czy takie elementy wrzucane w dobre ustawy nie psują po prostu państwa.

To może znaleźć i powinno znaleźć się w jednej uporządkowanej ustawie.

Ja też nie rozumiem tego lęku przed wsparciem pierwszego dziecka. Szanowni państwo, każde dziecko jest nam potrzebne, pierwsze też, tym bardziej że rzeczywiście wskaźniki dotyczące posiadania pierwszego dziecka są naprawdę niepokojące, bo to one nam zaniżają tę dzietność. Jeśli chodzi o cel dotyczący ubóstwa, też warto się zastanowić, patrząc na liczby i planując tu coś profesjonalnie, skoro 7% rodzin, które posiadają dwoje dzieci, żyje na granicy ubóstwa, już nie mówiąc o tym, że ten wskaźnik jest najwyższy w przypadku posiadania co najmniej jednego dziecka niepełnosprawnego (Dzwonek), 7,5%. Przechodzimy do pytań. Zamykam listę osób. Ależ oczywiście. Wyznaczam czas - 1 minuta. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Kapitał opiekuńczy to pomoc na drugie i kolejne dziecko. Jednak eksperci alarmują, że projekt zupełnie pomija rodziny, które znajdują się w dramatycznej sytuacji, a ta propozycja jeszcze bardziej wypycha ich na margines życia społecznego. Jak pokazują dane GUS, skrajne ubóstwo wśród małżeństw z dwójką dzieci wyniosło w 2020 r. 2,7%, a wśród gospodarstw domowych z jednym dzieckiem niepełnosprawnym aż 7%, zaś w rodzinach z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną nawet 7,5%. Koszty związane z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością są o wiele wyższe, dlatego wiele rodzin, w których chore dziecko rodzi się jako pierwsze, nie decyduje się na kolejne dziecko. Kapitał opiekuńczy dodatkowo ma pomóc w łączeniu wychowywania dzieci z pracą zawodową. Tymczasem w przypadku rodzin, w których są niepełnosprawne dzieci (Dzwonek), obecne przepisy wymuszają wybór: praca albo pomoc. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na s. 5 uzasadnienia czytam, że środki będą stanowiły impuls powstrzymujący odpływ z rynku pracy, w szczególności matek niepodejmujących lub przerywających zatrudnienie ze względu na ograniczony dostęp do instytucji opieki nad dziećmi. I to jest de facto przyznanie się rządu Prawa i Sprawiedliwości do porażki w tworzeniu warunków do wychowywania dzieci. Mówiłem o tym podczas omawiania ustawy 500+, że takie ukształtowanie programu spowoduje odpływ matek z rynku pracy. że opieka nad dziećmi leży, że edukacja leży, że tym trzeba się zająć. Wtedy też posłanki Prawa i Sprawiedliwości krzyczały, że to nieprawda. I dzisiaj przyznajecie się do błędu. Przez 6 lat PiS nie zrobił nic dobrego w tych najważniejszych sprawach, o których mówiłem. Teraz znów chcecie naprawiać te swoje błędy, dając kolejne środki.

Bardzo proszę. Pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł, zadać pytanie. Wysoka Izbo! Znów pomija się pierwsze dziecko, co dla wielu rodzin jest bardzo krzywdzące, bo jak mówią matki - tutaj cytuję - albo dotuje się wszystkich, albo nikogo i nawet gdyby rząd dał mi 50 tys., to nie skłonni mnie to do urodzenia kolejnych dzieci, bo dzieci ma się z miłości, a nie dla kolejnego programu politycznego. Rząd w swoich działaniach zawsze kogoś lub coś pomija. Oczywiście jak najbardziej jestem za tym programem, który wspiera rodziny w trudnej sytuacji finansowej, ale po raz kolejny sygnalizuję i proszę, abyście zajęli się problemem niań, których pomoc obecnie przysługuje od 20. tygodnia życia dziecka. Czy okres zaraz po urodzeniu i wyjściu ze szpitala nie jest dla rodziny bardziej trudny i wyczerpujący? Chcecie dać 12 tys. na drugie i kolejne dziecko, a nie chcecie pomóc matce (Dzwonek), która wraca zaraz po porodzie ze szpitala.

Pani poseł, przepraszam, trzymajmy się czasu. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! To ważny instrument wsparcia państwa, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, możliwość łączenia pracy zawodowej oraz systemowe wsparcie dla funkcjonowania instytucji opieki nad małym dzieckiem. Ten projekt przewiduje również możliwość wsparcia gmin w powoływaniu, budowaniu i funkcjonowaniu placówek takich jak żłobki czy kluby dziecięce. Do tej pory tylko w połowie polskich gmin funkcjonują właśnie te instytucje opieki nad małym dzieckiem. Ustawa przewiduje również trzy moduły pomocy dla samorządów.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Dyskusja klubowa pokazywała, że jest dosyć duża zgodność co do samego projektu ustawy. To świadczy o tym, że ta ustawa jest dobra dla Polaków. Obecna sytuacja demograficzna jest trudna. Utrzymujący się od 30 lat spadek dzietności powoduje wyludnianie się Polski. Dlatego aktywna polityka prorodzinna powinna łagodzić te tendencje. Pomoc kierowana do rodzin z dziećmi do 3 lat jest znaczącą pomocą dla rodzin, ale jest też znaczącą inwestycją w rodziny. Przecież rodzina jest podstawową komórką, czyli świadczy o dobrej kondycji państwa. Pytanie do pani minister: W jakim stopniu proponowane rozwiązania dotyczą dzieci.

Było to określone. Bardzo proszę.

Pani Minister! Wysoka Izbo! Intencje tej ustawy są dobre, idą w dobrym kierunku, natomiast ona wprowadza. Może inaczej: nie wprowadza systemowych rozwiązań. Natomiast te zapisy tyczą się znowuż dziecka drugiego, nie pierwszego. Rozumiem, że państwo nie chcecie pochylić się i wprowadzić tej ustawy dla rodzin z pierwszym dzieckiem, ale czy może - i tu poproszę panią minister o odpowiedź - jednak ministerstwo pokusiło się i dokonało wyliczeń, jak sytuacja wyglądałaby przy wprowadzeniu tych rozwiązań już od pierwszego dziecka? Jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne, myślę, z perspektywy rodzin, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością.

Nie ma. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Z prognoz Eurostatu wynika, że w ciągu najbliższej dekady populacja naszego kraju zmniejszy się o prawie 1 mln osób. Jest to w dużej mierze wasza zasługa. Procedowana ustawa ma być niejako odpowiedzią na to negatywne zjawisko. W jej uzasadnieniu postawiono dość śmiałą tezę, że wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego zachęci rodziców do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Rzeczywistość pokazała, że wasze socjalne zachęty wprowadzone w celu poprawy demografii nie odniosły spektakularnego sukcesu w tym zakresie, do czego nawet sami się przyznaliście. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie: Na jakiej podstawie stwierdzono, że w wyniku procedowanej ustawy nastąpi zwiększenie dzietności w Polsce? Czy posiadacie państwo odpowiednie wyliczenia potwierdzające prawdziwość tego stwierdzenia? Dlaczego nowego świadczenia nie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej? Wysoka Izbo! Programy socjalno-społeczne w pierwszej kolejności - wydaje mi się, że to jest logiczne - zawsze powinny być dedykowane i kierowane do ludzi i do rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej, społecznej czy rodzinnej.

Mam konkretne pytanie, bo tego w ogóle nie rozumiem.

Wysoka Izbo! Wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że rodzina to podstawa budowania społeczeństwa. Obecnie akcentowanym problemem jest demografia, malejąca dzietność rodzin. Dlatego aktywna polityka rodzinna powinna łagodzić negatywne trendy demograficzne i obejmować działania szczególnie w takich obszarach jak zdrowie, opieka nad dzieckiem czy też możliwość godzenia ról zawodowych i rodzinnych. Skuteczna realizacja takiej polityki wymaga działań skoordynowanych i długofalowych. Zapewnia je Polski Ład. Propozycja wprowadzenia rodzinnego kapitału opiekuńczego to czynnik finansowy, który ma zachęcić do posiadania dzieci, ale przede wszystkim środki, które pomogą w zapewnieniu opieki dla dziecka między 12. a 36. miesiącem życia właśnie w żłobku czy w instytucjach prowadzących taką formę opieki. To również kolejny element łączenia rodzicielstwa z pracą zawodową kobiet. To również znacząca pomoc finansowa w zapewnieniu i opłaceniu opieki nad dzieckiem dla matek, które wychowują kilkoro dzieci (Dzwonek), ale też możliwość realizacji inwestycji związanych z tworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3, jak również nowe miejsca pracy.

Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję, jako młody rodzic, za ten program. Rozmawiam z wieloma moimi rówieśnikami i ludźmi, którzy spodziewają się dzieci bądź mają większe rodziny i dzieci im się rodzą. Stąd też dziękuję za to, że te osoby również będą mogły być objęte tym programem.

Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Wysoka Izbo! Mamy najwyższą inflację od 20 lat. Realne podwyżki płac w okresie ostatnich 5 lat zostały pochłonięte przez inflację w zaledwie kilka miesięcy mijającego roku. Gdzie są zapewnienia o dostawach taniego gazu w obliczu kolejnych podwyżek? Co robi rząd w sytuacji, gdy ceny paliw zbliżają się do kolejnego rekordu? Czy rząd nie obawia się, że przy obecnym wzroście cen kapitał, o którym dzisiaj dyskutujemy, zostanie przejedzony w ciągu pierwszego roku życia dziecka? Wiem, że nie chcecie wprowadzić kapitału opiekuńczego na pierwsze dziecko. Apeluję do waszego sumienia, wprowadźcie ten kapitał dla pierwszego dziecka niepełnosprawnego. Wysoka Izbo! Można tego wysłuchiwać w nieskończoność. Dziękuję bardzo tym klubom opozycyjnym, które popierają tę ustawę. Strategia demograficzna 2040” przygotowana przez ministerstwo rodziny jest rewelacyjnym dokumentem. Warto się z nim zapoznać. To nie tylko kapitał opiekuńczy, lecz także mieszkanie bez wkładu własnego i reforma podatków.

Powstało wiele programów i doskonale o tym wiecie. Chodzi o pierwsze dziecko niepełnosprawne, które rodzi się w rodzinie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę. Państwa posłów proszę, żeby nie pokrzykiwać. Wysoka Izbo! Dzisiaj rozmawiamy o rządowym projekcie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, o środkach, które mają otrzymać rodziny. Jak rząd planuje rozwiązać problem wykluczenia cyfrowego tej grupy osób? Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Omawiany projekt jest kolejnym instrumentem wspierającym polską rodzinę. Poprawa wskaźników demograficznych jest wyzwaniem dla całej klasy politycznej. Cieszę się, że pojawiły się zapowiedzi poparcia dla tego projektu ze strony opozycji. Chciałabym, aby pani minister odpowiedziała na pytanie dotyczące opieki instytucjonalnej i jej dalszego rozwoju w świetle proponowanej ustawy. Jaką szansą dla mamy, która chce wrócić do pracy i dla babci, która chce być aktywna zawodowo, jest ten projekt? Czy obydwie panie będą mogły pogodzić swoje ambicje zawodowe?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Takiej katastrofy, jeżeli chodzi o demografię, jeszcze w Polsce nie było.

Polaków więcej niż się urodziło.

Szanowni państwo, przez 6 lat nie zrobiliście nic, a teraz chcecie wrócić do programu, który był realizowany przez rząd Platformy Obywatelskiej. Cena mieszkania. Dzięki programowi dopłaty do kredytów udało się zapewnić 340 tys. [[Dzwonek]] nowych mieszkań. Uprzejmie proszę o zadanie pytania. Pani Marszałek! Trudno się nie odnieść do wypowiedzi mojego poprzednika, bo właśnie pochwalił program mieszkaniowy Platformy Obywatelskiej. Z badań wynika, że najwięcej mieszkań kupiono w dużych miastach i są to kawalerki, a nie mieszkania dla rodzin. To były mieszkania dla bogatych.

Bo wracamy do dyskusji o 500+. Opozycja chciałaby więcej, a my musimy patrzeć na możliwości budżetowe, analizować program, wyciągać wnioski i zmieniać go dla dobra rodzin. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Katarzyna Kotula, klub Lewica. Bardzo proszę. Podczas kiedy Prawo i Sprawiedliwość z Platformą Obywatelską licytują się na to, kto co zrobił gorzej, ja chcę państwa zapewnić, że Lewica ma całościowy plan na dobrą i skuteczną politykę społeczną i na pewno nie zostawimy rodzin osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym chciałabym zapytać. Koleżanki przywoływały tutaj dane GUS-u a propos skrajnego ubóstwa: wśród małżeństw z dwójką dzieci - na poziomie 2,7%, wśród gospodarstw domowych z jednym dzieckiem niepełnosprawnym - aż 7%, zaś co najmniej z jedną osobą z niepełnosprawnością - 7,5%. Pomimo tych danych nie dokonano waloryzacji świadczeń rodzinnych w ostatnim terminie ich ustawowej weryfikacji, co najdotkliwiej odczuwane jest właśnie przez rodziny osób z niepełnosprawnościami. Następna taka weryfikacja nastąpi dopiero za kolejne 3 lata. Chciałabym zapytać przy okazji: dlaczego? Sytuacją społecznie niesprawiedliwą jest utrzymywanie na poziomie 215 zł zasiłku pielęgnacyjnego na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością (Dzwonek) do samodzielnej egzystencji. Pani minister, czy możemy dzisiaj usłyszeć jasną deklarację, kiedy wszystkie te obietnice dotyczące rodzin osób z niepełnosprawnościami zostaną spełnione? będzie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko, tymczasem w ich sytuacji nic się nie zmienia. Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wszelkie programy, które dotyczą wzrostu dzietności, wsparcia dla rodziny, zawsze będą miały moje poparcie. Po pierwsze, kobieta musi jasno wiedzieć, co ją czeka, jeśli decyduje się na urodzenie dziecka, ale również co ją czeka, kiedy zachodzi w ciążę, co ją czeka, jeśli chodzi o pracę, i jakie później będą wszelkie działania. Nie może być, po pierwsze, takiej sytuacji, że musi być wybór: albo rodzenie dzieci, albo praca. My musimy stworzyć taki system, który będzie dawał gwarancję, że jeśli kobieta decyduje się na urodzenie pierwszego, drugiego czy piątego dziecka, będzie bardzo mocno przy tym wspierana. na to się decyduje. Zapraszam, panie pośle. Pani Minister! Wysoka Izbo! Od 2015 r. nastąpił przełom w polityce społecznej w Polsce. Dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma świadomość, że nakłady, zwiększanie nakładów na rodzinę to przede wszystkim inwestycja. I dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym idziemy krok do przodu, inwestujemy dalej, bo wiemy, jak ważne jest dobro polskich rodzin. Szanowni państwo, niecały rok temu u boku pani minister miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu 100 miejsc żłobkowych w Wieluniu. Obok, w gminie wiejskiej Osjakowie, 25 miejsc żłobkowych. W najbliższą sobotę w imieniu pana wójta zapraszam panią minister do również małej wiejskiej gminy Galewice. Ale zapraszam także przedstawicieli opozycji, bo myślę, że jak zobaczą, to uwierzą. Ostatnie pytanie, pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Bardzo proszę. Szanowna pani poseł tutaj powiedziała, że zahamowaliście trend spadkowy. To nie jest prawda. Według danych GUS-u ostatnie miesiące to są miesiące rekordowych spadków właśnie, jeżeli chodzi o liczby urodzeń, to po pierwsze. Ja odpowiem, bo nie ma sensu ukrywać: Nie ma tego teraz na pierwsze dziecko, dlatego że zrobicie to najprawdopodobniej za 2 lata.

To jest oczywiste. Od połowy 2017 r., szanowni państwo, sukcesywnie spada liczba nowych urodzeń. 500+ to nie był żaden program demograficzny. RKO również nim nie jest. To jest program propagandowy, polityczny, którym chcecie kupić wyborców. Jeżeli chcecie poważnej polityki rodzinnej, obniżajcie podatki, dawajcie ludziom się wzbogacić (Dzwonek) normalnymi pieniędzmi. Proszę to powiedzieć rodzinom, które dzięki 500+ wyjechały po raz pierwszy na wakacje. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. O udzielenie odpowiedzi na pytania uprzejmie proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej panią minister Barbarę Sochę. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam, nie ukrywam, przyjemność odpowiedzieć na różne państwa opinie, pytania i komentarze dotyczące procedowanego projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Cieszę się, że państwo też widzicie potrzebę spójnego i strategicznego podejścia do tego tematu, jakim są wyzwania demograficzne, przed którymi stoimy.

Na tej sali też już wiele razy o tym rozmawialiśmy.

To jest dosyć oczywiste i myślę, że nie wymaga dalszych wyjaśnień. Jeśli chodzi o kapitał opiekuńczy, to jest to program, którego celem jest ułatwienie rodzicom podjęcia decyzji o drugim, kolejnym dziecku.

To nie są bariery związane z ceną żłobków czy ich dostępnością. Pierwszą i podstawową barierą związaną z urodzeniem pierwszego dziecka jest mieszkanie. Drugą bardzo ważną barierą związaną z urodzeniem pierwszego dziecka jest stabilna praca. Jeśli chodzi o problem mieszkaniowy, to następny punkt porządku obrad dotyczy właśnie zmian w polityce mieszkaniowej i właśnie te zmiany mają na celu likwidację m.in. właśnie tej bariery związanej z urodzeniem pierwszego dziecka. Jeśli chodzi o kwestie związane ze stabilną pracą, to przedstawiając strategię demograficzną wraz z panem premierem, z panią minister Maląg, w czerwcu tego roku przedstawiliśmy propozycję pakietu: elastyczna i stabilna praca. Bardzo intensywnie spotykam się z różnymi środowiskami, nie ukrywam, że głównie pracodawców, bo to od pracodawców bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o zatrudnianie, politykę zatrudniania i poczucie stabilności pracowników.

I to tyle, jeśli chodzi o pierwsze dziecko.

Nie dalej jak wczoraj miałam okazję przysłuchiwać się debacie nad ustawą podatkową, gdzie właśnie padł zarzut kompletnie odwrotny, czyli nie jedna ustawa, która ma 700 stron, ale właśnie po kawałku.

Jeśli chodzi o kwestie związane z tym, dlaczego ta ustawa dotyczy każdego drugiego, kolejnego dziecka, to padło tu takie zdanie, że jest to niezrozumiałe, bo powinniśmy wspierać tych, którzy są w trudnej sytuacji, którzy potrzebują, a nie tych, którzy mają duże dochody i mają dwoje lub troje dzieci. No właśnie nie, szanowni państwo.

I dlatego bardzo się cieszę, że program 500+ jest programem powszechnym, uniwersalnym, tzn. uniezależnionym od kryteriów dochodowych. Tak samo rodzinny kapitał opiekuńczy jest pozbawiony kryterium dochodowego, bo nie jest to program socjalny. To nie jest program, którego celem jest obniżenie ubóstwa w rodzinach w najtrudniejszej sytuacji.

Myślę, że każda kobieta, która przeżywa macierzyństwo, doskonale wie, o jakich dylematach mówimy.

Są kobiety w Polsce, które uważają, że rok to jest optymalny czas, ale są takie, które uważają, że 2 lub 3 lata to jest ten optymalny czas, który powinny poświęcić wyłącznie wychowaniu małych dzieci.

Wspieramy wszystkie formy rozwoju. Dlatego ten kapitał opiekuńczy służy też tym rodzicom, którzy nie decydują się na opiekę instytucjonalną. Mówiąc o opiece instytucjonalnej, chciałabym powiedzieć, że trochę w tej debacie nam umknęła bardzo ważna kwestia, że ten projekt, oprócz tego, że wprowadza rodzinny kapitał opiekuńczy, wprowadza również to, o co od jakiegoś czasu apelowały samorządy, czyli stały mechanizm finansowania, współfinansowania, utrzymania miejsc w opiece instytucjonalnej. Zgodnie z tymi zmianami każdy rodzic pierwszego dziecka, który będzie chciał skorzystać z opieki instytucjonalnej i wysłać dziecko do żłobka, otrzyma obniżenie opłaty żłobkowej o 400 zł.

Przypominam, w przypadku pierwszego dziecka, więc to nie jest tak, że pierwsze dzieci na tym nie korzystają.

Właśnie dlatego wprowadziliśmy zmiany w programie 500+, żeby zaoszczędzić spore środki, które były do tej pory przeznaczane na obsługę, na realizację programu 500+.

Tak, trzeba odróżnić liczbę urodzeń od dzietności. Liczba urodzeń w Polsce spada i będzie spadać. Szanowni państwo, będzie spadać, nie pierwszy raz o tym mówię w tym miejscu, przez kolejne lata, długie lata, dlatego że bardzo dynamicznie ubywa nam kobiet w wieku prokreacyjnym. Kilka lat temu mieliśmy 10 mln kobiet w wieku prokreacyjnym, dzisiaj już jest mniej niż 9 mln. To jest ogromna różnica. Przy czym te kobiety, które ciągle są zaliczane do wieku prokreacyjnego, jak chociażby ja, już na pewno dzieci nie urodzą.

To się zmieni w ciągu najbliższych kilku lat.

Dzietność w Polsce wzrastała, zaczynała wzrastać po 2016 r. To się załamało, załamał się ten trend, to prawda, załamał się na całym świecie, we wszystkich krajach, które obserwuję, a bardzo bacznie się przyglądam tym procesom, szczególnie w Unii Europejskiej. Są rekordowe spadki dzietności, które są związane oczywiście z pandemią, związane z poczuciem ogólnego zagrożenia i niestabilności. I myślę, że o wiele dłużej będzie trwało wychodzenie z tego stanu takiego poczucia zagrożenia niż wejście w ten stan.

Naszym celem jest to, by w sposób spójny i konsekwentny wprowadzać kolejne elementy związane z polityką prorodzinną, oczywiście nie tylko związane z transferami bezpośrednimi, ale wszystkie inne, o których już była mowa. Dziękuję bardzo, pani minister. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Minister!

Wnioskują oczywiście, mają swoje pomysły, takie jest ich prawo. Natomiast chciałabym przypomnieć moment, w którym wprowadzaliśmy program „Rodzina 500+” Przypominam sobie dyskusję tutaj, na tej sali.

Tam we wnioskach było jasno i wyraźnie powiedziane, że za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL nie było spójnej, kompleksowej polityki prorodzinnej. To właśnie program 500+ był historycznym programem, który zmieniał całą optykę patrzenia na rodzinę. Rodzina za rządów Prawa i Sprawiedliwości stanęła w centrum uwagi. Tak naprawdę przez kolejne lata naszych rządów udoskonalamy, wprowadzamy kolejne elementy.

Mówicie państwo o skrajnym ubóstwie, zwłaszcza o ubóstwie, które dotyczyło rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

W związku z tym, że w czasie. Pani poseł, może pani przestać krzyczeć? Bardzo proszę. Właśnie, to taki zwyczaj tutaj, rzeczywiście. Jest pani na sali plenarnej. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego (druki nr 1541 i 1596) Uprzejmie proszę panią poseł Gabrielę Masłowską o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

W naszym systemie bankowym obowiązują takie zasady i takie przepisy, że kredytem na ogół pokrywa się co najwyżej 80%, w niektórych przypadkach 90% wartości nieruchomości, co oznacza, że pozostałe 20% kosztu danego lokalu mieszkalnego czy domu, czy prawa własności w lokalach wielobudynkowych pokrywa się wkładem własnym, czyli zgromadzonymi środkami własnymi. Okazuje się, że brak środków własnych na pokrycie wkładu własnego jest dla wielu rodzin, zwłaszcza rodzin młodych, na dorobku, podstawową barierą, w ogóle jeśli chodzi o ubieganie się o kredyt, o jakichkolwiek marzenia o własnym mieszkaniu. Podczas prac połączonych komisji były prezentowane badania prowadzone pod kierunkiem prof. Andrzejewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dotyczące preferencji Polaków, jeśli chodzi o formę mieszkania, a także o bariery, które utrudniają zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

W tym względzie projekt, nad którym pracujemy, wychodzi naprzeciw takim preferencjom, takiemu zapotrzebowaniu Polaków, dlatego że ułatwia uzyskanie mieszkania na własność, z prawem własności. Po drugie, z badań wynika, że najważniejszą barierą zgłaszaną przez rodziny zarówno wielodzietne, jak i rodziny młode, barierą, jeśli chodzi o zdobycie mieszkania czy potem powiększenie mieszania w związku z powiększeniem rodziny, jest właśnie brak środków na wkład własny.

Dlatego przedłożona przez rząd propozycja dokładnie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom Polaków i właściwie łączy zalety wszystkich innych dotychczasowych programów, tym bardziej że nie ma tutaj zastosowanego kryterium dochodowego, czyli jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jest to ogromny postęp, ogromny krok do przodu. Jest to nowa propozycja, wydaje się, atrakcyjna dla wielu rodzin. Ale nie jest to realizacja tylko polityki mieszkaniowej. Otóż proszę zwrócić uwagę, że na etapie spłaty kredytu również mamy do czynienia z pewnym wsparciem. Dotyczy to tych rodzin, tych sytuacji, kiedy powiększa się rodzina, przychodzą nowe dzieci na świat. Otóż w takiej sytuacji istnieje możliwość przejęcia spłaty kredytu - nazywa się to spłatą rodzinną - przez bank.

Spłaty te będą dokonywane z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który ma właśnie temu służyć i ma być utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Otóż to są najważniejsze elementy. A więc tym drugim filarem jest jednocześnie zahamowanie poprzez tego typu propozycję rządową negatywnych tendencji demograficznych, a raczej zachęta do powiększania rodziny. To są dwie najważniejsze kwestie, czyli projekt łączy zadania polityki mieszkaniowej i polityki prorodzinnej, łączy te dwie kwestie, rozwiązuje te dwa problemy.

Oczywiście celem jest zapewnienie mieszkania, dachu nad głową, przede wszystkim potrzeb mieszkaniowych. Oczywiście, że także rynek wtórny.

Czy korzyści, które osiągnie rodzina, która skorzystała ze spłaty rodzinnej, czyli spłaty ze środków publicznych części zaciągniętego kredytu, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Będą one wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, należy to również podkreślić, bo to jest także ważna informacja. Będzie to wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym.

Do projektu zgłoszono 12 poprawek, oczywiście 10 poprawek przyjęto i dwie zostały przez komisję odrzucone.

Jeśli w wyniku tego powstanie lokal mieszkalny, z takiej formy dostępu do własnego kąta często korzystają osoby, które mają np. dom jednorodzinny pozwalający na nadbudowę i stworzenie lokalu w miarę niezależnego od rodziny. Tak że są precyzowane przepisy, co w sytuacji, kiedy zarówno kredyt gwarantowany, jak i spłata zostały osiągnięte w wyniku przestępstwa, w wyniku oszustwa. Jakie wtedy będą obowiązywać procedury zwrotu i powiadamiania o tym wyroku sądu.

Szanownymi Państwo!

O dziwo głosowanie nad tym projektem było bardzo pozytywne i jednomyślne. To jest też pocieszająca wiadomość i za to dziękujemy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Anna Milczanowska. Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, druk nr 1541. Po pracach połączonych Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury i po pierwszym czytaniu projektu z druku nr 1596 trudno nie dostrzec pozytywnych zmian zachodzących w obszarze polityki prorodzinnej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Symbolem skutecznego wsparcia polskich rodzin są programy takie jak: „Rodzina 500+” , „Dobry start” czy „Maluch+” oraz dziesiątki innych działań niwelujących negatywne tendencje w zakresie demografii.

Aż ponad 55% badanych uznało, że najpierw powinno się mieć własne mieszkanie, dopiero potem planować dzieci. Rzeczywistość zarysowała potrzebę wprowadzania w życie kompleksowego programu społeczno-gospodarczego, który pozwoli nie tylko odbudować kraj po kryzysie związanym z pandemią COVID-19, lecz także wykonać duży skok cywilizacyjny do przodu.

Jest to znakomita odpowiedź na te oczekiwania.

Tak jak mówiła przed chwilą pani poseł sprawozdawca Gabriela Masłowska, przy pojawieniu się drugiego dziecka w rodzinie Bank Gospodarstwa Krajowego dokona spłaty kredytu w kwocie 20 tys. zł, a jeżeli pojawi się trzecie lub następne dziecko - w kwocie 60 tys. zł. W zakresie proponowanych rozwiązań projekt ustawy łączy cele polityki mieszkaniowej i polityki prorodzinnej. Nie mniej ważne są zapisane w projekcie mechanizmy sprzyjające utrzymaniu wysokiej jakości portfeli kredytowych w sektorze bankowym oraz mechanizm minimalizujący stymulowanie postaw spekulacyjnych, zabezpieczające gospodarstwa domowe przed niekorzystnymi fluktuacjami rynku oraz stabilizujące sytuację finansową polskich rodzin. Mając na uwadze dalszą konsekwentną poprawę stopy życiowej polskich rodzin, w odpowiedzi na wyzwania demograficzne Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Pan poseł Cezary Grabarczyk w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Coraz częściej rozmawiamy o problemach mieszkaniowych w kraju. To dobrze, bo to palący problem. Opozycja chętnie włącza się w prace, gdy projekty mogą realnie zmienić trudną sytuację mieszkaniową, w szczególności młodych ludzi. Dlaczego? Dlatego że to w istocie hołd oddany twórcom programu „Mieszkanie dla młodych” Była o tym mowa także podczas wczorajszych prac na posiedzeniu komisji. Dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość zreflektowało się, dostrzegło błędy, które popełniło jeszcze w poprzedniej kadencji. Cieszę się, że na sali widzę pana ministra Smolińskiego, bo to on był piewcą skasowania tego programu. To pan minister był przeciwnikiem projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Miałem zaszczyt być przedstawicielem wnioskodawców, chcieliśmy wówczas pomóc PiS-owi i zwiększyć pulę środków na program „Mieszkanie dla młodych” Niestety te apele, całej wówczas opozycji, nie spotkały się z aprobatą rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Ale uważamy, że pomoc państwa musi być realna, dlatego proponujemy, aby ten gwarantowany kredyt mógł być także udzielony w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, z wykończeniem nabywanego mieszkania bądź domu jednorodzinnego. Co bowiem młodym ludziom po pustych ścianach, po stanie deweloperskim? Jeżeli już korzystają z pomocy państwa, to niech mogą uwzględnić także wydatki związane z wykończeniem, wówczas ta pomoc będzie realna. Proponujemy także, aby spłata rodzinna obejmowała dwa przypadki losowe. Żyjemy w czasie pandemii i wiemy, jak wiele rodzin poniosło straty bliskich i najbliższych, także wśród ludzi młodych mamy śmiertelne ofiary pandemii. Co wówczas, gdy młodzi ludzie zaciągną kredyt gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i jedno z nich umrze? Sytuacja dramatyczna, trudna do wykluczenia w dzisiejszych czasach. Dlaczego państwo nie chce pomóc w tak trudnej sytuacji? Składamy odpowiednią poprawkę i liczymy na to, że państwo zweryfikujecie swój pogląd. To samo w sytuacji, gdy osoba z powodu długotrwałej choroby, trwającej 18 miesięcy, utraci zdolność zarobkowania i nie będzie mogła obsługiwać kredytu.

Jeszcze raz podkreślam, że będziemy pomagali, chociaż obawiamy się, że tym razem pomoc państwa będzie nie w porę, bo ceny materiałów budowlanych rosną. Wskaźniki, które są zawarte w ustawie, mogą być zbyt wysokie. Na szczęście jest szansa, że Rada Ministrów będzie mogła je obniżyć i stąd moje dwa pytania. Pani marszałek, nie mogę zadać pytań, bo jestem przewodniczącym podkomisji, która zaczyna pracę. Dwa krótkie pytania.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jednym z najważniejszych problemów, z którym obecnie muszą mierzyć się młodzi ludzie, jest dostęp do samodzielnego mieszkania. Na pytanie, czy ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego rozwiąże ten problem, odpowiedź brzmi: nie. Krótkowzroczna polityka rządu jedynie pogłębia problem, zamiast szukać jego rozwiązania.

Rząd brakiem działań w zakresie polityki mieszkaniowej doprowadził do sytuacji, w której boom na rynku napędzają ci, którzy widzą w mieszkaniach jedynie lokatę kapitału, tym samym pozbawiając tysiące osób szans na jego zakup. Zamiast refleksji nad powrotem do budownictwa społecznego nastawionego na zaspokojenie potrzeb polskich rodzin nadal będziemy świadkami rozwoju rynku tzw. korporacji kamieniczników i mieszkaniowych spekulantów. Nie tędy droga. Zrozumieli to nawet nasi zachodni sąsiedzi, którzy podczas przeprowadzonego w ostatni weekend referendum opowiedzieli się za uspołecznieniem tysięcy lokali mieszkalnych. Mieszkańcy Berlina zagłosowali za wywłaszczeniem korporacji i funduszy kapitałowych, które hurtowo skupowały z rynku setki tysięcy mieszkań pod inwestycje i windowały czynsze w całej stolicy Niemiec. Tymczasem polski rząd jedyne co ma do zaoferowania polskim rodzinom, to drenaż ich budżetów domowych na rzecz banków. Państwo powinno powołać państwowego dewelopera odpowiedzialnego za budowanie tanich mieszkań na wynajem czy też przywrócić budownictwo realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Państwo, które podejmuje się budowy mieszkań, nie będzie ich sprzedawać za więcej niż koszt ich wybudowania. Mieszkania będzie można w ten sposób kupić na raty z maksymalnym oprocentowaniem 3%. Chcielibyśmy, żeby tym rozwiązaniom towarzyszyło także utworzenie agencji nadzorującej pozyskiwanie gruntów pod budownictwo społeczne. Tylko w ten sposób w Polsce zaczną powstawać nowe osiedla dla młodych. Nie zwalczymy patologii na rynku mieszkaniowym, ale wprowadzimy nowe. Podczas posiedzenia połączonych Komisji Finansów Publicznych i Infrastruktury nie dowiedzieliśmy się nic o tym, jak w przyszłości przy ewentualnym wzroście stóp procentowych będzie się kształtować zdolność kredytowa przyszłych kredytobiorców. Nie dowiedzieliśmy się, jaki wpływ proponowana ustawa będzie miała na kolejny wzrost cen nieruchomości na rynku, a co do tego akurat możemy być wszyscy pewni przy tej inflacji, która jest. Nie przedstawiono także badań z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na których podobno oparto założenia niniejszej ustawy. Dlaczego nie uzyskaliśmy tych informacji? Bo rządu nie interesują młodzi ludzie i ich rodziny. Gdy pierwsi kredytobiorcy będą popadać w problemy finansowe związane z napisaną na kolanie ustawą o kredycie hipotecznym, PiS będzie już po wyborach, a skutki tych decyzji nie będą ich obchodzić. Ustawa w tym kształcie i z tymi założeniami nie pomoże polskim rodzinom. To kolejne obietnice bez pokrycia, podobne do tych, kiedy rząd obiecywał wybudowanie 100 tys. mieszkań czy wprowadzenie milionów elektrycznych samochodów na nasze ulice. Lewica nie poprze tak przygotowanego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jacek Tomczak w imieniu Koalicji Polskiej. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL - Koalicja Polska w sprawie projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Deklarowanym celem wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez eliminację barier braku własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny przy udzielonym kredycie hipotecznym oraz powstrzymanie negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności, odniesienie się do sytuacji rodzin spłacających kredyt hipoteczny zaciągnięty w związku z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych. Tak więc projekt ustawy łączy cele polityki mieszkaniowej i polityki prorodzinnej. Na poziomie celów wypada nam docenić projekt i dać zielone światło do dalszych prac nad nim. Jak wiemy, jednak diabeł tkwi w szczegółach i warto zadbać o to, aby w tak ważnej ustawie te szczegóły były należycie dopracowane. Warto przypomnieć, że ten projekt pojawia się po 6 latach braku jakichkolwiek sensownych działań ze strony rządu w ramach polityki mieszkaniowej i jest pewnym oddaniem hołdu najlepszemu programowi mieszkaniowemu, jaki był realizowany, a został stworzony przez rząd PO-PSL, czyli programowi „Mieszkanie dla młodych”, gdyż jest bliźniaczo podobny do tego projektu. Natomiast zauważamy w nim szereg mankamentów, dlatego chcemy złożyć szereg poprawek, które troszeczkę zmienią jego kształt. Pierwsza rzecz jest taka, iż nie wiadomo, dlaczego dzisiaj z powodu tego, że przez 6 lat nie było żadnego programu mieszkaniowego, który by uwzględniał elementy polityki prorodzinnej, w tym programie będą uwzględnione tylko te rodziny, które w przyszłości złożą wnioski o udzielenie kredytu gwarantowanego, natomiast nie będą te, które już złożyły. Dlaczego rodzina, która złożyła wczoraj taki wniosek, uzyskała kredyt w banku, nie będzie mogła skorzystać ze spłaty rodzinnej, skoro dziecko urodzi się za rok, za dwa, tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość to narzędzie tworzy dzisiaj? Dlaczego szereg rodzin ma być z tego wykluczonych?

Nie tylko te, które pójdą w trybie tej ustawy dopiero w przyszłym roku, kiedy zostanie ona uchwalona i kiedy te przepisy wejdą w życie.

Każde dziecko w każdej rodzinie, które się rodzi, jest ważne.

Co jeszcze? Chcielibyśmy też, żeby w ten sam sposób były traktowane wszystkie dzieci, więc proponujemy, ażeby.

Nie widzimy powodu, ażeby rodzina, która spodziewa się drugiego dziecka, tę spłatę miała niższą niż rodzina, która spodziewa się trzeciego dziecka. Dzisiaj wszystkie polskie rodziny chcą sobie poprawić sytuację mieszkaniową. Szukają mieszkań większych ze względu na pracę online. Ojciec potrzebuje osobnego gabinetu do tego, żeby mógł spokojnie pracować.

Państwo ciągle nie rozumiecie, że sytuacja na rynku mieszkaniowym to nie jest jakiś dopust boży, tylko rezultat tego, co robiliście wcześniej. I to nie tylko w sprawach ściśle związanych z samymi mieszkaniami. Dlaczego więc mieszkania są drogie? Po pierwsze, Prawo budowlane jest przeregulowane. Wszystkie te regulacje powodują wzrost cen pośrednio lub bezpośrednio.

Im więcej regulacji, tym mniej mieszkań powstaje. Im mniej jest danego produktu w stosunku do zapotrzebowania, tym jest on droższy. Więc recepta: deregulacja, głęboka deregulacja.

Znowu, recepta: mniejszy budżet, mniej regulacji, mniej podatków. Niestabilność prawa, niepewność rynku. Ciągle zmieniająca się sytuacja powoduje, że inwestycje długoterminowe stają się bardziej ryzykowne.

Do tego dochodzą niskie stopy procentowe. Pieniędzy nie opłaca się trzymać nawet na lokatach. W takiej sytuacji szuka się bezpiecznej inwestycji, nawet o niskiej stopie zwrotu. Jeśli więc sztucznie jest zbyt łatwo dostępny dla nich kredyt, a sytuacja jest niepewna, nie ma wielu dobrych miejsc, w których można go zainwestować, ludzie wybierają kapitały chłonne i niskodochodowe, ale za to bezpieczne inwestycje i w ten sposób pompują bańkę na rynku nieruchomości. Recepta: uwolnienie stóp procentowych, deregulacja, stabilizacja prawa, zakończenie koronapaniki. Ale wy nie leczycie przyczyn tylko bohatersko zagłuszacie objawy. W ten sposób tego pacjenta tylko zabijecie. Co robicie w tej ustawie? Namawiacie ludzi do tego, żeby się zapożyczali i kupowali pomimo drożyzny. Kiedy napompowaliście ten balon, to zamiast pozwolić, żeby zmniejszony popyt spowodował, iż ceny będą spadać, mówicie temu młodemu człowiekowi: weź zapłać, ja ci pomogę z kredytem.

Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Ktoś, kto zarabia średnią krajową i chciałby za tę cenę kupić w Polsce mieszkanie, musi nie jeść, nie kupować, nie jeździć i spać kątem u rodziców przez 7 lat, by nabyć lokal w Kielcach lub w Łodzi. Natomiast na lokal w Warszawie odkładać trzeba 13 lat, przypomnijmy, nie wydając na nic innego. Jeśli nasz bohater nie ma kąta u rodziców i musi wziąć kredyt, okresy te wydłużą się około dwóch razy z uwagi na odsetki i koszty. A przecież ludzi umiejących nie jeść przez 26 lat mamy w Polsce nader mało. Wy przychodzicie z ustawą, która niby coś ludziom daje, ale tak naprawdę jeszcze bardziej te ceny mieszkań w Polsce napędza. Eksperci w zakresie mieszkalnictwa, wasi również, ostrzegają, że skutkiem będzie tu nie jakaś zwyżka cen, ale przeniesienie całego rynku na nowy poziom. Nie będę się znęcać nad badaniem mającym uzasadnić ten kompletny zwrot mieszkaniowy w Polskim Ładzie, szanowni państwo.

Kosmiczne ceny mieszkań to jest miara nieudolności tego rządu. To rząd nakręcił spiralę inflacji, zwiększenie kosztów materiałów, pracy, ale też ucieczkę kapitału prywatnego w jedyną inwestycję, na której jeszcze w miarę się nie traci, czyli w nieruchomości. To rząd położył program dostępnych mieszkań na wynajem, wpychając całe pokolenie w konieczność zaciągnięcia kredytów, które spłaca się całe życie. To rząd trzyma w lodówce ustawę o REIT-ach i jest bezbronny wobec zagranicznych funduszy, które wkrótce spowodują kryzys podobny do tego, jaki mamy w tej chwili w Niemczech. To rząd przynosi nam właśnie podpisany akt kapitulacji w postaci tej ustawy, którą można nazwać tylko Bank+, bo to pompa zasysająca z kieszeni młodych Polaków i tłocząca wprost do puli zysków banków i deweloperów. Namawiam opozycję: nie dokładajcie ręki do pompowania cen na rynku mieszkań w Polsce. Bo kiedy przyjdą gorsze czasy, wyższe stopy, będzie problem tak jak w przypadku frankowiczów. My jako Polska 2050 na pewno ręki do tego nie przyłożymy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Ministrze! Wysoka Izbo! Porozumienie co do zasady popiera działania rządu z zakresu mieszkalnictwa, które doprowadzają do polepszenia sytuacji mieszkaniowej, ale chodzi o te działania przygotowane w ówczesnym ministerstwie rozwoju jeszcze pod kierownictwem Jarosława Gowina. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na problemy na rynku mieszkaniowym, które wciąż nie zostały rozwiązane. Przedmiotowy projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym tworzy bowiem jedynie połowiczne rozwiązania. Dziś mamy do czynienia z galopującymi cenami na rynku mieszkaniowym. Popyt przewyższa podaż.

Można temu przeciwdziałać na bardzo wiele sposobów i dziś właśnie tego oczekujemy od rządzących. Gdzie jest złożona i gotowa do procedowania ustawa o bonie mieszkaniowym? Jaki jest los prac nad ustawą o planowaniu przestrzennym czy ustawą o polskich funduszach inwestycyjnych w nieruchomości? Dzisiejsza sytuacja jest zła. Ten projekt w swojej istocie miał być połączony z projektem ustawy o bonie mieszkaniowym, a nie jest. Porozumienie poprze te rozwiązania, ale oczekujemy na kolejne pakiety ustaw gotowe do procedowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas na zadanie pytania na 1 minutę. Zapraszam, pani poseł.

Wysoka Izbo! Kolejny państwa program w ramach Polskiego Ładu to „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do uzyskania własności mieszkania poprzez wzmocnienie zdolności kredytowej.

Zaznaczyć także trzeba, że kredyt na 15 lat to kredyt na bardzo długi czas.

Dziękuję bardzo. Nie ma. Bardzo proszę. Chcę panie i panów posłów zapytać: Gdzie jest 3 mln mieszkań obiecywanych przez PiS? Nie ma. Gdzie jest 100 tys. mieszkań obiecywanych przez PiS? Nie ma.

Nie ma żadnej pomocy. Obiecanki. Dziwi mnie metoda przedstawiania taniego oprocentowania w bankach. Przecież pani poseł Masłowska powinna wiedzieć, że żeby udzielić kredytu, to starsza pani musi przynieść to, co sobie składa na czarną godzinę. A ona odkłada na czarną godzinę. Czy pani to rozumie? Chciałabym powiedzieć, że rząd tu czarował i nie powiedział całej prawdy o tym projekcie. Państwo powinni powiedzieć: masz kredyt, jeśli jesteś młody, ale jeżeli masz zdolność kredytową.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 6 lat działalności rządu Prawa i Sprawiedliwości to 6 lat błędów, wypaczeń i zwykłej nieudolności w dziedzinie polityki mieszkaniowej. Ta ustawa, którą próbujecie to w jakiś sposób naprawiać, spowoduje. Jednym z jej skutków będzie niestety dalszy wzrost, dynamiczny wzrost cen mieszkań. To przypomina trochę taki mechanizm, w którym 6 lat psujecie, próbujecie naprawiać, a niestety sposób, w który to naprawiacie, znowu spowoduje kolejne zepsute elementy i tym zepsutym elementem będzie właśnie wzrost cen mieszkań. Należałoby po pierwsze zapytać, co będzie następne. W jaki sposób następny raz będziecie naprawiać to, co dzisiaj psujecie? Po drugie, w jaki sposób zabezpieczycie ludzi, którzy wezmą dzisiaj kredyty nisko oprocentowane (Dzwonek), a stopy procentowe pójdą w górę i kredyty podrożeją? Zapraszam. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. w Polsce urodziło się nieco ponad 356 tys. dzieci, z czego 93 tys., czyli co czwarte dziecko, w związkach nieformalnych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w projekcie ustawy znalazła się definicja gospodarstwa domowego rozumianego jako gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną. Czy zapis ten dotyczy jedynie tradycyjnego modelu rodziny, czy też osób pozostających w związkach nieformalnych? Czy na pomoc z tytułu: mieszkanie bez wkładu własnego mogą liczyć rodziny, w których jeden z partnerów ma dziecko, a drugi po prostu go nie przysposobił? Pan poseł Władysław Kurowski, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym to kolejny element spójnej polityki prorodzinnej skierowany do rodzin przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Daje dwie możliwości. Jedna to brak konieczności posiadania swojego wkładu, a druga to możliwość umorzenia części kredytu w związku z rodzeniem się kolejnych dzieci. Pytanie mam takie: Czy ustawa określa maksymalny czas realizacji inwestycji, czyli budowy np. domu?

Trzecie pytanie: Jaka jest maksymalna kwota (Dzwonek) umorzenia kredytu przy rodzeniu się kolejnych dzieci? Zapraszam. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Podstawą do udzielania kredytu jest zawsze zdolność kredytowa i wkład własny. My pomagamy z wkładem własnym, my pomagamy też z kolejnym dzieckiem w spłacie tego kredytu kolejnymi kwotami, którymi będziemy tak jakby wspomagać młode małżeństwa i rodziny. Rozumiem, że każde młode małżeństwo, każda osoba, która bierze kredyt, jest racjonalna i umie policzyć, że my pomagamy tylko z wkładem własnym, pomagamy w spłacie tego kredytu, ale także rozumiem, że ta zdolność jest nadal wymagalna. Czy faktycznie tak jest, że zdolność kredytowa jest nadal podstawą do udzielenia tych kredytów? A my po prostu pomagamy z wkładem własnym i w drugim elemencie pomagamy w spłacie wraz ze wzrostem liczby dzieci w danej rodzinie. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Czy przedmiotowa regulacja prawna przewiduje dotację państwa na tzw. wkład własny do kredytu bankowego i na jakich warunkach? Czy kredytobiorca będzie musiał wpłacić finalnie tę kwotę do banku i w jakim terminie będzie musiał wnieść wkład własny? Czy program oferowany jest tylko tym, którzy mają zdolność kredytową, tylko nie mają żadnych innych swoich oszczędności? Jak w takim razie będą w stanie spłacić kredyt? Czy państwo chce im w tym pomóc? Pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Muszę przyznać, że takie powiązanie polityki mieszkaniowej z polityką prorodzinną w ustawie teoretycznie nie jest pomysłem złym, ale szkoda, że za słowami nie idą czyny. Rodzice będą czuli się bezpiecznie, gdy uwolni się ich od wieloletnich kredytów hipotecznych. Bezpieczeństwo umożliwi im dopiero dostęp do żłobka, przedszkola, ośrodka zdrowia i mieszkań większych niż kawalerka. Tymczasem kosmiczne ceny mieszkań to skala porażki tego rządu. Państwo powinno stworzyć dostępny system mieszkań na wynajem, które wybudowane zostaną w przemyślanych lokalizacjach i w przyjaznym otoczeniu. W Narodowym Programie Mieszkaniowym - sami o tym wspominacie - skończyło się na dosypywaniu pieniędzy bankom i wspieraniu patodeweloperki. Przestańcie leczyć dżumę cholerą. Przestańcie udawać, że robicie cokolwiek, żeby rozwiązać kryzys demograficzny. Dziękuję. Wysoka Izbo!

Ale raczej wątpię, żeby ono pomogło komukolwiek, bo wygląda na to, że jeśli je uchwalimy, to w średnio krótkim czasie te mieszkania bardzo zdrożeją. Czy państwo w ogóle monitorujecie rynek sprzedaży mieszkań? W samej Warszawie. To był pierwszy fundusz, a za chwilę przyjdą następne.

Chciałem wiedzieć, czy monitorujecie rynek mieszkań. Zapraszam, pani poseł. Wysoka Izbo! Procedowana ustawa może skutkować pewną poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce, jednak poszczególne jej zapisy wymagają gruntownego przeformułowania. Największe obawy budzi ograniczenie możliwości uzyskania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego poprzez odwołanie się do kryterium ceny. Mając na uwadze już i tak gwałtowny wzrost cen mieszkań, chcę powiedzieć, że zaproponowane ograniczenie w praktyce uniemożliwi skorzystanie z programu tam, gdzie jest on potrzebny, czyli w szczególności w miastach, co już samo w sobie rodzi absurd. Jaką rząd ma pewność, że wprowadzenie proponowanych przepisów przy obecnych warunkach rynkowych nie zwiększy bańki cenowej na rynku mieszkaniowym? Spowodowałoby to, że mieszkania byłyby jeszcze droższe i dostępne dla coraz mniejszej (Dzwonek) grupy osób, a przecież nie o taki efekt chodzi. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W tej ustawie panujemy.

Chciałabym zapytać, panie ministrze. Pani poseł, pani przewodnicząca.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Robert Obaz, klub Lewicy. Pani Marszałek! Pani przedmówczyni pochwaliła, jak ten program dobrze wygląda i jak państwo panują nad cenami mieszkań.

Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Obecna polityka rządu, mieszkaniowa polityka rządu to namawianie młodych ludzi do zaciągania zobowiązań bankowych, zaciągania kredytów za pośrednictwem BGK na swoje wymarzone mieszkanie, w momencie kiedy mamy w Polsce najniższe stopy procentowe i najwyższe ceny mieszkań. Kieruję pytania do pana ministra: Czy jesteście w stanie zagwarantować stałe stopy oprocentowania przez cały okres kredytowania, czyli przez 15 lat? I po drugie, dlaczego BGK w czasie udzielania takich kredytów nie zrezygnuje z opłat i prowizji bankowych, tak aby nie wprowadzić młodych ludzi w spiralę zadłużenia, jak to było w przypadku frankowiczów? Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cieszę się, że PiS powraca do naszych dobrych rozwiązań. Dzięki programowi MdM powstało ponad 100 tys. mieszkań. Dziwię się, że czasami państwo zachowujecie się jak komuniści po II wojnie światowej i wszystko, co nie wasze, po prostu likwidujecie bez względu na to, czy to działa dobrze, czy działa źle. Państwo w to miejsce obiecywaliście 100 tys. mieszkań i wiemy, jakim to się zakończyło sukcesem. Powstało bardzo, bardzo niewiele mieszkań. Po drugie, nasz program dawał konkretne pieniądze, pieniądze wpływały na konto tego, który kupował mieszkanie. Państwo nie dajecie pieniędzy, tylko dajecie gwarancję. Stąd wnioskuję o to, by pójść dalej: trzeba wprowadzać zwolnienie podatkowe dla tych, którzy decydują się na zakup własnego mieszkania. I ostanie pytanie do pana, panie ministrze. Pani poseł Magdalena Filiks, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Do pani poseł Milczanowskiej się zwrócę, bo o to jest właśnie moje pytanie. Pani poseł, z całym szacunkiem, ale pani nie zrozumiała, co wy macie w projekcie. Wy nie macie limitu ceny, żeby zagwarantować ceny, tak jak pani przed chwilą powiedziała, tylko macie limit, w którym poruszać się mają rodziny - tylko w takim limicie będą mogły kupić mieszkanie. Ja pani powiem, do czego to doprowadzi. Im jest mniejsze - to widać po kawalerkach - tym jest droższe.

Wasz program już dzisiaj, jak mówią eksperci, te ceny podniesie. Ludzie wezmą te kredyty przy bardzo niskich stopach procentowych, które wcześniej czy później wrócą do swoich poziomów, zakredytowani będą olbrzymimi kwotami wartości kredytu, żeby spełnić wasz wskaźnik. A więc ja pytam, czy ktoś się zastanowił nad tym (Dzwonek), żeby chociaż, jak już takie rzeczy ludziom robicie, ściągnąć te wskaźniki. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę. Ojej, ale pani musi zawsze krzyczeć, tak? Tak na co dzień już pani ma? Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Gratuluję pani i pani rodzinie współczuję. Wysoka Izbo! 6 lat czekamy na realny projekt mieszkaniowy, bo w tym obszarze dzisiaj rządząca koalicja nie może mieć żadnego orderu, który sobie do klapy przytwierdzi. Dlaczego nie wróciliście wprost do założeń tego programu, który był sprawdzony, który dobrze funkcjonował na rynku i z jednej, i z drugiej strony?

Wiecie ile? O połowę mniej.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Do tego projektu dobrze pasuje sformułowanie: lepiej późno niż później. Później - bo ceny mieszkań są maksymalne, a podwyżka stóp procentowych jest niestety za rogiem, przekroczyliśmy próg inflacji 5%. Teraz wyraźnie widać, jak bardzo się spóźniliście, by wesprzeć waszą politykę prorodzinną filarem mieszkaniowym. Teraz chcecie to na gwałt uzupełnić. Ale trzeba zauważyć, że problem pułapki kredytowej jest absolutnie realny, absolutnie realny. I teraz pytanie jest takie: Ile dochodu rozporządzalnego musi mieć rodzina pięcioosobowa - bo wasze preferencje wystarczą tak naprawdę na mały pokoik dziecięcy, i to wspólny - żeby utrzymać ten nowy dom? Czy będą musieli wszystko zwracać? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wiceminister rozwoju i technologii powiedział publicznie: projekt ma łączyć cele polityki mieszkaniowej i prorodzinnej, przewidujemy mechanizm limitowania cen transakcyjnych, by ustawa nie spowodowała wzrostu cen na rynku. Niebezpiecznie przypomina to sytuację i podobną ustawę w Stanach Zjednoczonych, która ostatecznie doprowadziła do potężnego krachu w 2008 r. Proszę zatem o informację: Co to jest ten mechanizm limitowania cen transakcyjnych? Bardzo jestem ciekawa, panie ministrze, jak będziecie to regulować. I proszę o szczegółową informację na piśmie. Pan poseł Jacek Tomczak, Koalicja Polska. Zapraszam.

Oczywiście, że ceny mieszkań będą rosły.

I tutaj jest konieczna bardzo jasna, stanowcza polityka, ażeby wesprzeć chociażby dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, poprawić jakość i tempo wykonywania planów, udzielenia pozwoleń na budowę - wiele, wiele narzędzi.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jesteśmy świadkami zmiany paradygmatu rządów.

Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia program dla rodzin, dla Polaków, którzy tych pieniędzy zbyt dużo nie posiadają. Do tego również dochodzi problem odwrócenia negatywnych tendencji demograficznych. Chciałem zapytać: Ile polskich rodzin może skorzystać z tego programu według waszych wyliczeń? Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zadanie pytania pana posła Jana Szopińskiego. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wiemy już, że proponowane gwarancje mogą stanowić pułapkę dla kredytobiorców, gdyż ułatwiają zaciągnięcie kredytu, aby następnie możliwie szybko uwolnić bank od ewentualnego ryzyka oraz pozostawić beneficjentów tych gwarancji samym sobie. Mam pytanie do pana ministra.

Czy rząd proponuje w tej sprawie jakieś rozwiązanie? Uprzejmie proszę pana ministra o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Pytanie zada teraz pan poseł Dobromir Sośnierz.

Nigdy nie przychodzi im do głowy, żeby przyznać się do błędu i poustawiać wszystko tak jak było. Jeśli nie podoba wam się, nie wiem, kolor oczu waszej dziewczyny, to nie możecie wziąć łyżki i wydłubać jej oczu, bo widzieliście, że koleżanka ma lepsze. Tak samo nie da się w tak niemiłosiernie przeregulowanej gospodarce z niskimi stopami, inflacją i loterią różnych przepisów i obostrzeń przeszczepić (Dzwonek) niskich cen mieszkań czy dostępności mieszkań ot tak. Pan poseł Siekierski chciałby zabrać głos? To prosimy pana posła Smolińskiego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przez to zabrakło jakiegokolwiek wsparcia dla budownictwa społecznego. Zlikwidowaliście nasz dobry program „Rodzina na swoim” Pytanie zada pan poseł Krzysztof Paszyk. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Odpowiadam panu posłowi Smolińskiemu. Panie pośle, jaki wpływ na ilość powstających mieszkań ma polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości?

Dobrze prowadzona polityka prorodzinna przede wszystkim (Dzwonek) powinna cechować się sprawiedliwością. Dlatego zachęcamy do merytorycznej rozmowy z Koalicją Polską, z panem posłem Jackiem Tomczakiem, który złożył poprawkę.

O to prosimy i zachęcamy do dialogu w sprawie tej ustawy. Proszę teraz pana posła Romualda Ajchlera. Wysoka Izbo! Nie wychodzę na mównicę po to, żeby przypominać o 3 mln mieszkań, które były obiecane.

Mieszkańcom naszego państwa nie chodzi o obietnice, o kolejne programy, bo mamy już kolejny, ale o konkretną pomoc. Czy nie warto by było, czy rząd rozważał taką sytuację, na wzór tego, co ma być w rolnictwie, zająć się budową przez deweloperów czy przez holdingi, które stworzy, czy spółki, których jest tyle w Polsce, by wybudować mieszkania i postawić te mieszkania do dyspozycji?

Dziękuję bardzo.

Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Instrumenty wsparcia budownictwa, które proponuje rząd, niestety nie są dla wszystkich. Są elementem strategii demograficznej, a nie rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby, zwłaszcza potrzeby młodych ludzi. Rząd, realizując politykę podatkową w ustawie, o której będziemy rozmawiać za chwilę, pogarsza sytuację osób posiadających mieszkania na wynajem, czyli tych, którzy zainwestowali z własnych pieniędzy i robią to na rynku. Dzięki tym rozwiązaniom, tzw. rozwiązaniom podatkowym, pogorszy się sytuacja m.in. studentów i młodych ludzi, którzy wynajmują te mieszkania. Moje pytanie dotyczy Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Odbudowy. Tam zapisano m.in. możliwość wsparcia inwestycji: zielone budownictwo wielorodzinne. Na wniosek Lewicy wpisano możliwość budowy mieszkań na wynajem (Dzwonek), 75 tys. mieszkań na wynajem. Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Czesław Siekierski.

Panie Marszałku! Wszyscy wiemy, że dla stabilizacji funkcjonowania rodziny, szczególnie młodej rodziny, podstawowy wpływ mają dwa obszary: praca i mieszkanie. One ograniczają wszelkiego rodzaju wyjazdy zagraniczne, poszukiwanie swojego miejsca poza krajem, mają także wpływ na poprawę sytuacji demograficznej. Na ile przeprowadziliście analizę, także analizę innych rozwiązań? Jaki wywoła efekt, jeśli chodzi o zainteresowanie?

Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Paweł Krutul. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o mieszkania w woj. podlaskim, w Białymstoku, w stolicy województwa, ceny dochodzą do 10 tys. za metr. Kiedy państwo rządzący, Prawo i Sprawiedliwość, przystąpią z całą klasą polityczną do planowania projektu na wiele, wiele lat, na 10, 15, 20 lat?

Tak że proszę o zaproponowanie takich spotkań, żeby wszystkie kluby opozycyjne mogły się również wyrazić, żeby taki plan był stworzony na więcej niż rok, 2 lata, 5, 10 czy 20 lat. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pana Piotra Uścińskiego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za tą debatę, za pytania, które padły podczas tej debaty. Faktycznie dzisiaj pracujemy nad projektem ustawy nieco poprawionym przez komisję, projektem o skróconej nazwie: o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Bardzo często ten problem wychodzi również w badaniach. To problem braku pieniędzy na wkład własny przy kredycie na zakup pierwszego mieszkania, na wybudowanie domu czy na powiększenie mieszkania, jeśli jest to rodzina, która na małym metrażu, w kawalerce, wychowuje już np. dwoje, troje dzieci.

Być może singlowi, nie tylko rodzinie.

Tak jak zostało powiedziane, ten projekt łączy w sobie politykę mieszkaniową z polityką prorodzinną.

Przy okazji powiem, że osoba, która bierze ten kredyt, nie płaci żadnych wielkich prowizji do BGK ani większych odsetek od kredytu.

Jaka jest maksymalna kwota? Nie ma maksymalnej kwoty.

Bo dlaczego jeśli w rodzinie jest już kilkoro dzieci, nie spłacać za kolejne?

Państwo, gdy rządziliście, stworzyliście program, który faktycznie pomagał ludziom nabywać mieszkania, tylko tam pieniądze przekazywane na zakup mieszkania trafiały bezpośrednio do deweloperów. My robimy program, który ma spowodować też wzrost dzietności. Nie tylko pomagamy ludziom kupić mieszkania, ale mamy spowodować wzrost dzietności.

My w tym programie też nie zakładamy, że powstanie więcej mieszkań, ale spójrzcie na całokształt polityki państwa za czasów Prawa i Sprawiedliwości i za waszych czasów. Za waszych czasów budowano w Polsce rocznie.

Za naszych czasów dzięki polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości podaż na rynku mieszkaniowym jest o 50% większa. Budujemy 76% więcej budynków wielorodzinnych niż wy. Dzięki naszej polityce budują to Polacy.

Ona pomoże ludziom decydować się na budowę własnego domu, bo przecież wielu Polaków te własne domy chce budować. Ale nie chcę przechodzić do innej ustawy przy tej wypowiedzi. Szanowni Państwo!

Taka rodzina chciałaby powiększyć swoje mieszkanie, kupić większe. Dla tej rodziny też jest to możliwe. Jeśli jest trójka dzieci, to ten limit to 75 m2, przy czwórce dzieci – 90 m2.

Pytaliście państwo o mechanizm zabezpieczający przed wzrostem cen mieszkań, czyli taki mechanizm limitowania cen mieszkań.

Ale nie chcemy finansować, nie chcemy, żeby przy tym kupowano mieszkania, które będą sprzedawane dużo powyżej wartości.

Wprowadzamy tutaj też taki mechanizm, że w zależności od sytuacji rynkowej i społecznej Rada Ministrów będzie mogła obniżyć ten wskaźnik.

Każdy kredytobiorca powinien dostać taką ofertę, kiedy bierze kredyt, żeby mógł wybrać. A więc kredytobiorca ma prawo wybrać kredyt ze stałą stopą procentową, jeśli tego chce. UOKiK i KNF rekomendują zresztą i promują stałą stopę procentową.

Było też pytanie opozycji dotyczące zakupów pakietowych mieszkań. Faktycznie takie transakcje na rynku się zdarzają. Widzimy i obserwujemy to, co dzieje się w Berlinie.

Intensywnie pracujemy nad tym, żeby zapobiec tego typu problemom, jakie teraz są w Berlinie.

Szanowni Państwo! Te odpowiedzi zostaną udzielone. Jeszcze tak na szybko sprawdzam, czy czegoś nie ominąłem z tego, co wynotowałem. Chyba nie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za tę debatę, za pytania i bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie tego projektu ustawy w trzecim czytaniu. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Teraz głos zabierze sprawozdawca komisji pani poseł Gabriela Masłowska. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku.

Jest to konsekwentne działanie. Może należałoby tylko zwrócić uwagę na kwestię przeciwdziałania spekulacjom w obrocie tego typu mieszkaniami, bo one będą nabywane na korzystnych warunkach.

Nie wiem, czy tego typu zabezpieczenia są wystarczające, ale miejmy nadzieję, że tak. Jednocześnie padały tutaj często opinie, jak zwykle bywa niemal przy każdej ustawie, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy nie wywiązuje się z obietnic, że nie buduje, że jest katastrofalna sytuacja mieszkaniowa itd., itd. Proszę państwa, katastrofalna sytuacja mieszkaniowa rzeczywiście była, dopóki rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wkroczył ze swoimi programami, wspierającymi także samorządy.

Tak budowali mieszkania. Dopiero teraz, kiedy rząd wkroczył ze wsparciem budownictwa czynszowego, w którym dopłaca 80% środków na budowę, trochę to ruszyło, ale ostatnio także program SIM, społeczna inicjatywa mieszkaniowa, którą wreszcie zauważają samorządy. Próbują się na tej zasadzie zaangażować w budownictwo mieszkaniowe, bo dostają 80% środków od państwa. Oczywiście wtedy są plany budowy kilkuset mieszkań, nagłośnione w prasie lokalnej jako ich sukces. Jest to możliwe tylko dzięki temu, że rząd ze środków publicznych Banku Gospodarstwa Krajowego tak mocno wspiera samorządy w budownictwie czynszowym, komunalnym czy tym społecznym. Inaczej byłaby tragedia.

Była też wypowiedź guru Platformy Obywatelskiej, guru ekonomii, pani poseł Skowrońskiej, która z wielką lubością poucza innych posłów, dyscyplinuje, co powinni wiedzieć, a nie wiedzą. To jest jej stała metoda pracy parlamentarnej, komisyjnej itd.

A po drugie, nie tędy droga, jak powiedziałam.

Bardzo dziękuję, pani poseł. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druki nr 1502 i 1594) Proszę pana posła Jana Dudę o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie połączonych komisji o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zawartym w druku nr 1502. Kilka słów o projektowanej ustawie.

Struktura rynku rolno-spożywczego sprawia, że w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych często występują znaczne różnice w sile przetargowej pomiędzy dostawcami a nabywcami produktów rolnych i spożywczych. W praktyce stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych ma miejsce w całym łańcuchu dostaw żywności. Na poszczególnych etapach łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych funkcjonuje różna liczba podmiotów o różnym rozmiarze działania. W Polsce oraz niektórych innych krajach Unii Europejskiej występują silne, ekonomicznie skonsolidowane podmioty sektora produkującego surowce rolne i artykuły spożywcze. Różnice w potencjale ekonomicznym między dostawcą a nabywcą mogą prowadzić do narzucenia nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty większe podmiotom mniejszym. Nieuczciwe praktyki stosowane przez podmioty z przewagą kontraktową wywierają presję na marże i zyski podmiotów gospodarczych, co może prowadzić do niewłaściwej alokacji zasobów, a nawet spowodować wyparcie z rynku podmiotów, które w przeciwnym razie byłyby rentowne i konkurencyjne. Dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i żywnościowych jest niezbędne zachowanie dobrych relacji między wszystkimi jego ogniwami.

Co prawda w naszym kraju od 12 lipca 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, jednakże w obowiązującej ustawie nie wprowadzono np. zamkniętej listy nieuczciwych zachowań, określając je bardzo ogólnie.

Dziękuję bardzo panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję.

Ale przedtem jeszcze, szanowni państwo, mam przyjemność przekazać, że naszym dzisiejszym obradom przysłuchuje się obecnie delegacja Parlamentarnej Grupy Przyjaźni z Rzecząpospolitą Polską Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii z przewodniczącą panią Alenką Jeraj na czele. Serdecznie witamy naszych szanownych gości. Wracamy do porządku obrad i proszę teraz panią poseł Teresę Hałas o przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pierwsze czytanie omawianego projektu odbyło się 17 września na 37. posiedzeniu Sejmu i projekt skierowany został do rozpatrzenia w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 28 września te komisje się zebrały i na swoim posiedzeniu ten projekt został bardzo wnikliwie przeprocedowany. Przedstawiony projekt ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. W strukturze rynku rolno-żywnościowego zauważa się zjawiska nieuczciwych praktyk handlowych pomiędzy dostawcami a nabywcami produktów rolnych i spożywczych w całym łańcuchu dostaw żywności. Takie praktyki obserwowane są niemalże we wszystkich krajach Unii Europejskiej z uwagi na fakt występowania silnych i ekonomicznie skonsolidowanych podmiotów sektora dystrybucji, a często nawet przetwórstwa, względem słabszych i rozdrobnionych podmiotów produkujących surowce rolne i artykuły spożywcze. Z tego powodu na rynku dochodzi do nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez te podmioty, co często powoduje wyparcie słabszych podmiotów z rynku. Dla prawidłowości funkcjonowania łańcucha dostaw żywności jest niezbędne zachowanie dobrych relacji pomiędzy wszystkimi ogniwami.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest przyjęcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi, a implementacja znacznie zmienia zakres obowiązującej dotychczas ustawy z 15 grudnia 2016 r. W stosunku do obowiązujących przepisów projekt ustawy wprowadza nowe zmiany polegające m.in. na rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych, zmianie definicji nabywcy, zdefiniowaniu nieuczciwych praktyk, określeniu dysproporcji w potencjale ekonomicznym czy wprowadzeniu procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. Projektowana ustawa w swoim założeniu gwarantuje bardziej przejrzyste warunki funkcjonowania podmiotów w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Dostawcy, w tym rolnicy, oraz mali i średni przedsiębiorcy wytwarzający produkty rolne i spożywcze będą mieli większą pewność funkcjonowania na rynku wspólnotowym, w tym rynku krajowym, co powinno przełożyć się na działania prorozwojowe, w tym inwestycyjne i innowacyjne tej grupy społeczno-zawodowej. Projekt zakłada szereg zapisów kompetencyjnych dla prezesa UOKiK-u, w tym nakładanie kar odpowiednio skatalogowanych w poszczególnych artykułach, czy możliwości zastosowania przepisów dobrowolnego poddania się karze stronom sporu, czyli dostawcy lub nabywcy. Projekt pozwala zgodnie z art. 47 na określenie okoliczności łagodzących przy ustaleniu wysokości kar. Wejście w życie projektowanej ustawy nie wyłącza wystąpienia przez przedsiębiorcę z roszczeniem do sądu powszechnego na drodze cywilnoprawnej. Projekt nie zakłada zwiększenia wydatków z budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego. Ponieważ zakładany projekt ustawy wypełnia zapisy dyrektywy, klub parlamentarny popiera tę ustawę, jednakże, panie marszałku, składa jedną poprawkę. Za praktyki nieuczciwe wykorzystujące przewagę kontraktową uznaje się w szczególności praktyki polegające - i w uzasadnieniu są wymienione te wszystkie praktyki. Nie będę już miała czasu na ich wymienienie. Bardzo dziękuję, pani poseł. Teraz głos zabierze pan poseł Piotr Borys, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Szanowny i Drogi Marszałku! Wysoka Izbo! Zgromadzenie Przedstawicieli Parlamentu Słowenii!

Faktycznie jest potrzeba stworzenia nowej ustawy. Ta przestrzeń regulacji znalazła swoje odzwierciedlenie w prawie europejskim, które dzisiaj wdrażamy do prawa polskiego.

Zostali na nowo określeni także nabywcy, mówimy o przedsiębiorcach, ale także o organach publicznych, które podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych.

Ja tę poprawkę przedstawię panu marszałkowi.

My tę ustawę poprzemy, co podkreślam raz jeszcze. Składamy poprawkę praktyczną w interesie polskich rolników. Mamy nadzieję, że będziemy sukcesywnie eliminować te fatalne, często zbójeckie praktyki, które wymierzone są w polskich producentów, w polskich przetwórców, że praktyka pozwoli niwelować te fatalne doświadczenia, że skrócimy łańcuchy dostaw, że kwestie marży będą uczciwie dzielone pomiędzy tymi, którzy wytwarzają lub przetwarzają produkty, a właśnie odbiorcami.

Proszę panią poseł Katarzynę Kretkowską o przedstawienie stanowiska klubu Lewica. Klub Parlamentarny Lewica opiniuje pozytywnie projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ten projekt stanowi wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy nr 633 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw rolnych i spożywczych.

Dyrektywa jedynie poszerzała bądź umożliwiała poszerzenie zakresu jej obowiązywania, zatem wdrożenie tak naprawdę polega na nowelizacji już obowiązującej ustawy. Ustawa winna chronić interes przede wszystkim rolników indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego i przez to środowisko jest oczekiwana. Jest zatem dla nas rzeczą zupełnie niezrozumiałą i nie zostało to wyjaśnione w czasie prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad tą ustawą, dlaczego ministerstwo rolnictwa zabrało się za te prace dopiero 2 lata po wejściu w życie dyrektywy, i to dopiero po kilkukrotnych ponagleniach ze strony Komisji Europejskiej. Przez ponad 2 lata ministerstwo rolnictwa ignorowało żywotne interesy 940 tys. polskich rolników, producentów żywności i 160 tys. przetwórców lokalnych, którzy czekają na te zapisy, zapisy eliminujące nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nad nimi przez przede wszystkim wielkie sieci handlowe, nabywców ich produktów.

Czy został dotrzymany? Postępowanie naruszeniowe w tej sprawie prowadzone jest w oparciu o art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Gdy dojdzie do wniesienia skargi do TSUE, Komisja będzie w niej wnioskować o nałożenie na Polskę ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej, o czym od wiosny alarmuje zarówno premiera, jak i ministra rolnictwa minister ds. Unii Europejskiej. Ponawiam pytanie: Czy 2 lata zwłoki z implementacją dyrektywy to tylko bałagan i dyletantyzm w ministerstwie rolnictwa czy celowe działanie w interesie wielkich sieci handlowych? W toku konsultacji projektu złożono do niego 253 uwagi, z których 150 nie uwzględniono lub uwzględniono w bardzo ograniczonym zakresie. Wśród tych nieuwzględnionych dominują uwagi polskich rolników, producentów żywności bądź lokalnych przetwórców wskazujące na nieprecyzyjność proponowanych zapisów, ich możliwą wieloznaczność i kłopoty interpretacyjne, co, jak wiemy, jest powszechną zmorą polskiego prawodawstwa. W czasie prac komisji rolnictwa na pytanie o te odrzucone uwagi otrzymywaliśmy wyjaśnienia, że owe wątpliwości będą rozstrzygane w toku stosowania tej ustawy przez UOKiK na korzyść rolników bądź że już obowiązująca ustawa i praktyka jej stosowania nie potwierdziły przypadków uzasadniających te wątpliwości. Ciężar odpowiedzialności za dobre stosowanie projektowanych zapisów i ich mądrą interpretację ministerstwo proponuje zatem przerzucić na barki prezesa UOKiK-u. Należy jedynie przestrzec urząd przed nadgorliwością i apelować o zdrowy rozsądek. W otrzymanym przez posłów i posłanki piśmie od np. kilku mleczarskich branżowych organizacji zrzeszonych w Porozumieniu dla mleczarstwa czytamy o postępowaniu wyjaśniającym prezesa sprzed 5 lat w związku z wejściem w życie ustawy o tym samym tytule, w którym prezes wezwał wiele podmiotów przetwórczych, które nierzadko prowadziły transakcje z wieloma dostawcami, np. największe polskie spółdzielnie mleczarskie zrzeszające po kilka tysięcy członków, największe spółki prawa handlowego zajmujące się przetwórstwem mleka, do przygotowania i dostarczenia zestawień dostaw mleka za 3 lata wstecz, odrębnie dla każdego dostawcy, z kopiami umów zawartych z każdym dostawcą pod groźbą nałożenia kary pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość 50 mln euro, jeżeli przedsiębiorca choćby nieumyślnie nie udzielił żądanych informacji lub udzielił informacji wprowadzających w błąd. Te spółdzielnie mleczarskie tutaj wnoszą, żeby nie brać przykładu z tej praktyki. Już jej nie będę opisywać szczegółowo. Tak że chciałabym te zastrzeżenia i apel o zdrowy rozsądek przekazać panu prezesowi UOKiK, na którym spoczywa ciężar dobrego stosowania tej ustawy.

Panie Marszałku!

W związku z tym dobrym zwyczajem byłoby, abyśmy pismo, które rząd musiał przedstawić Komisji Europejskiej do 27 września, otrzymali. Dziękuję bardzo panu posłowi. Głos zabierze pan poseł Mirosław Maliszewski, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Dyskutujemy dzisiaj o wprowadzeniu przepisów, które mają ukrócić zjawisko wykorzystywania przewagi rynkowej nazywanej przewagą kontraktową, nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej do tego, aby narzucać dostawcom produktów rolno-spożywczych do sieci sklepów niekorzystne warunki tej współpracy. Otóż w drodze rozwoju gospodarczego każda firma dąży do tego, żeby mieć jak najlepszą pozycję na rynku i w przypadku sieci supermarketów tę pozycję na rynku zdobywają one poprzez budowanie nowych obiektów, poprzez zwiększanie powierzchni handlowej. Już dzisiaj mamy w Polsce takie sieci, które mają nie kilkadziesiąt, nie kilkaset, ale nawet kilka tysięcy sklepów. W związku z tym one dysponują miejscem, na którym następuje styk sprzedający - kupujący, czyli półką sklepową i miejscem, do którego dociera konsument finalny i podejmuje decyzję, jakie produkty kupić. Nawiasem mówiąc, położenie półki ma również ogromny wpływ, a więc to, czy jest to półka w zasięgu tego konsumenta, czy jest nisko położona, do której on się musi schylić. Można by powiedzieć, że przewaga kontraktowa nie jest zjawiskiem obcym, ale najgorsze jest to, że te sieci, te sklepy próbują nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec tych, którzy dostarczają do tego sklepu, którzy biją się między sobą o to, aby mieć dostęp do półki sklepowej, która z kolei pozwoli im dotrzeć do konsumenta.

Dyrektywa europejska Parlamentu Europejskiego i Rady przedstawia szereg czynności, które państwa członkowskie powinny w swoim prawie zastosować, aby ten proceder nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej na rynku, a więc tej dominującej pozycji na rynku, ukrócić.

Komisja Europejska zaproponowała szereg czynności, które mają wdrożyć państwa członkowskie, aby temu zjawisku zapobiec. Po pierwsze są to czynności niedopuszczające do tego, aby słabszy podmiot był ogrywany przez silniejszy podmiot. I po drugie Komisja Europejska proponuje, żeby państwa członkowskie mogły zastosować system kar, jeżeli dochodzi do tego procederu, czyli wykorzystywania nieuczciwego przewagi kontraktowej.

Nie ma wzmocnienia jego pozycji. Nie ma zapisanych elementów, które nie mogą się w tej umowie znaleźć, a wprost jest zapis, który mówi, że można w drodze dobrowolnych umów zrezygnować z zapisów, które są dla dostawcy niebezpieczne. To niestety otwiera precedens, który będzie prowadził do tego, że sieci w drodze negocjacji, w momencie kiedy będą decydować o tym, od kogo będą kupować i za ile, będą wymuszały zgodzenie się przez dostawców na określone warunki. Niestety ustawa w obecnym kształcie to umożliwia. Ustawa jest dobra i o tym było już dzisiaj mówione. Jest dobra w zakresie możliwości dawanych prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale to już jest następny etap. To jest etap mający zastosowanie wtedy, kiedy już nastąpiło przestępstwo, a nie ma w tej ustawie zabezpieczenia przed popełnieniem przestępstwa. Dlatego my jako klub składamy kilka poprawek, które będą bardziej się odnosiły do intencji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady, uwzględniających wzmocnienie pozycji dostawcy względem sieci supermarketów, a nie tylko udostępnienie systemu kar prezesowi UOKiK-u, w przypadku kiedy już dochodzi do naruszenia prawa i wykorzystania przewagi kontraktowej. Wydaje się nam (Dzwonek), że wprowadzenie tych poprawek - one nie są skomplikowane, są dopuszczone dyrektywą Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Rady - spowoduje, że ta ustawa będzie bardziej życiowa i będzie bardziej efektywna w swoim zastosowaniu. Pamiętam tę dyskusję kilka lat temu, kiedy w podobnym tonie się wypowiadałem, mówiąc, że błędy, które w ustawie sprzed kilku lat są popełnione, będą skutkowały tym, że ona praktycznie nie będzie miała żadnego odniesienia praktycznego. I dzisiaj z perspektywy kilku lat możemy dojść do wniosku, że niestety miałem rację, bo tych przypadków, gdzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainterweniował, wymierzył karę finansową za wykorzystywanie nieuczciwych praktyk, było stosunkowo niewiele. W związku z tym, panie marszałku, składam szereg poprawek. Proszę pana ministra, proszę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o poważne potraktowanie tych poprawek. To nie są poprawki polityczne, tylko merytoryczne, które nam, wam, a przede wszystkim dostawcom do sieci supermarketów pozwolą mieć lepszą pozycję niż dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

A najczęściej tej pozycji nadużywają właśnie międzynarodowe sieci handlowe, które wykorzystują fakt, że są duże, są silne, mają nieograniczony kapitał w przeciwieństwie do polskiego producenta, do polskiego rolnika.

Pozwolę sobie wykorzystać ten czas, ponieważ widzimy problem choćby producentów owoców miękkich, którzy sprzedawali swoje towary poniżej opłacalności. To wychodzi też z tragicznych zapóźnień, zaniechań ze strony ministerstwa. Nie mówię, że to się dzieje od wczoraj, bo poza zwalczaniem pomysłów Komisji Europejskiej dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu - które, mam nadzieję, państwo będą jednak zwalczać, a nie się na to zgadzać - jest jeszcze kwestia choćby rosyjskiego embarga nałożonego na jabłka, a to przekłada się na ogromny problem ze sprzedażą.

Oczywiście też kwestia wzmocnienia naszych rodzimych producentów, tych mniejszych producentów wiąże się z naszymi wyborami konsumenckimi. Apeluję, aby każdy, kto idzie do sklepu, wybierał zawsze polskie produkty. Bardzo dziękuję panu posłowi. Teraz głos zabierze pan poseł Mirosław Suchoń i przedstawi stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050. Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi po przedstawieniu sprawozdania komisji. Szanowni Państwo!

Należy mieć na względzie, i myślę, że wszyscy podzielamy tę opinię, że jeśli chodzi o ukształtowanie rynku w Polsce, na którym działają z jednej strony bardzo silne grupy handlowe, głównie międzynarodowe, ale nie tylko, również nasze, krajowe, a z drugiej strony podmioty producenckie, to jest ono pełne nierówności, cechuje je nierównowaga. Bardzo silne grupy, słabsze grupy dystrybucyjne, słabsze grupy producenckie - to powoduje zaburzenie rynku i zaburzenie pewnej równowagi w zakresie zawierania kontraktów. Takie ukształtowanie rynku sprawia, że te różnice w sile przetargowej powodują skłonność do stosowania właśnie nieuczciwych czy wątpliwych praktyk handlowych. Natomiast warto pamiętać, że jednym z głównych zadań państwa jest dbanie o właśnie to, żeby te warunki udziału, warunki gry handlowej, warunki gry rynkowej były równe dla wszystkich i żeby nie dochodziło do sztucznej nierównowagi, w której potencjał ekonomiczny jednego z podmiotów decyduje o tym, że drugi podmiot zawiera bardzo niekorzystne dla siebie porozumienie dotyczące wspólnych relacji. I ta ustawa ma temu zapobiegać. Myślę, że warto wspomnieć o kilku takich artykułach.

Natomiast narzędzia do kontroli rynku otrzymuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tak naprawdę od urzędu będzie zależało, jak to prawo zadziała i czy będzie skuteczne. Natomiast w toku dyskusji w komisji pojawiła się wątpliwość dotycząca sytuacji małych i średnich polskich przetwórni. W związku z tym Polska 2050 przedstawia poprawkę (Dzwonek), zgodnie z którą taki kontrakt pomiędzy z jednej strony pośrednikiem, nie rolnikiem, ale przedsiębiorcą, który jest pośrednikiem, a z drugiej strony przedsiębiorcą, który jest przetwórcą, będzie możliwy do podziału w takiej strukturze, że 50% płatności będzie do 30 dni po dostarczeniu surowca, natomiast pozostałe 50% - w terminie do 6 miesięcy, wraz z odsetkami i marżą WIBOR. Wydaje się, że to jest sprawiedliwe i bardzo potrzebne dla rynku właśnie małych i średnich polskich przetwórni, które w wyniku przyjęcia tych przepisów mogą po prostu znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Na ręce pana marszałka składam tę poprawkę i proszę o poparcie. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy wystąpienia klubowe i przedstawicieli kół. Do pytań zapisało się 15 posłów. Jeśli ktoś z państwa posłów chciałby się jeszcze do listy dopisać, to zapraszam. Jeżeli nie, to zamykam listę i ustalam czas na zadanie pytania na 1 minutę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałem zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie tego, w jaki sposób zostanie wzmocniony UOKiK, dlatego że to jest bardzo ważny obszar funkcjonowania gospodarki i rzeczywiście trzeba będzie podjąć wiele różnych działań, które zabezpieczą polskich, naszych, zwłaszcza małych producentów.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł. Nie widać, nie słychać. Pan poseł Artur Łącki. Nie ma. Zatem niezawodna pani poseł Małgorzata Pępek. Wysoka Izbo! Procedowana ustawa ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego unijnej dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Niedawna pikieta przed siedzibą jednej z sieci handlowych pokazała, jak bardzo te przepisy są wyczekiwane przez rolników i producentów. Do tej pory dostawca w zasadzie nie był partnerem w procesie uzgadniania warunków dostawy. Sieci, wykorzystując swoją przewagę kontraktową na rynku, wymuszały na dostawcach niekorzystne warunki w postaci niskich cen dostarczania. Przepisy powinny być stosowane najpóźniej od dnia 1 listopada 2021 r., a my procedowaną ustawą wdrażającą dyrektywę zajmujemy się dopiero teraz. Co jest powodem tak długiego opóźnienia? Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Krystyny Skowrońskiej nie widzę na sali. A zatem pytanie zada pan poseł Jan Szopiński. Wysoka Izbo! Bardzo dobrze, że rząd pochyla się nad problemami małych i słabszych ekonomicznie podmiotów w konfrontacji z gigantami dyktującymi warunki obrotu towarowego. Ale niedobrze się składa, że jest to prowadzone w takim tempie. Przeczytam wyjątki z pisma pana ministra do spraw Unii Europejskiej: Należy się spodziewać, że jeżeli dojdzie do wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja będzie w niej wnioskować o nałożenie na Polskę ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej. Z tego też względu należy dążyć do jak najszybszego przyjęcia procedowanych regulacji, niezwłocznego przekazania Komisji Europejskiej informacji o przyjętych przepisach w celu wdrożenia dyrektywy. Z tego miejsca powinien też płynąć apel do Senatu (Dzwonek) o przyjęcie jak najszybciej tej ustawy i do pana prezydenta. Liczę na to, że pan minister wypowie się, dlaczego tak długo trwało procedowanie w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Norberta Kaczmarczyka. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za tę ustawę. Panie ministrze, jednocześnie chciałbym zapytać o prace nad ustawą o podwykonawcach w rolnictwie, która została zainicjowana poprzez współpracę Ministerstwa Sprawiedliwości z ministerstwem rolnictwa. Ta ustawa rzeczywiście ma doprowadzić do sytuacji, w której rolnicy, którzy kontraktują swoje towary, mają pewnego rodzaju zabezpieczenia bankowe. Dzięki temu nie będzie dochodziło do takich sytuacji jak chociażby w 2014 r., kiedy rolnicy zostali pokrzywdzeni przez firmy tytoniowe, które kontraktując u nich towar, surowiec tytoniowy, nie wypłaciły im 15 mln zł, jeżeli chodzi właśnie o te kontrakty, o te należności. Udało się to odzyskać poprzez pomoc de minimis, w postaci 70% tych kwot. Natomiast te ustawy mają dobezpieczyć polskich rolników. Bardzo dziękuję za tę ustawę i proszę powiedzieć (Dzwonek), jakie programy w dalszej kolejności będą dobezpieczać interes polskich rolników. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pani poseł Magdalena Łośko. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tym projektem ustawy rząd potwierdza jedno: wbrew temu, co mówi premier, to, że rosną ceny chleba, to nie wina rosnących cen skupu zbóż i większych zysków rolników, tylko rosnących cen energii elektrycznej, benzyny, gazu, składek ZUS, zwiększonych lub nowych parapodatków oraz przede wszystkim rosnącej inflacji. Być może dzięki temu projektowi premier dowie się, ile kosztuje chleb i ktoś z PiS-u wyjaśni mu, że wyższa cena chleba nie wiąże się wcale z większym zyskiem dla polskiego rolnika. Pytanie jest takie. Zasadnicza jest dla nas informacja, czy ministerstwo przygotowało jakiekolwiek obliczenia lub symulacje dotyczące tego, w jakim stopniu omawiana ustawa przyczyni się do zwiększenia zysków producentów rolnych oraz czy i w jakim stopniu omawiana ustawa będzie miała wpływ na ostateczną cenę produktów rolnych dla konsumentów. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Rafał Adamczyk. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - sam zarys i zamysł są bardzo dobre. Sprawa dotyczy ponad 900 tys. producentów rolnych.

Czemu to jest robione na ostatnią chwilę, 4 miesiące po wyznaczonym terminie? Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Krzysztof Grabczuk. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wsparcie polskich rolników jest obowiązkiem Sejmu Rzeczypospolitej. Dzisiaj w konflikcie pomiędzy rolnikiem a sieciami praktycznie rolnik nie ma najmniejszych szans.

Zawsze jest taka sytuacja, że każdego roku okazuje się, że rolnik czasami z powodu, że ceny są bardzo niskie, nie zbiera danego produktu. W tym roku bardzo dużo rolników nie zebrało czerwonej porzeczki, ponieważ były tak niskie ceny. Oczywiście przed nami, bardziej przed UOKiK-iem wytężona praca, ponieważ po stronie UOKiK-u widzę wciąż bardzo duże możliwości.

Wszystkich państwa zachęcam: kupujcie produkty polskie, a zwłaszcza ze znakiem: Marka Lubelskie. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Paweł Krutul. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mówię w imieniu podlaskich rolników, którzy w ostatnim czasie zgłaszali się do mojego biura poselskiego w Białymstoku. Chodzi o to, żeby skończyć z zalewaniem rynku detalicznego produktami z zagranicy, gdyż przez takie praktyki rodzime rolnictwo polskie nie jest w stanie konkurować, choć polskie produkty pod względem jakości są cenione na całym świecie. Pytam więc: Skąd się wzięły 2 lata zwłoki z wprowadzaniem tych zapisów? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana posła Romualda Ajchlera. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Projekt ustawy, który został przedstawiony, idzie w dobrym kierunku.

Mówił o tych kwestiach pan poseł Maliszewski. Rzeczywiście, ona daje duże uprawnienia UOKiK-owi. Zresztą aktywność pana przedstawiciela UOKiK-u na posiedzeniu sejmowej komisji, kiedy rozpatrywaliśmy różne kwestie dotyczące projektu czy funkcjonowania projektu ustawy, była bardzo dobra. Chciałbym, panie ministrze - i tu mam pytanie - abyście tak korzystali z tej ustawy, która zostanie uchwalona, jaka była pana aktywność podczas posiedzenia (Dzwonek) sejmowej komisji.

Jakie środki wpłynęły? Ostatnia kwestia dotycząca tej ustawy.

Pytanie zada pan poseł Mirosław Maliszewski.

Ja takich podmiotów nie znam. Dostawcy w obawie przed wykluczeniem z rynku po prostu takich pozwów nie składają. To pokazuje, że system tylko i wyłącznie karania za nieuczciwe praktyki bez wzmocnienia pozycji dostawców wobec sieci supermarketów jest systemem nieefektywnym. W praktyce nie będzie on skuteczniejszy od obowiązujących przepisów. Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytania pana posła Czesława Siekierskiego. Panie Marszałku! Problem narasta na skutek koncentracji i monopolizacji po stronie handlu.

Nie wiem, dlaczego brakuje - to jest nie tylko problem Polski - dialogu między rolnikami a odbiorcami. Problem niezorganizowania się rolników jest duży, ale potrzebna jest większa aktywność ministra rolnictwa.

Wobec tego trzeba także zastosować inną politykę wobec sieci handlowych. Ważne, żeby działać na rzecz tworzenia pewnych dodatkowych obiegów dla sprzedaży poza siecią handlową.

To będzie kształtowało pogląd konsumenta, pogląd rolników i pogląd handlowców. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zadanie pytania pana posła Dobromira Sośnierza. Ta ustawa to kolejny bubel, kolejny kawał przeregulowanego, nieprecyzyjnego prawa dającego ogromną władzę arbitralną urzędnikom. Przytoczę fragment: Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Co to znaczy: jest sprzeczne z dobrymi obyczajami?

Już nie można było.

Problem bierze się z przeregulowania rynku. To regulacje powodują nadmierną monopolizację i przewagę kontraktową, a redukowanie tego w taki kazuistyczny sposób jest po prostu absurdem. Na tym zakończyliśmy turę pytań. Teraz proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana ministra Ryszarda Bartosika o udzielenie odpowiedzi.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować wszystkim klubom parlamentarnym, państwu posłom za wstępne poparcie tej ustawy. Dziękuję za wcześniejszą pracę nad tą ustawą. Jak wiemy, projekt ustawy ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Chcę raz jeszcze podkreślić, że w naszym kraju od 2017 r. obowiązują przepisy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Polska jako jeden z pierwszych krajów członkowskich wprowadziła takie przepisy, zanim zostały przyjęte regulacje na szczeblu unijnym. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w wyniku rozszerzenia definicji produktów rolnych i spożywczych, będą mogły również być badane relacje dotyczące skupu m.in. pasz, żywych zwierząt, nasion i owoców oleistych. Przypomnę, że zmianie uległa również definicja nabywcy, którym może być również organ publiczny.

Szanowni Państwo! W wielu państwa wypowiedziach padała kwestia opóźnień związanych z przyjęciem i implementacją przepisów unijnych. Raz jeszcze podkreślę, że w Polsce od 2017 r. obowiązują takie przepisy.

Opóźnienie wynika z tego, że na etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych zgłoszonych zostało wiele uwag, które wymagały wnikliwej analizy i dokonania zmian w projekcie ustawy. Wydłużone zostały konsultacje społeczne z uwagi na szerokie zainteresowanie przedsiębiorców projektowanymi przepisami. Przyjęte w naszym kraju rozwiązania systemowe, tzn. oddzielne przepisy odnoszące się do relacji w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych i oddzielne przepisy w zakresie konkurencji, również wpłynęły na opóźnienie we wdrożeniu dyrektywy.

Regulacje w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych są znane, a do momentu wejścia w życie przepisów projektu ustawy dostawcy produktów rolnych lub spożywczych są chronieni przecież mocą obowiązujących przepisów zakazujących nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Przepisy projektowanej ustawy mają obowiązywać zgodnie z dyrektywą od dnia 1 listopada i wszystko wskazuje na to, że ten termin zostanie dochowany.

Szanowni państwo, w naszym kraju obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych jest wpisany w przepisy prawa. Umowa taka musi zawierać istotne elementy, m.in. cenę, terminy zapłaty.

Taka odpowiedź została skierowana i będzie dostarczona panu posłowi do wglądu.

Utworzona została komórka w UOKiK-u, która jest dedykowana działaniom w zakresie przewagi kontraktowej. Prezes podejmuje odpowiednie działania mające na celu zapewnienie stosownych zasobów kadrowych do realizacji swoich kompetencji i działania w tym zakresie są przez urząd wykonywane.

Jeden z panów posłów pytał, jakie ministerstwo planuje programy i projekty celem zabezpieczenia rolników w przypadku dostarczania produktów w przyszłości. Proponujemy, aby w krajowym programie odbudowy były zaprojektowane przede wszystkim środki, tj. ponad 1 mld euro. Będą interwencje skierowane do podmiotów łańcucha żywnościowego, sektora rolno-spożywczego, w tym do rolników. Ten 1 mld euro, ogólnie rzecz ujmując, zostanie przeznaczony na przetwórstwo, na centra dystrybucyjno-logistyczne, redystrybucję żywności, tworzenie miejsc dla bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

Były pytania o rabaty dystrybucyjne. Nie mamy wiedzy, ile podmiotów wystąpiło na drogę sądową przeciwko takim decyzjom. Nie ma takiego obowiązku, abyśmy taki rejestr prowadzili, niemniej jednak nowa ustawa daje prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów możliwość wspierania rolników w sprawach sądowych w tym zakresie.

Aby warunki współpracy były odpowiednie, podmioty powinny działać na równych prawach.

Wysoki Sejmie! Kontrole w zakresie nieuczciwych praktyk przeprowadza prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast minister rolnictwa nie ma do tego uprawnień, nie ma uprawnień do przeprowadzania kontroli. Były też pytania, czy są informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli. Decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są one publikowane na stronie urzędu. Są to informacje publiczne. Szanowni Państwo! Jak mówiłem na wstępie, ustawa w naszym kraju funkcjonuje. Jej wprowadzenie poprzez implementację przepisów unijnych wprowadza pewne zmiany, ale uczestnicy rynku są przyzwyczajeni do tego rodzaju rozwiązań i przepisów. Rozszerzamy je jeszcze. Żywię nadzieję, że wpłyną one na lepsze stosunki między dostawcami, między odbiorcami, że umożliwią Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolowanie zawierania tych umów, czy są one zgodne z prawem, że wpłynie to bardziej korzystnie na działanie na rynku. Wszystkim państwu dziękuję za ogólne poparcie tej ustawy i proszę o jej przyjęcie. Dziękuję bardzo panu ministrowi.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim członkom komisji, tak Komisji Gospodarki i Rozwoju, jak i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za bardzo merytoryczną pracę w komisji, za zgłaszane poprawki i zgłaszane uwagi.

On wiedział, że zbyt duża konsolidacja kapitału, bo tak naprawdę o tym mówimy, prowadzi do wypaczeń.

To również jest bardzo niepokojące, zwłaszcza w świecie, w którym żyjemy, czyli przy takiej totalnej globalizacji wszystkiego, co tylko możliwe. Oczywiście ta globalizacja jest tłumaczona tym, że ceny będą niższe. Okazuje się, że nie do końca jest to prawda. Jak się głębiej zastanowimy, głębiej popatrzymy na to, co się dzieje w gospodarce, zwłaszcza w gospodarce żywnościowej, to się okazuje, że my za to płacimy dużo drożej.

Poseł Maliszewski mówi: Tak, rzeczywiście mówiłem, że to jest za mało.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druki nr 1590 i 1604) Proszę pana posła Dariusza Olszewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Szanowni Państwo! Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 29 września br. pod przewodnictwem zastępcy przewodniczącego komisji pana posła Marka Matuszewskiego na 73. posiedzeniu przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie, druk nr 1590, a następnie rozpatrzyła projekt i przyjęła sprawozdanie o nim. W procedurze pierwszego czytania uzasadnienie projektu przedstawił minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pan wicepremier Piotr Gliński. Uzasadniając projekt, premier podkreślił, że wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom środowisk sportowych i ma na celu wsparcie karier sportowych członków kadr narodowych, zawodników i trenerów poprzez umożliwienie przyznawania im stypendium sportowego w maksymalnej wysokości do dwukrotności podstawy. W dyskusji nad tym punktem odniesiono się m.in. do kwestii: zapewnienia pomocy materialnej dla sportowców w okresie pomiędzy zawodami i igrzyskami; umożliwienia kontynuacji treningów w związku z zabezpieczeniem sytuacji materialnej; uaktualnienia poprzez projekt świadczenia olimpijskiego - tutaj trzeba podkreślić, że od 2016 r. nie było takiej waloryzacji, ale w 2016 r. ta waloryzacja była; uwzględnienia możliwości objęcia ustawą również świadczeń dla sportowców z katalogu sportów nieolimpijskich i tym samym zapewnienia elastycznej możliwości finansowania sportowców różnych dyscyplin; szczegółowych kryteriów, jakimi wnioskodawcy posługiwali się, zapewniając finansowanie dla poszczególnych rodzajów sportów przewidzianych w projekcie; wreszcie systemowej pozycji i kompetencji Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. Po zakończeniu pierwszego czytania komisja przystąpiła do szczegółowego rozpatrzenia projektu. Do projektu zgłoszono pięć poprawek. Poprawki dotyczyły m.in. kategorii podmiotów, na wniosek których właściwy minister przyznaje stypendium, a także szczegółowego trybu wyboru ofert przez właściwego ministra w zakresie działań związanych z dofinansowaniem sportu. Komisja przyjęła dwie poprawki dotyczące rozszerzenia świadczeń na osoby niezdolne do trenowania na skutek ciąży lub urodzenia dziecka, a także poprawkę legislacyjną, a trzy poprawki odrzuciła. Bardzo dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Marek Matuszewski, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przypadło mi w udziale wystąpienie w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie, druk nr 1590. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że klub Prawa i Sprawiedliwości popiera rządowy projekt ustawy. Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości przyznawania przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, zawodników i trenerów, umożliwienia wzrostu wysokości świadczenia określonego w art. 36 ust. 1 oraz zmiany jego zakresu podmiotowego przez dodanie do katalogu osób uprawnionych do świadczenia reprezentantów Polski na olimpiadzie szachowej. Te rozwiązania, które zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, były bardzo oczekiwane przez środowiska sportowe, olimpijczyków, trenerów. Bardzo się cieszę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan premier wyszedł naprzeciw oczekiwaniom sportowców. Myślę, że te zmiany w ustawie o sporcie jeszcze bardziej podniosą rywalizację, a co za tym idzie, poziom sportu wyczynowego w Polsce. Wymiar ekonomiczny też jest dla sportowców, medalistów, trenerów, sportowców czynnych i tych, którzy już zakończyli swoje kariery, ważny. Tak jak tutaj było powiedziane, zgłoszono do projektu pięć poprawek, trzy zostały odrzucone, dwie zostały przyjęte.

Bardzo dziękuję. Proszę teraz panią poseł Małgorzatę Niemczyk o przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Panie Premierze! Mam zaszczyt w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu nowelizującego ustawę o sporcie. Ten projekt jest krokiem w dobrym kierunku i potrzebnym. Zapewnienie sportowcom i trenerom wsparcia jest niezwykle ważne. Kierunek noweli jest słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Projekt tworzy nowy katalog stypendiów dla trenerów i zawodników, uzupełnia lukę, szczególnie dla młodych zawodników pomiędzy 16. a 23. rokiem życia, a to jest bardzo ważny moment w rozwoju ich kariery. Stypendia muszą być przyznawane w oparciu o wskazania polskich związków sportowych, Instytutu Sportu i ich przyznawanie musi podlegać określonym regułom i zasadom. Nam zależy, aby nie było tutaj uznaniowości. Stąd złożona przez nas poprawka. Bo w sporcie doszło już do centralizacji w wyniku zlikwidowania tzw. kopert wojewódzkich. W wyniku tej centralizacji alokacja środków na infrastrukturę sportową nie jest równomierna i są województwa uprzywilejowane, a utalentowani sportowcy i świetni szkoleniowcy są w całej Polsce. Nie chcemy zobaczyć za rok, że te stypendia dla zawodników i trenerów czy też środki przekazane podmiotom działającym w sporcie w nowym trybie bezkonkursowym będą skoncentrowane znów we wschodnich województwach. Z tego powodu złożyliśmy naszą kolejną poprawkę, gdyż jak czytamy w uzasadnieniu, tryb bezkonkursowy jest potrzebny ministrowi w celu odformalizowania i uelastycznienia wydatkowania środków. Przypominam, że są już narzędzia: dotacje celowe, niewygasy. Do tej pory dużo środków w sporcie było wydawanych w ramach konkursów. Obawiamy się i bardzo się martwimy, czy czasem te środki nie będą wydawane na zlecenia z Nowogrodzkiej. Panie Ministrze! Zapytam jeszcze z drugiej strony: Czy jest zagrożenie, że ten nowy zapis o bezkonkursowym wskazywaniu podmiotów działających w sporcie może spowodować, że sportowe wydarzenia będą organizowane w regionach, gdzie PiS potrzebuje lub będzie potrzebował najwięcej głosów wyborczych lub będzie potrzebował poprawić notowania? W naszej ocenie proponowany zapis przeczy także sprawiedliwości społecznej. Część podmiotów musi przejść pozytywnie konkurs, aby uzyskać środki na realizację, a inne podmioty będą wskazane. Panie ministrze, mam nadzieję, że też pan widzi, że trochę dziwnie to wygląda. Dobrym krokiem w nowelizacji jest podwyższenie wskaźnika stałej bazy dla świadczeń olimpijskich i zwiększenie krotności dla stypendiów. Ważne jest urealnienie świadczeń w wyniku wzrostu cen, opłat czy inflacji. Panie Ministrze! Sprawa nie do końca została omówiona wczoraj na posiedzeniu komisji sportu, z wielkim szacunkiem dla szachów oraz z wielkim uznaniem dla zasług całego środowiska. Wprowadza pan do ustawy o sporcie zapis dla jednej dyscypliny sportu, a z pana ust na posiedzeniu komisji padło, że szachy są na igrzyskach głuchych. Panie ministrze, polski sport ma wielu świetnych sportowców w wielu dyscyplinach sportu. Może warto pomyśleć o stworzeniu nowego katalogu dożywotnich świadczeń dla sportowców nieolimpijskich, w ramach którego będzie możliwość uhonorowania najlepszych i najznakomitszych zawodników. Bo co pan zrobi, jeśli za jakiś czas zapukają do pana gabinetu świetni polscy brydżyści, alpiniści czy przedstawiciele innych sportów? Nie zdołam ich tutaj wszystkich wymienić. Ale niektóre sukcesy chciałabym zaakcentować. Zacznijmy od przypadku Sebastiana Kawy. Trzy medale światowych igrzysk lotniczych, 20 medali mistrzostw świata, dziewięć medali mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik, dwukrotny mistrz świata. Podobnie Aleksandra Mirosław, która specjalizuje się tylko w jednej konkurencji, wspinaczce na szybkość, w której jest dwukrotną mistrzynią świata oraz rekordzistką świata.

Są jeszcze inne, mniej popularne dyscypliny sportu. Trójbój siłowy. W tej dyscyplinie mamy siedemnastokrotnego mistrza świata Jarosława Olecha. Ciekawym przypadkiem jest także bardzo dynamicznie rozwijająca się, bo efektowna dla kibiców, dyscyplina narciarstwo wodne. Nasza reprezentacja wywalczyła pięć medali indywidualnych i dwa drużynowe. Na koniec wspomnę sport motorowodny. Wczoraj komisja przyjęła poprawkę dającą ochronę stypendystkom: członkiniom kadr narodowych, zawodniczkom, trenerkom w okresie ciąży oraz przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Ta poprawka to od dawna postulowany głos środowiska sportowego, głos kobiet, zawodniczek, trenerek. Mamy nadzieję, że ta poprawka zostanie przyjęta przez komisję. Jak mówiłam na wstępie, klub Koalicji Obywatelskiej wspiera rozwój sportów w Polsce. Ale już dzisiaj obiecujemy, że będziemy się bacznie przyglądać każdej złotówce wydawanej w nowych trybach stypendialno-konkursowych. Wnosimy o poparcie i prosimy, żeby to wszystko było transparentne, jeśli chodzi o wydawanie środków publicznych na sport. Sport powinien być apolityczny, równo rozwijający się w całej Polsce i na takich samych zasadach. Nie powinno być obszarów, regionów ani podmiotów bardziej uprzywilejowanych. Bardzo dziękuję, pani poseł. Proszę teraz pana posła Tadeusza Tomaszewskiego o przedstawienie stanowiska klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Nie dostrzegam w nim cech walki politycznej. Możemy w tej Izbie przyjąć rozwiązania zawarte w tej ustawie ponad podziałami politycznymi.

Wielu z nich ginęło, ze swoimi osiągnięciami nie dochodziło do wieku seniora. Ta kwota również jest zwiększona do dwukrotności podstawy, czyli podstawa wynosi 2300 zł, to kwota bazowa. Po drugie dlatego, że te stypendia, wszystkie razem, będą w gestii ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, czyli będą prowadzone i wypłacane przez Instytut Sportu.

Dziś we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez ministerstwo uczestniczy blisko 90 tys. młodych zawodniczek i zawodników z blisko 5 tys. klubów, więc to jest potencjał, w którym można łapać perełki. To przewiduje ta ustawa. Ponadto to jest kwestia zwiększenia kwoty świadczenia olimpijskiego. Ale chcę też wspomnieć, że w 2015 r. na tej sali opozycja zaproponowała zwolnienie tych świadczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych. Miałem zaszczyt zgłosić ten wniosek i prowadzić tę ustawę. Prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę i od 2016 r., szanowni państwo, te świadczenia są świadczeniami honorowymi, tak jak powinno być. Medalista olimpijski ma świadczenie honorowe, zwolnione przez polskie państwo z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ale chciałem przypomnieć tym, którzy może nie pamiętają, że kiedy z tej Izby udało nam się projektem komisyjnym wprowadzić świadczenia dla medalistów olimpijskich, a później paraolimpijskich, światowych igrzysk głuchych - dzisiaj rozszerzamy je dla medalistów olimpiady szachowej - wówczas to świadczenie wynosiło średnią obliczaną do celów ZUS-u.

Ale po drodze zgubiliśmy tę wartość. Mówię o parlamencie, rządzie. Szanowni Państwo!

Poprawka ówczesnego prezesa PKOL, posła klubu SLD mówiąca o tym, że wprowadzamy to i dla wszystkich tych, których zdobyli medale, i dla tych na przyszłość, uzyskała większość tamtej Izby i od tamtego czasu to rozwiązanie funkcjonuje. Panie Premierze! Ta ustawa jest na szóstkę, minus poprawka nr 1. W poprawce nr 1 pan minister mówi, że jako jedyny z wszystkich rządzących chce mieć wszystkie pieniądze dostępne bez procedury konkursowej.

Zostały tylko pieniądze budżetowe, te pozostałe, które tym rozwiązaniem będą zwolnione. To nie jest coś, co by dyskwalifikowało tę ustawę, ale budzi wątpliwości.

Dlatego też zgłaszamy tę wątpliwość, uważając, że takie rozwiązania powinny być wprowadzane ostrożnie, zwłaszcza po konsultacjach społecznych z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi. Klub parlamentarny Lewicy wesprze to rozwiązanie, będzie głosował za zmianą ustawy o sporcie. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz pana posła Ireneusza Rasia o przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, druk nr 1590, a druk przedłożenia rządowego - nr 1604.

Nie doszukuję się w nich zmian, które w innych obszarach tak często spotykamy na tej sali. Uważam je za mądre również z mojej perspektywy.

Uważam, że ona się wpisuje w logikę ustawy z 2010 r., która w ogóle na nowo opisywała zaangażowanie sfery publicznej w polski sport. Podobają mi się te zmiany, ponieważ są komplementarne. Bardzo mi się podoba, że odchodzimy od tej protezy, panie premierze, którą wykorzystywał minister sportu, jeśli chodzi o finansowanie najpierw Klubu 100, a potem jeszcze tego rozrośniętego klubu przez Polską Fundację Narodową. Uważam to za absolutnie cenne i właściwe.

Podejmują te decyzje. Więc to na pewno będzie narzędzie absolutnie sprzyjające. Według mnie bardzo dobrą rzeczą jest wreszcie powiązanie bardziej do tego procesu wnioskowania o stypendia dla polskich sportowców Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego, dlatego że od dawien. Zawsze powtarzaliśmy, od wielu lat, że trzeba przebadać polskich sportowców, żeby poznać ich motorykę, ich możliwości osiągania wyników w perspektywie i dzięki temu w sposób łatwiejszy, gdy będziemy korzystać z nauki, będziemy mogli powiedzieć: Tak, w biegach narciarskich ta osoba może uzyskać taki, a nie inny wynik, a w innych sportach to ta osoba ma lepsze predyspozycje. Nauka ze sportem musi być powiązana. Oczywiście stypendia, które umożliwiają ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej wsparcie zawodników, którzy znaleźli się w szczególnie złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, a którzy chcą kontynuować karierę sportową, też to jest zapis niebudzący żadnych wątpliwości, bo są przypadki losowe, długotrwałe kontuzje. Pan minister to w uzasadnieniu wypisywał. Z tym się trzeba zgodzić. Konflikty z działaczami sportowymi, też znamy ich trochę. Przerwa w karierze sportowej. Ale ta poprawka, proszę się zastanowić, pani poseł Niemczyk, może trochę zmodyfikowana, byłaby fajnie czytana, żeby te sportsmenki i trenerki, które są na odpowiednim poziomie, zachodzą w ciążę, nie jest tych przypadków przecież tak wiele. Oczywiście przepisy, które pan proponuje, dają taką możliwość, ale rozumiem, że temat jest otwarty i myślę, że gdyby się jakieś powtórzenie znalazło, to nie byłoby takie złe. Jeżeli chodzi o kwestię świadczeń olimpijskich, to waloryzacja jest jak najbardziej właściwa. Za medale w olimpiadach szachowych. Szachy mają pewien potencjał niewykorzystany, jeżeli chodzi o proces edukacyjny, więc też to popieramy.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi.

Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Pojawiające się tam przepisy, tak jak przyznanie medalistom w olimpiadzie szachowej bliźniaczych świadczeń z tymi, które otrzymywali - w cudzysłowie - zwykli medaliści olimpijscy, to dobry krok. Zwłaszcza w kontekście ostatnich sukcesów Polaków. Gratulacje z tego miejsca dla pana Jana Krzysztofa Dudy, który jako pierwszy zdobył puchar świata w szachach. Będzie to nie tylko nagroda dla tych zasłużonych, ale także zachęta dla osób młodych, które chcą się rozwijać w tej dziedzinie. Będą one wiedziały, że w swoich marzeniach i ambicjach są wspierane. Dzięki temu więcej osób podejmie się treningów i przez to reprezentowania Polski na wyższym poziomie. Oby te środki trafiły do nich bez politycznych rozdań. Także osoby, które wcześniej nie mogły sobie pozwolić na poświęcenie się sportowi, po wejściu w życie ustawy będą miały możliwość skupienia się i profesjonalnego trenowania. Pozwoli to wyrównać szanse reprezentantom Polski z tymi z innych najlepszych krajów, w których podobne świadczenia funkcjonują. Uruchomi dodatkowy potencjał drzemiący w Polakach. Wsparcie dla sportowców należy pochwalić, jednak trzeba zwrócić uwagę na kontekst. W Polsce panuje drożyzna, benzyna kosztuje już niemal 6 zł, gaz samochodowy 3 zł, cena chleba wzrosła w zeszłym roku 25% względem tego samego miesiąca rok wcześniej. Może dlatego pan premier nie zna ceny chleba. Ceny mieszkań urosły do poziomu europejskiego. Niestety, nie równomiernie do wzrostu płac. Rządzący powinni dbać o zwiększenie dobrobytu wszystkich obywateli, a nie o zwiększanie podatków i dobrobytu rządu i dbania, dopieszczania ekonomicznego wyłącznie swojego elektoratu. Ale wracając do sportu: należy wspierać sportowców, zwłaszcza młodych, i propozycja zawarta w tej ustawie, by można było przyznać stypendium już 16-latkowi, jest dobra. Pomijając trudności związane z wchodzeniem w dorosłość takiego człowieka, to jest kluczowy czas dla kariery sportowej, również ze względu na zbliżające się pierwsze występy w kadrze seniorskiej. W kontekście poprawnego wychowania młodzieży pochwalić należy odebranie stypendium z mocy prawa w chwili przyłapania na dopingu czy z chwilą skazania za przestępstwo umyślne. Przepis ten oprócz ukarania sprawców pełni także rolę wychowawczą potępiającą osoby postępujące wbrew etyce. Podsumowując, zależy nam na wychowaniu narodu, szczególnie młodzieży, w duchu zwalczania własnych słabości, w duchu rozwoju nie tylko duchowego, ale również z dużym naciskiem na rozwój fizyczny i intelektualny, a wszystko to w zgodzie z zasadami fair play, bez oszustw, dopingu, używek.

Stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 przedstawi pan poseł Tomasz Zimoch. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! Sport łączy i jest ponad podziałami. Pokazują to prace nad projektem tej ustawy. Pan minister woli sprint od biegów długodystansowych, szybkie procedowanie, ale to w tym przypadku jest ogromnym atutem. Brawo. Nie pamiętam, kto jest autorem słów, że sport jest siłą zbawczą tego świata, ale to celne stwierdzenie. O zbawienie należy się troszczyć. Sport zatem należy dowartościowywać. Dlatego ze strony Koła Parlamentarnego Polska 2050 jest poparcie dla tej ustawy, czyli poparcie m.in. dla - by się nie powtarzać - dofinansowania sportowców, przyznawania stypendiów młodym, zdolnym zawodnikom, ale także często niedostrzeganym trenerom. Popieramy oczywiście zwiększenie emerytury dla medalistów olimpijskich, także pomoc dla tych sportowców, którzy często nie z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Mamy nadzieję, że dofinansowanie sportu nie będzie w sprzeczności z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dlatego ponawiamy naszą poprawkę, a drugą składamy w związku z przyznawanym Instytutowi Sportu prawem wnioskowania o wsparcie stypendialne. Panie Premierze! Gorąco popieramy, i to od dawna, potrzebę naukowego wsparcia sportu i sportowców. Ale instytut niech pozostanie ośrodkiem badawczym, a nie zastępuje trenerów i związki sportowe. Nawet proponujemy jako koło następny krok - może pan, panie premierze, przekona także ministra Czarnka, by szachy stały się obowiązkowym przedmiotem w szkołach podstawowych. Szukajmy w szkołach cnót właśnie szachowych. Szachy są żywiołem dla milionów. Frank Marshall, zwycięzca olimpiad, arcymistrz amerykański, niemal 100 lat temu powiedział, że szachy uczą życia, uczą, jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się wycofać, żeby potem ruszyć do ataku - i właśnie na tym polega urok tej królewskiej gry. Ta ustawa pomaga nie tylko szachistom. Raz jeszcze słowa uznania.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam wielką przyjemność w imieniu mojego środowiska politycznego przedstawić stanowisko na temat nowelizacji ustawy o sporcie. Popieramy ten projekt, popieramy ten kierunek i cieszymy się, że sport jest właśnie tym momentem, tym elementem, w przypadku którego można ponad podziałami porozmawiać o tym, co dobre, i wspólnie wypracować lepsze stanowiska. Przez lata środowisko sportowe wskazywało na potrzebę większego wsparcia sportowców, zwłaszcza tych, którzy w momencie dochodzenia na szczyt są w najtrudniejszej sytuacji finansowej.

Zwraca się uwagę na sportowców, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji finansowej - także należy pochwalić ten kierunek.

Panie Premierze! Przez lata polskie środowisko sportowe zwracało uwagę na konieczność większego dofinansowania właśnie tych, którzy w tej trudnej drodze na szczyt, bogatej w wiele wyrzeczeń i trudnych decyzji, potrzebują szczególnego wsparcia. Ten projekt jest krokiem w dobrym kierunku. Popieramy ten projekt, liczymy na więcej. I jeszcze raz w imieniu mojego środowiska politycznego powiem: cieszę się z tego powodu, że cała sala sejmowa, i myślę, że środowisko sportowe w Polsce też, podziela to zdanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Ta wypowiedź kończy prezentację stanowisk klubów i kół. Przystępujemy do zadawania pytań. Bardzo proszę, jeśli ktoś z państwa posłów chciałby jeszcze dopisać się do listy, to jest ta możliwość. Proszę bardzo. A zatem po dopisaniu się pana posła Baszki zamykam listę posłów zadających pytania. Ustalam czas na zadanie pytania na 1 minutę. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Mirosław Suchoń. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To bardzo często kończy się tym, że albo wyniki sportowe tych osób ulegają pewnej stabilizacji, albo z drugiej strony czasami takie osoby rezygnują, bądź na stałe, bądź też na jakiś czas, i odchodzą z dyscypliny, co oczywiście - widać to w sposób bardzo jasny i czytelny - nie powinno mieć miejsca. W związku z tym chciałem zapytać pana ministra, jakie rozwiązania zostaną wdrożone, tak aby z tych stypendiów mogły właśnie korzystać również takie osoby, które znajdują się pod jakąś presją i być może w taki bardzo delikatny, a czasem gwałtowny sposób (Dzwonek) są przez środowisko odsuwane do tego głównego nurtu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Tadeusz Tomaszewski. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Premierze! Ustawa mówi o tym, że na realizację jej przesłania, czyli na podwyżki świadczeń medalistów olimpijskich oraz rozszerzenie stypendiów, zabezpieczona jest kwota 51 mln zł przez najbliższe 10 lat w każdym budżecie. Po pierwsze, chcielibyśmy wszyscy razem, żeby liczba medalistów olimpijskich, paraolimpijskich, światowych igrzysk głuchych i od ostatniego czasu olimpiad szachowych rosła.

Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią poseł Jagnę Marczułajtis-Walczak. Wysoka Izbo! Polski sport jest mocno niedofinansowany, więc każdą złotówkę w kierunku sportu i sportowców należy przyjąć z radością. Niemniej jednak obawy budzi zapis, który umożliwi ministrowi sportu realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kto będzie miał nadzór nad tym, do kogo i na co trafią te pieniądze? Panie Ministrze!

Czy utrzymacie tę poprawkę, czy może w trzecim czytaniu zagłosujecie przeciw? To niewielki koszt dla budżetu państwa, a wielka pomoc dla naszych zawodniczek i trenerek. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo pana posła Norberta Kaczmarczyka. Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o sport i politykę, to mówi się, że wszyscy polscy obywatele znają się na tym najlepiej. W ogóle w tej walce politycznej pokazujemy różne stanowiska. Dzisiejsza debata pokazuje, że rzeczywiście dofinansowania dla sportu łączą. Chciałbym zapytać przy tej okazji pana premiera o sytuację, w której będzie możliwość dofinansowania również obszarów wiejskich, jeżeli chodzi o te stypendia. Czy planowane są programy wdrożeniowe, które pozwoliłyby na dofinansowanie chociażby zakwaterowania czy zwrot kosztów podróży dla tych osób? Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Krzysztof Grabczuk. Wysoka Izbo! To jest projekt ustawy, który zmierza w dobrym kierunku, bowiem sport to piękno, sport to szacunek dla przeciwnika, sport uczy pokory, sport uczy ciężkiej pracy, ale pamiętajmy, że sport to również wielka promocja naszych miast i naszego kraju, sport to duma.

Talent - bogactwo narodu.

Uważam, że gdybyśmy przenieśli przynajmniej część zachowań, które obowiązują w sporcie (Dzwonek), do polityki, nasze życie polityczne byłoby dużo piękniejsze. Panie premierze, sport to reguły i zasady. Musimy tych reguł przestrzegać, zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie, bo jeśli nie będziemy ich przestrzegać, zaszkodzi to wszystkim tym, którzy uczestniczą w życiu sportowym. Pytanie zada pan poseł Jan Szopiński.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo dobra ustawa, ale. Minister będzie mógł skorzystać z trybu zlecania realizacji zadań publicznych w formie dofinansowania wszelkich działań związanych ze sportem. Dotychczasowa praktyka wzmocniona doświadczeniami pandemii wskazuje na konieczność wypracowania elastycznego podejścia do kwestii dofinansowania zadań z zakresu sportu. Chciałbym uprzejmie prosić pana, panie premierze, żeby pan powiedział, z którymi związkami i stowarzyszeniami sportowymi konsultował pan takie rozwiązanie.

Gdyby pan opowiedział mi w tej sprawie na piśmie, to będę panu zobowiązany. Do pani poseł Wolskiej, do całej listy wybitnych sportowców, którzy zdobywali medale dla polskiego sportu (Dzwonek), chciałbym dołożyć imię i nazwisko Jana Wróblewskiego, dwukrotnego mistrza świata w szybownictwie w latach 70., a przypomnieć należy, że wtedy mistrzostwa odbywały się co 4 lata. Być może dla tych sportowców, którzy osiągnęli już określony wiek, tak jak pan Jan, znajdą się jakieś rozwiązania, które docenią ich sportowe dokonania. Pytanie zada pan poseł Jakub Rutnicki. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Im więcej pieniędzy dla polskiego sportu, tym lepiej. Ale już wielokrotnie podczas dzisiejszej debaty padało, że sport to przede wszystkim gra fair play. Chodzi o to, panie premierze, że rzeczywiście są pewne zmiany, które nie dają pewności, w jaki sposób te środki będą przyznawane. Dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniu komisji, ale niestety, panie premierze, mamy złe doświadczenia, jeżeli chodzi o Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, bo przypominam: to była zła decyzja - likwidacja kopert wojewódzkich, co wpłynęło na to, że niestety poszczególne województwa różnie są, nazwijmy to, nagradzane, jeżeli chodzi o poszczególne inwestycje sportowe. Mówiła o tym pani poseł Niemczyk: wszyscy szanujemy szachistów, to jest rzecz oczywista, ale też mamy wielu wybitnych sportowców. Za chwilę będą brydżyści, za chwilę będzie wiele innych osób, które być może z perspektywy czasu po prostu będą potrzebować pomocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Kiedyś w tej Izbie było kilka kwestii ponad podziałami, m.in. polska polityka zagraniczna, obronność państwa.

Wtedy nam odpowiedziano, że nie ma środków. Przeszliśmy ogromną drogę, bo po 2000 r. taką ustawę lewica przyjęła, a dzisiaj rozszerzamy to o kolejnych sportowców, którym chcemy pomóc. Była teza, że niewidzialna ręka rynku wszystko załatwi, państwo nie musi się interesować sportem czy innymi dziedzinami, a dzisiaj widać, że można to zrobić.

Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Maciej Lasek. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Pozwolą państwo, że przytoczę kilka liczb. Samolotowe mistrzostwa świata w lataniu precyzyjnym, klasyfikacja medalowa, Polska na pierwszym miejscu, 34 złote medale, 20 srebrnych. Rajdowo-nawigacyjne mistrzostwa świata, w klasyfikacji medalowej Polska na pierwszym miejscu, 27 złotych medali, 22 srebrne, 13 brązowych. Szybowcowe mistrzostwa świata, Polska na drugim miejscu, 25 medali złotych, 18 srebrnych. Przytoczyłem tylko niektóre z dyscyplin, sportów lotniczych, w których jesteśmy najlepsi. Panie ministrze, chyba nie ma wielu dyscyplin sportowych, w których Polacy zdobyliby tyle medali i tytułów mistrzowskich, co w sportach lotniczych. Na jaką pomoc mogą liczyć lotnicy sportowcy, którzy rozsławiają polskie skrzydła na świecie? Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Każde dodatkowe dofinansowanie to bardzo, bardzo dobra wiadomość, jednak, panie ministrze, tryb bezkonkursowy to chyba wolne żarty. Prawo i Sprawiedliwość niejednokrotnie udowodniło, że dofinansowania kierowane były do działaczy, sympatyków związanych z państwa ugrupowaniem. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Tomasz Zimoch. Wysoki Sejmie!

Pytanie drugie.

Chodzi o to, ile to jest osób, które otrzymują to świadczenie honorowe, o którym tak pięknie powiedział poseł Tomaszewski (Dzwonek), oczywiście z podziałem na olimpijczyków, paraolimpijczyków, głuchych itd. Proszę o zadanie pytania panią poseł Małgorzatę Niemczyk.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Poproszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Wczoraj na posiedzeniu komisji sportu w ramach udzielania odpowiedzi pan, panie premierze, powiedział, że dzięki nowemu trybowi pozakonkursowemu ministerstwo, czyli pan będzie mógł dać podmiotom działającym w sporcie środki publiczne na realizację zadań podmiotowych, które odpadły w konkursie, chociażby ze względów formalnych. Panie Premierze! Jest to określenie nieostre, nie funkcjonuje ono w żadnym dokumencie w polskim systemie prawnym, który jest obowiązujący. Jaka będzie możliwość odwołania się od decyzji, jeżeli będzie ona wydana na podstawie karty olimpijskiej?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sport łączy, a nie dzieli, i to było widać po dzisiejszych wystąpieniach, może z małymi wyjątkami. Wielki szacunek dla pana premiera za tę bardzo dobrą ustawę. Bo ci, co tak delikatnie, ale jednak krytykują pana premiera, jak myślę, robią to nie z powodów merytorycznych, a tylko politycznych. Dziś trzeba się cieszyć, że tak dobre projekty ustaw są dla środowiska sportowego tworzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Na sport w Polsce przeznaczane są ogromne środki, bo te środki zaprocentują. Panie Premierze!

Dziękuję bardzo. Proszę panią poseł Agnieszkę Hanajczyk. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Dudzie nie tylko niebywałych światowych sukcesów, ale też tego, że niewątpliwie był sprawcą tych bardzo potrzebnych, pożądanych i cieszących zmian.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w zakresie działań związanych z dofinansowaniem sportu może zlecić podmiotom wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nie zakładam, panie premierze, że to będzie dotyczyło dziedziny sportu, ale taka pokusa może wystąpić w odniesieniu do pieniędzy, które w sposób niekontrolowany, nieprzejrzysty, nietransparentny, poza konkursem ofert zostaną przekazane do podmiotów. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Mieczysław Baszko. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! No cóż, tylko trzeba pochwalić taką ustawę, która została przygotowana, procedowana była na komisji.

Cieszę się bardzo, że sporty umysłowe są zauważone przez pana ministra. Bardzo dziękuję. Listę posłów zapisanych do pytań zamyka pan poseł Dobromir Sośnierz.

A więc cóż stoi na przeszkodzie dalszej hojności? Rozrywki, gry, zabawy, tańce, hulanki, swawole. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo. Tak to nieraz bywa, pani poseł, że dobra wola jest nadużyta. Proszę o odniesienie się do wystąpień oraz pytań wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pana Piotra Glińskiego. Bardzo proszę, panie premierze. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w pracach nad tą ustawą, także tym, którzy wypowiadali się teraz w dyskusji. Dziękuję, bo zdecydowanie większość z nas ma chyba podobną opinię na temat tej ustawy. Widziałem tutaj, co faktycznie może nie jest zbyt częste na tej sali, znacznie więcej dobrej woli niż złej woli, choć pewne elementy, powiedziałbym, niezrozumienia cały czas są powtarzane. To mnie trochę martwi, bo znaczy, że zupełnie nie mam żadnych talentów dydaktyczno-eksplanacyjnych, bo powtarzam, powtarzam i powtarzam, a niektórzy z państwa też powtarzają - cały czas to samo. Jeszcze raz powtórzę, powiem, o co chodzi. Dziękuję oczywiście. Te podziękowania należą się także środowisku sportowemu.

Bardzo się cieszę, że też udało się je włączyć.

Dziękuję bardzo. Zacznę od pewnych nieścisłości, żeby je na początku wyjaśnić. To jest tylko tryb, który się nie odwołuje do definicji otwartego konkursu ofert z pewnej ustawy, której notabene byłem współautorem przed laty jako działacz społeczny, działacz organizacji pozarządowej. Dlaczego? Dlatego że w praktyce pracy ministerialnej ten tryb się nie do końca sprawdza.

Kto wtedy rządził i kto to rozporządzenie przygotował?

To m.in. kryteria, terminy, wysokość naboru itd. Jest to faktycznie prostsze rozwiązanie niż ten skomplikowany i trudny do realizacji, zwłaszcza pod koniec roku, jak się uwalniają środki budżetowe - kto się zajmował pracą w ministerstwach, wie, o czym mówię - tryb. Codziennie. Chcemy wprowadzić to także dla tych projektów.

Tak bywa. Praktyka, tylko i wyłącznie praktyka zadecydowała o tym, że chcemy uprościć ten tryb. Nie zgodzi się Sejm? Trudno. Będzie trochę trudniej, ale będziemy dalej to realizowali.

Ustalmy to raz na zawsze. Inne nieścisłości, które tu padały.

Piękne są szybowce. Tak, wielkie osiągnięcia.

Między nami mówiąc, ten sport olimpijski, jakim są szachy, jeszcze raz przypominam, wygenerowałby świadczenia dla pięciu osób. Miałbym szacunek dla tego, co pan mówi, gdyby. Dobrze, nie będziemy tego kontynuowali, panie pośle.

Już ją uprawia. Ona jest już włączona. Pani Poseł! Myśmy prostowali. Wspinaczka, jedna z trzech dyscyplin alpinistycznych, została włączona do programu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jest to dyscyplina olimpijska, więc w ogóle nie ma sensu o tym dyskutować. Zarzut dotyczący Instytutu Sportu.

Nie słyszałem żadnych zarzutów co do tego programu. Właśnie Instytut Sportu pewnie to gwarantował. Przypominam, że Instytut Sportu jest usytuowany przy ul. Trylogii, a nie przy ul. Nowogrodzkiej, i to też nieprzypadkowo, ponieważ Instytut Sportu jest wyspecjalizowaną jednostką, która będzie najlepszym operatorem dla tych programów, które chcemy wprowadzić. Tam było nieco ponad 10 mln, włączając pieniądze operacyjne. Jeżeli tu mamy cztery nowe programy, to cztery razy 10 równa się 40 plus pieniądze operacyjne.

Jeszcze taka kwestia z tych poważniejszych, kwestia przedłużenia stypendiów dla pań, które zachodzą w ciążę i zmienia się ich sytuacja życiowa.

To stypendium może dostać ktoś, kto już jest w ciąży. To stypendium, które wprowadzamy, jest jedynym stypendium po raz pierwszy wprowadzonym, którego kryteria wprowadzenia nie są związane bezpośrednio z wynikami sportowymi, a z całokształtem sytuacji życiowej.

To już jest kwestia decyzji indywidualnych itd. I takie stypendium może dostać od ministra. To wprowadzamy, czyli ta opieka jest, pani poseł. Po raz pierwszy coś takiego robimy. Mam jeszcze trochę czasu.

Są koszty kwalifikowane, tego nie można wydać na papierosy, powiedzmy sobie, ale właśnie na mieszkanie, na dojazdy. Te systemy stypendialne przecież po to robimy, żeby obejmowały mieszkańców całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób, dla których takie wsparcie jest zasadnicze. Przypominam, Kajetan Duszyński, rozmawialiśmy przy jakiejś okazji po zdobyciu złotego medalu, powiedział, że gdyby on nie miał stypendium Team 100 z Polskiej Fundacji Narodowej, toby nie pojechał do Tokio, bo to było jedyne stypendium, które on dostał, i to tylko rok przed igrzyskami olimpijskimi. Takie sytuacje były. Pan Dawid Tomala, który doszedł do złotego medalu, pracował na budowie.

Tak, odpowiadam, przygotowujemy także szerszą nowelizację, na posiedzeniu komisji o tym mówiliśmy. Zbieramy różne postulaty, tak że jesteśmy otwarci na postulaty z wszystkich stron. Z góry mówię, że kwestii tych rydwanów nie będę rozpatrywał, panie pośle, ale oczywiście możemy dalej dywagować na tym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o wsparcie, to też przy okazji powiem państwu, że oprócz tych 44 mln na te rozwiązania tutaj i na świadczenia, czyli 51 mln, łącznie w przyszłym roku, z czego jestem w jakimś sensie dumny czy zadowolony, zwiększyliśmy budżet sportu o 284 mln. To jest mniej więcej prawie połowa tego wzrostu, który przez ostatnie 6 lat nastąpił. Dzięki temu większość tego, żeby było też jasne, idzie na sport powszechny, nawet więcej niż na wyczynowy, niewiele więcej, bo to jest zrównoważone mniej więcej wsparcie wszystkich naszych programów. Może przy innej okazji.

Jest to najwyższe finansowanie dla dyscyplin nieolimpijskich w naszym resorcie. Mam nadzieję, że płynnie i szybko przeprowadzimy tę ustawę, bo chcielibyśmy, i to też jest ważne, od stycznia wprowadzić te programy, żeby one działały. Dziękuję bardzo panu premierowi. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Ogłaszam 15 minut przerwy. Proszę bardzo.

Bardzo podobny jest przykład Aleksandry Mirosław, która brała udział w igrzyskach, ale w programie olimpijskim znajduje się konkurencja łącząca wszystkie specjalności wspinaczkowe, natomiast pani Aleksandra Mirosław specjalizuje się tylko w jednej konkurencji - wspinaczce na szybkość, gdzie jest dwukrotną mistrzynią świata oraz rekordzistką świata. Dziękuję bardzo.

Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdań komisji zawartych w drukach nr 1615 i 1616. Wysoka Izbo!

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła w dniu dzisiejszym te projekty ustaw. Jeśli chodzi o ustawę zmieniającą ustawę budżetową na rok 2021, komisja przeanalizowała wszystkie zmiany wydatkowe, ale przede wszystkim skupiła się na stronie dochodowej. Wiele było pytań dotyczących tego, skąd wzięły się te dochody, można by powiedzieć, jakim sposobem w tym roku mamy dochody planowane w tej chwili w nowelizacji o prawie 80 mld większe, niż były w ustawie budżetowej uchwalonej na początku roku na 2021 r. Z dyskusji wynikało, że te dochody budżetowe pojawiły się w znacznej części dzięki temu, że rząd prowadzi odpowiedzialną politykę gospodarczą, w okresie pandemii COVID nie wzrosło bezrobocie dzięki pomocy dla firm w różnej formie, zarówno z PFR-u, jak i z ZUS-u, ale też i z innych instytucji, urzędów pracy, stąd zachowane miejsca pracy pozwoliły na bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy w tym roku i stąd znaczące dochody. Jeśli chodzi o poprawki, które komisja rozpatrzyła, to było zgłoszonych kilka poprawek, m.in. przyjęto dwie poprawki w części tabelarycznej, które zmieniały, właściwie przesuwały środki finansowe w obrębie części sprawy wewnętrzne w kwocie 20 mln z przeznaczeniem na ochronę zdrowia, w obrębie części sprawy wewnętrzne, i ponad 260 mln na doposażenie służb mundurowych, m.in. Policji, straży pożarnej i Straży Granicznej, czyli na wydatki majątkowe. Te zmiany były dokonane w obrębie jednej części budżetowej na zasadzie przesunięcia.

To tak naprawdę de facto zwiększenie środków na wynagrodzenia na rok 2021 o 6%, a więc jest to bardzo znacząca kwota, stąd m.in. ta ustawa okołobudżetowa pozwala na wykorzystywanie tej kwoty zarówno w roku 2021, jak i w roku 2022. Jeśli chodzi o poprawkę, która została przyjęta w ustawie okołobudżetowej, to poprawka rozszerzała podmioty uprawnione do skorzystania z tego zapisu m.in. o państwowe jednostki prawne, agencje, aby te wszystkie podmioty również mogły korzystać z tych warunków 6-procentowego dodatku motywacyjnego jak inna administracja. Obydwie ustawy komisja zaaprobowała i rekomenduje Wysokiej Izbie ich przyjęcie.

Szanowny Panie Marszałku!

Nie będę ich powtarzał. Oczywiste jest, że klub Prawo i Sprawiedliwość gorąco popiera ten projekt ustawy. Cała ustawa i nowelizacja budżetu to jasny dowód na znakomicie prowadzoną politykę gospodarczą rządu Prawa i Sprawiedliwości. Warto podkreślić jeszcze raz, że jest to bardzo głęboka zmiana.

Panie Marszałku! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę złożyć jedną poprawkę.

Oczywiście klub Prawo i Sprawiedliwość będzie popierał tę ustawę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Teraz w imieniu klubu Koalicja Obywatelska pan poseł Dariusz Rosati.

Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska ma bardzo wiele zastrzeżeń wobec projektu nowelizacji budżetu na 2021 r. z kilku powodów. Po pierwsze, wbrew temu, co powiedział pan przewodniczący Kowalczyk, dodatkowe dochody, jakie pojawiają się w budżecie, nie są wcale wynikiem fantastycznej polityki gospodarczej rządu Mateusza Morawieckiego. Krótko mówiąc, nie są zasługą rządzącej większości.

Już w trakcie dyskusji w pierwszym czytaniu wskazywałem na te mankamenty. Państwo zaniżyli dochody budżetowe zarówno w nowelizacji budżetu na 2020 r. - dokładnie rok temu - jak i w projekcie budżetu na 2021 r. - również dokładnie rok temu. Wbrew temu, co pan mówi, panie przewodniczący, można sięgnąć do stenogramu, z którego pan się dowie, że posłowie Koalicji Obywatelskiej ostrzegali, że dochody są zaniżone i wskazywali na to, że trzeba je podnieść. Jest też inna interpretacja, że nie było to zrobione w sposób świadomy, tylko wynikało z nieudolności. Zostawiam państwu wybór interpretacji faktu, który pozostaje bezsporny: dochody zostały zaniżone.

Do tego dochodzi wyższa inflacja w tym roku, za którą ponosicie odpowiedzialność.

Macie państwo z tego tytułu 38 mld zł. Nie wspomniał pan, panie przewodniczący, że zarobiliście także na sprzedaży pozwoleń na emisję.

Wreszcie, macie 7 mld zł dodatkowego zysku z Narodowego Banku Polskiego, który dwoi się i troi, żeby wesprzeć rząd Zjednoczonej Prawicy, oczywiście kosztem wzrostu inflacji.

Efekt jest taki, że rzeczywiście więcej jest pieniędzy w budżecie. To jest główny powód, dla którego nie będziemy głosować przeciwko tej nowelizacji, bo jeżeli rzeczywiście jest więcej pieniędzy, to te pieniądze trzeba wykorzystać dla dobra Polaków.

W proponowanym wzroście wydatków państwo w ogóle nie uwzględniacie najważniejszej sprawy, prawdziwego frontu, na którym umierają Polacy, mianowicie systemu opieki zdrowotnej i zapaści w systemie opieki zdrowotnej.

Jest szereg innych programów, które obiecaliście i które nie są realizowane, jak choćby mieszkalnictwo czy restrukturyzacja energetyczna.

Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub Lewicy. Panie pośle, a te poprawki? Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Tam jest ukryta inflacja. Opłata mocowa, czyli to wszystko, za co płacimy w cenie prądu. To nie jest przypadek, że dzisiaj koncerny energetyczne mówią o 40-procentowej podwyżce prądu, ceny energii. To są rzeczy, które na końcu i tak uderzą w nas, czyli uderzą w tych wszystkich, którzy korzystają z usług: chodzą do sklepu, kupują, więc ceny w sposób naturalny będą rosły. Ale ładnie to wygląda, że znalazło się 80 mld zł, ładnie to można w tej chwili opowiadać, ładne story jest. 40 mld zł rozdzielimy na inne zadania.

Sprawy wewnętrzne to 3 mld zł, na samorząd chcecie dać 12 mld zł, ale 8 mld zł to jest ta słynna ustawa samorządowa, natomiast 4 mld zł chcecie podzielić na wodę i kanalizację, ale nie mówicie, na jakich zasadach to będzie dzielone, bo pewnie znowu będzie to jakiś fundusz i znowu przeznaczycie to dla swoich samorządów. Powiem o pierwszych trzech, a za chwilę pan poseł Zandberg powie o poprawkach pracowniczych.

Nie potraficie się dogadać, więc Lewica chce wam pomóc w tym projekcie i w tych poprawkach, żeby je przegłosować. Oczywiście od tego, jak się zachowacie, uzależniamy, jak się zachowamy przy całości nowelizacji budżetu. Pan poseł Adrian Zandberg, klub Lewicy, wykorzysta resztę czasu. Wysoka Izbo! Krótko. Musimy podnieść płace w budżetówce i musimy je podnieść zdecydowanie. Rośnie liczba wakatów, coraz więcej instytucji publicznych boryka się z tym, że nie jest w stanie zrekrutować pracowników. Jeżeli tego nie zrobimy, to państwo polskie będzie działało coraz gorzej i coraz gorzej. Spierałem się tutaj w kuluarach z panem przewodniczącym Kowalczykiem, który twierdził, że jednorazowe, hojnym gestem, wyznaczenie funduszu nagród rozwiąże problem. Panie Przewodniczący! Nie rozwiąże to problemu, trzeba słuchać pracowników, trzeba słuchać związkowców, tych z Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego AD REM, tych z OPZZ-u, tych z Konfederacji Pracy. Oni mówią jasno, że 12% normalnej podwyżki dla całej budżetówki to jest bardzo umiarkowany i skromny postulat, który pokazuje, że związkowcy, że pracownicy myślą o instytucjach, w których pracują, i o ich przyszłości.

Teraz głos ma pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Sytuacja w gospodarce jest dynamiczna, dała określony wzrost gospodarczy.

Wiemy, że mamy jeszcze jeden kwartał.

Słusznie, że podzielono, że częściowo obniżono wysokość deficytu, a jednocześnie przeznaczono na finansowanie pewnych działań. Szkoda, że nie znalazły się działania na rzecz wsparcia zaniedbanego problemu mieszkalnictwa, bo jest to ważne dla polskich rodzin, bo mieszkanie daje stabilizację, wpływa na demografię, młodzi ludzie zostają w Polsce.

Niekoniecznie trzeba dokonywać takiego obniżenia deficytu, stąd nasza poprawka dotycząca tego, żeby deficyt został powiększony o 7 mld, żeby zabrać 3 mld z obrony i 10 mld przeznaczyć na sprawy oddłużenia szpitali powiatowych. Jest taki moment, że jeszcze można utrzymać pewien poziom zadłużenia, bo reguła wydatkowa będzie nas obowiązywała od roku 2023.

Bardzo dziękuję. Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacznijmy od tego, że podatki to kradzież, i chwalenie się przez rząd, że w tym roku wpływy budżetowe wzrosły, to jak chwalenie się przez złodzieja, że w tym roku udało mu się obrabować o kilka domów więcej. Rozumiem, gdybyście się chwalili innym złodziejom, ale państwo się chwalą tym przed obywatelami, których wysokimi, coraz wyższymi podatkami rabujecie w biały dzień - nie tylko podatkami, ale także inflacją. Właśnie w inflacji tkwi odpowiedź na pytanie, skąd te wyższe wpływy. Przez państwa politykę monetarną i fiskalną inflacja szybuje aż do 5% w tym roku i tym samym wpływy z budżetu po prostu rosną, bo rosną ceny w sklepach i rośnie kwota podatków, jakie płacimy, np. za artykuły spożywcze. Dlaczego państwo założyli w ustawie budżetowej na ten rok - rok temu, jak nad nią procedowaliśmy - że inflacja będzie niższa?

Przypomnijmy, w styczniu 2020 r. prezes Glapiński mówił, że nie obawia się ekspertyz analityków mówiących o tym, że inflacja będzie wynosiła 4%.

Przypomnę: mamy 5%. I stąd się biorą te wyższe wpływy budżetowe. Państwo zamiast odpowiedzialnie odpowiedzieć: okej, udało nam się ograbić obywateli z trochę większej ilości pieniędzy poprzez nasze podatki i inflację, to w takim razie zniwelujmy dług tych obywateli, który zaciągnęliśmy. I zamiast obniżyć dług, to państwo stwierdzili: super, mamy więcej pieniędzy obywateli, wydajmy je szybko, zanim ktoś pomyśli o tym, żeby np. obniżyć podatki albo żeby załatać dziurę budżetową.

Zacytuję jeszcze inne słowa: Inflacja to jest jeden z najgorszych podatków, ponieważ jest to taki podatek, który można wprowadzić bez zmiany prawa. A więc państwo mają szereg możliwości na łupienie obywateli.

Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku chyba warto zadać pytanie panu premierowi, a może panu przewodniczącemu Kowalczykowi, który tak się chwalił, że rząd prowadzi wspaniałą politykę gospodarczą. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość, panie przewodniczący, mówi prawdę? Kiedy mówicie prawdę?

Te dwie rzeczy wykluczają się wzajemnie. Albo nie ma pieniędzy i podnosicie podatki, albo są pieniądze i cały ten lament Prawa i Sprawiedliwości to jedna wielka bzdura. A więc, panie premierze, panie przewodniczący, co jest prawdą? Jest też pytanie o rzetelność ustawy budżetowej, bo wartości pokazane na początku roku i te pokazane dziś spektakularnie się rozchodzą, pokazując albo niekompetencję i brak rzetelności, albo zamierzone wprowadzanie w błąd. I też chcemy wiedzieć, cała Polska chce wiedzieć, gdzie leży prawda? Ale trzeba też wyraźnie powiedzieć, że są to pieniądze, które rząd wyciągnął ludziom z portfeli. Z jednej strony szalejąca drożyzna inspirowana niestety przez rząd serią podwyżek, która napędza dochody z podatków, z drugiej strony frywolna polityka Narodowego Banku Polskiego, który spekuluje i pompuje wynik finansowy, zamiast dbać o stabilność pieniądza, żeby inflacja po prostu nie zżerała dochodów i oszczędności Polaków. O tym pan prezes narodowego banku nie pamięta. Pojawiają się nowe środki z praw do emisji CO2. Te środki powinny być znaczone i przeznaczone na zieloną energię, tymczasem wkładacie je do budżetu, zamykacie program wsparcia dla fotowoltaiki. Jeżeli są środki, to ten program dotyczący rozwoju fotowoltaiki powinien zostać wzmocniony. W tym budżecie jest przeznaczone 800 mln zł na Narodowy Fundusz Zdrowia.

To daje 9 mld zł w sytuacji, w której ochrona zdrowia umiera. Co wy w ogóle robicie?

Szanowni Państwo! Koło Parlamentarne Polska 2050 składa poprawki do tego projektu. Proponujemy, aby z obrony narodowej 3 mld zł poszło na ochronę zdrowia. Proponujemy (Dzwonek), żeby tę kwotę przeznaczyć na rzecznika praw obywatelskich. Te dwie poprawki składam na ręce pana marszałka.

Dziękuję bardzo.

Zamykam listę zgłoszonych do pytań. Wyznaczam czas pytania na 1 minutę. Dlaczego nie mogą mieć wprost zapisanych pieniędzy w budżecie: konkretnie ile i na co? Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami muszą ciągle walczyć, ciągle prosić, dopominać się? Jak mają składać jakiś wniosek o dofinansowanie czy do NFZ-u, czy do PFRON-u, to muszą śpieszyć się z tymi wnioskami na początku stycznia, żeby zdążyć, bo potem już tych pieniędzy nie ma. A teraz jak dokładacie te pieniądze w budżecie, np. 200 mln zł, to dajecie je do rezerwy celowej premiera, z której są realizowane różne bardzo istotne zadania typu: jakieś katastrofy związane z żywiołem i inne cele.

Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Chcę zapytać o środki, które pochodzą z handlu emisjami CO2 Te środki powinny służyć modernizacji naszego systemu energetycznego, powinny służyć transformacji energetycznej, inaczej ta energia, którą promujecie, po prostu nas zabije, a kolejne pokolenia będą żyły w świecie, który nie będzie się nadawał do życia na takim poziomie, jaki widzimy dzisiaj. Tymczasem zamykacie ten program, dzięki któremu Polacy mogą u siebie w domu, na domu, w ogrodzie montować panele fotowoltaiczne. Pomimo tego, że tak drastycznie wzrasta kwota, która pochodzi z handlu emisjami, wy tego nie wspieracie, nie chcecie wspierać tej transformacji, chcecie, żeby Polacy dalej umierali czy to z powodu zanieczyszczenia, czy z powodu zmian klimatycznych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chwała. Po kilkunastu dniach przeliczeń mówi: Drodzy Polacy, mamy tych miliardów 80. Jak można ufać takiemu gospodarzowi, który raz liczy tak, raz liczy tak. To teraz jest pytanie. Czy my dobrze rozdajemy te 80, bo jednak może powinniśmy rozdać 30? Ale jeżeli już rozdajemy te 80, to pytam: Kiedy podwyżkę otrzymają nauczyciele? Kiedy podwyżkę otrzymają pracownicy administracji? I w końcu kiedy przestaniecie kupować zabawki dla Ministerstwa Obrony Narodowej za granicą, a będziecie wspierać polskie zakłady zbrojeniowe? Kiedy przestaniecie kupować drony poza wszelką procedurą w Turcji, a rozpoczniecie kupować je w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy? Oczekuję na swoje pytania odpowiedzi na piśmie. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałam zapytać pana ministra o wydatki niewygasające. Pan, człowiek doświadczony, finansista, jak pan może godzić się z tym, że w tej chwili wydatki niewygasające to już jest zasada? Wydatki niewygasające znane są od lat, ale nigdy nie były na takie długie okresy ani też tak ogromne kwoty. Ile na tym stracimy? Z tych 40 mld ponad połowa to wydatki niewygasające, które mogą być wykorzystywane do końca listopada, a te, które pójdą na fundusze celowe, nie wiadomo kiedy, może 2, 3 lata. Jak można tak lekko traktować dyscyplinę finansów publicznych, nie dbać o pieniądze Polaków? Pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Już wiemy, że 80 mld, które niby znaleźliście państwo w budżecie, było tam wcześniej, bo je po prostu schowaliście. Otóż pan premier Morawiecki ma taką strategię, że najpierw pieniądze w budżecie na początku roku chowa, na koniec roku je znajduje i chce uchodzić za cudotwórcę. Natomiast mam pytanie o to, na co te pieniądze i dlaczego w ten sposób mają być wydane. Otóż chcecie państwo w czasie epidemii, kiedy wiemy, jak bardzo jest potrzebna każda złotówka w ochronie zdrowia, wydać zaledwie 1/80 tej kwoty na ochronę zdrowia, natomiast 10 razy więcej chcecie wydać na armię i na służby. Mam pytanie. Czy będziecie państwo do leczenia ludzi w czasie epidemii używać czołgów czy respiratorów? Pan poseł Arkadiusz Marchewka, Koalicja Obywatelska.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dodatkowe pieniądze w budżecie nie są wcale wynikiem jakiejś dobrej polityki gospodarczej, tylko waszych pomyłek w przygotowaniu budżetu. i m.in. tego, że jest wysoka inflacja, bo skoro Polacy płacą więcej za produkty i usługi, to macie więcej pieniędzy z VAT-u do dyspozycji. I największy problem jest w tym, że zamiast wydawać te pieniądze na sprawy najważniejsze, wydajecie na rzeczy, które dziś nie są wcale tak ważne jak służba zdrowia.

Jeżeli gdzieś trwa wojna, to trwa wojna w szpitalach, trwa wojna na SOR-ach i tam trzeba skierować wszystkie niezbędne środki.

Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Przewodniczący Pośle Sprawozdawco! W czasie prac nad ustawą zmieniającą ustawę budżetową na bieżący rok otrzymaliśmy jako parlamentarzyści mailem stanowisko „Solidarności” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ta komisja zakładowa zwraca się do nas z apelem, aby w ustawie budżetowej i ustawie wprowadzającej ustawę budżetową wprowadzić również środki, 6% dodatku motywacyjnego dla pracowników agencji, którzy w okresie pandemii pracują efektywnie i terminowo, obsługując m.in. dodatkowo osiem programów na rzecz wsi i rolnictwa. Wobec powyższego chciałem zapytać pana, prosiłbym pana ministra o odpowiedź na piśmie: W którym miejscu, w jakiej części budżetowej znajdują się środki na dodatki motywacyjne dla pracowników agencji, jaka to jest kwota oraz na jakich zasadach zostanie rozdysponowana?

Szanowni Państwo! W uzasadnieniu do uchwalonych na poprzednim posiedzeniu Sejmu zmian w ustawie podatkowej napisaliście: Kryzys związany z pandemią COVID-19 przekłada się nie tylko na zmniejszenie wpływów budżetowych, ale także na zwiększone wydatki. Z tego względu państwo zmuszone jest do szukania nowych rozwiązań wspierających wzrost nadwyrężonych wpływów budżetowych. Pytania do państwa z Prawa i Sprawiedliwości: Kiedy mówicie prawdę, a kiedy, oględnie mówiąc, mijacie się z prawdą? Gdy mówicie, że nie podnosicie podatków, a jednak przyznajecie się, że szukacie nowych rozwiązań wspierających wzrost nadwyrężonych wpływów, majstrując przy ustawach podatkowych? Czy może wtedy, gdy tuż po podniesieniu podatków znajdujecie w budżecie wolne 80 mld zł? A może wtedy, gdy podnosicie podatki rzekomo z powodu epidemii COVID-19, a potem z cudownie odnalezionych 80 mld zł na ochronę zdrowia przeznaczacie zaledwie 1 mld zł? Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Państwo Ministrowie!

Od 20 dni strajkują pracownicy ochrony zdrowia. Oni nie otrzymają żadnych pieniędzy.

Wprowadzacie stan wyjątkowy i my tego nie zobaczymy. To będzie na zaliczki? Żaden problem nie został rozwiązany. To wstyd. Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po wzburzeniu, jakie usłyszałem, chciałem zadać pytanie, czy podatki to kradzież, ale zorientowałem się, że pytanie polityków o to, czy podatki to kradzież, to jak pytanie się Robin Hooda czy Janosika, czy jest złodziejem. To jest bez sensu, bo w ich oczach są oni po prostu bohaterami.

Proszę chociaż o odpowiedź na takie pytanie. Ale proszę bardzo nie dyskutować. Bardzo proszę państwa posłów o nieprzeszkadzanie w prowadzeniu obrad. Wysoka Izbo! Przyzwyczailiście nas państwo już do takiego bezczelnego samozadowolenia przy przedstawianiu sukcesów waszego rządu, ale muszę powiedzieć, panie pośle, że pan jest jeszcze jajcarz do tego, bo żeby tak sobie przypisywać ten wielki sukces, że te pieniądze wpłynęły, bo wy tak genialnie zarządzacie. A propos tego genialnego zarządzania mam dwa bardzo konkretne pytania: Dlaczego w tym znowelizowanym budżecie nie zostały odłożone pieniądze na zadośćuczynienie, odszkodowania dla ludzi, którzy zgromadzili się w Polskiej Federacji Fitness, którzy wystąpili z protestem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa, którzy dostaną odszkodowania, bo to są te firmy, które w wyniku waszych decyzji w dużym stopniu zbankrutowały?

Jest możliwość. Pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Proszę nie przeszkadzać, pani poseł. Panie Przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Kaczyński! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Apeluję o prawdę o stanie polskiego budżetu. To jaka jest prawda? Z kolei według NIK w 2020 r. sam deficyt wyniósł 81 mld zł, ale deficyt całego sektora instytucji rządowych - aż 161 mld. Według metodologii unijnej dług publiczny w 2020 r. wzrósł aż o 290 mld zł i wynosił włącznie 1336 mld. Która z tych liczb jest prawdziwa?

Wysoka Izbo! Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że tobie zabierze, bo rząd nie ma własnych pieniędzy - mówiła swojego czasu Margaret Thatcher.

Za chwilę jednak Polacy zapłacą gigantyczne rachunki za energię cieplną i sfinansują te fanaberie rządu. I w tej sytuacji, kiedy cały świat walczy z COVID, nasz rząd nie dostrzega potrzeb służby zdrowia. Okazuje się, że to miejsce, w którym toczy się faktycznie wojna, walka o życie ludzkie, jest niedostrzeganym przez rząd PiS aspektem życia społecznego. Dziesięciokrotnie za to więcej wydajecie państwo na armię. Myślę, że to jest jasny dowód na to, jakie są wasze intencje. Pan poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Muszę przyznać, że zupełnie niezrozumiała jest praktyka nieobecności ministra finansów w trakcie debaty dotyczącej budżetu. Po raz kolejny nie ma ministra finansów, do którego mamy konkretne pytania i od którego oczekujemy odpowiedzi, chociażby tej dotyczącej sytuacji w ochronie zdrowia.

Tam niezbędne są płynące szerokim strumieniem środki finansowe, a tego dzisiaj nie mamy, tego dzisiaj nie widzimy w nowelizacji ustawy budżetowej. To jest skandal, taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca. Dlatego składamy stosowne poprawki, ważne poprawki, które zadecydują o naszym kolejnym, dalszym postępowaniu.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 dotyka w gruncie rzeczy nas wszystkich, gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorców. Zwalacie to tak naprawdę na Unię Europejską, a w tle dzięki temu przykrywacie złe zarządzanie w spółkach energetycznych, które jest fatalne i ma istotny wpływ na wzrost cen. Wy mówicie: to nie my za to odpowiadamy. Ale warto w tym kontekście podkreślić to, co już kilka razy tu wybrzmiało: rząd jest gigantycznym beneficjentem tego wzrostu.

Wysoka Izbo! Zawsze jest tak, że opozycja lepiej wie, na co wydać pieniądze, a rządzący zawsze nie wiedzą. Za każdym razem jest tak: jak rządzą tak czy inaczej, to tak jest.

W pewnym czasie przyjdzie zmiana, będą inni odpowiadać.

Mając tyle pieniążków, można było to zrobić, można było np. oddłużyć szpitale powiatowe i dać te podwyżki, o które walczy służba zdrowia.

Wysoka Izbo!

W związku z tym moje pytanie jest proste, bo znając procedurę, to w październiku pewnie dopiero ta nowelizacja będzie formalnie podpisana. W związku z tym jest pytanie, jak wygląda planowanie, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Nie przewiduję, że przez te 2 miesiące, biorąc pod uwagę zapóźnienia, które są, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, uda się wydać 5 mld czy dodatkowe 3 mld na drogi. Czy w tym zakresie te środki będą przechodzić na następny rok, czyli będą to wydatki niewygasające? Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Rosati, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Cała opozycja od Lewicy po Konfederację mówi jednym głosem: służba zdrowia. My, jako Koalicja Obywatelska, złożyliśmy do tej bardzo ważnej ustawy jedną poprawkę, słownie: jedną, o zwiększeniu dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o 10 mld zł. Zgódźcie się na to. My możemy dyskutować, gdy będzie dyskusja o budżecie na przyszły rok, o tym, żeby odpowiednio dostosować wydatki na armię czy na służby, czy na transport kolejowy. Ale ta sprawa jest w tej chwili najważniejsza. Wszystkie są ważne: i koleje, i obronność, ale ta sprawa, sprawa zdrowia i życia Polaków, jest najważniejsza. Pomyślcie jeszcze i zgódźcie się na tę propozycję. Dajcie ten sygnał, wyślijcie ten sygnał. Zlikwidujecie to miasteczko, będziecie postrzegani jako odpowiedzialna władza. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nikt z nas nie jest anarchistą, wszyscy rozumiemy, że w każdym państwie muszą istnieć podatki. Niestety, to, co wy robicie tą propozycją Polskiego Ładu, raczej antypolskiego ładu, jest duszeniem polskiej przedsiębiorczości i sprawieniem, żeby gospodarka zastopowała. Co więcej, chwalicie się co roku dziesiątkami miliardów złotych. Na co poszły przez 6 lat te dziesiątki miliardów złotych? Gdzie jest armia nowoczesna? Wydajecie pieniądze na zabawki z USA, za które nawet Amerykanie nie są wam wdzięczni, mają was gdzieś. Gdzie jest elektrownia atomowa? Jesteście kolejnym impotentnym rządem, który tego nie realizuje przez 6 lat. Mamy katastrofę w energetyce, katastrofę w górnictwie, mamy wysokie ceny prądu.

Teraz głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pan Marcin Ociepa. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Jestem porażony tymi słowami, które tutaj padały w czasie debaty, kiedy państwo podważaliście zasadność wydatkowania środków na obronność. Chcę państwu powiedzieć, że jesteśmy świadkami niestety pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu. Niemal wszystkie państwa NATO podnoszą wydatki na obronność. W naszym regionie państwa czy to skandynawskie, czy bałtyckie podwyższają budżety na obronność o kilkadziesiąt procent rok do roku, a w polskim parlamencie polska opozycja podważa zasadność tych wydatków. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Uprzejmie apeluję o odpowiedzialność i uświadomienie sobie, że bez bezpieczeństwa, w które trzeba inwestować nieustannie, i niestety podnosić na to nakłady finansowe, nie będzie ani tego parlamentu, ani szpitali, ani samorządów, ani kolei, bo nie będzie państwa polskiego, bo nie będzie suwerenności. Teraz głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Sebastian Skuza. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani poseł. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Odpowiadam na pierwsze pytanie dotyczące kwestii osób niepełnosprawnych. Kwota i zadanie, jakie ma być z niej finansowane, myślę, są zauważalne. Wczoraj w Komisji Finansów Publicznych dyskutowaliśmy o roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w tym zadaniu i o tworzeniu wypożyczalni sprzętu. Jak wczoraj już mówiłem, to zostało przygotowane przez pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych pana ministra Pawła Wdówika. Według mojej najlepszej wiedzy Ministerstwo Klimatu jest zobowiązane sporządzać raporty, które przekazujemy do Unii Europejskiej, że wypełniamy postanowienia dyrektywy klimatycznej.

W tym roku właśnie ustawa okołobudżetowa, jej nowelizacja umożliwia utworzenie funduszu motywacyjnego w wysokości 6%.

W czasie pandemii przerwane zostały łańcuchy dostaw, nie mogły być tak sprawnie, jak zakładano, przeprowadzone postępowania przetargowe, więc moim zdaniem jak najbardziej jest zasadne wydłużenie okresu wydatków niewygasających. Gdyby ta poprawka była przyjęta również bez wydatków niewygasających, to nie byłoby możliwe w tak krótkim okresie do zrealizowania. Co do nakładów na służbę zdrowia to przypominam, że w roku 2022 będzie przyspieszenie i nakłady będą stanowić 5,75% PKB.

Co do kwestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to nowelizacja ustawy okołobudżetowej będzie umożliwiać zwiększenie w planach finansowych na wynagrodzenia również agencji wykonawczych. W 2022 r. projekt ustawy budżetowej przewiduje również wzrost wynagrodzeń w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli zapadną takie wyroki. W budżecie państwa zawsze jest tworzona rezerwa na zobowiązania wymagalne i nie kojarzę jakichś przypadków, żeby był prawomocny wyrok i zasądzone środki nie były wypłacone z budżetu państwa w terminie. Co do transparentności finansów publicznych to chciałem przypomnieć, że jesteśmy zobowiązani do podawania wszelkich informacji do Eurostatu według metodologii Unii Europejskiej i te informacje są przekazywane, a dodatkowo nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 11 sierpnia wprowadza zasadę, że cały sektor general government pokazujemy tylko i wyłącznie według metodologii Unii Europejskiej, nie według metodologii Polski. Jesteśmy zobligowani umowami międzynarodowymi do wydatkowania określonej kwoty w relacji do produktu krajowego brutto właśnie na obronność. Co do systemu podatkowego i podatków to twórca ekonomii klasycznej Adam Smith mówił o dwóch rzeczach, które są na zawsze i są pewne, i jedną z tych rzeczy właśnie określał jako podatki. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Po pierwsze, takie bardzo odkrywcze: rząd nie ma własnych pieniędzy. Oczywiście rząd nie ma własnych pieniędzy. Obywatele wybierają większość parlamentarną i rząd i powierzają zarządzanie tymi pieniędzmi. I oczekują, aby to zarządzanie było odpowiedzialne. Wiem, że w poprzedniej ekipie mówiono: pieniędzy nie ma i nie będzie. Dlatego też Polacy powierzyli nam, nie raz, ale i kolejny raz, te pieniądze, bo czują, że te pieniądze obywateli z podatków są dobrze zarządzane, dobrze gospodarowane.

Jeśli pan poseł Kulesza nie jest przekonany, proponuję, aby pociągnąć do odpowiedzialności karnej, począwszy od Mieszka I, wszystkich zarządzających tymi podatkami, skoro mieli owoce z kradzieży.

Proszę się zastanowić nad słownictwem.

Rozumiem, że można takie rzeczy opowiadać, ale jednak apeluję o to, żeby rozmawiać merytorycznie o tym wszystkim.

Zawsze mówię, że liczb się nie oszuka. A jak za liczbami stoją pieniądze, tym bardziej oszukać się nie da. Naprawdę nie opowiadajmy rzeczy, które są zupełnie niestworzone.

Odsyłam wobec tego do ustawy okołobudżetowej, gdzie jest dział: Przepisy epizodyczne. Jest zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pomóżmy tym, którzy nie mają. Mało tego, nie tylko wyszczególnione są gminy, które mają to otrzymać.

Zamożniejsze gminy - mniejszy współczynnik, mniej zamożne - trochę więcej tych pieniędzy w przeliczniku. 3 mld na kanalizację - w sposób identyczny, tylko tu próg dostępu do kanalizacji jest obniżony do 60%. Zatem te gminy, które mają powyżej 60% dostępności, nie będą brały udziału w tym podziale. Gdzie tu uznaniowość, panie pośle? Proponowałbym, żeby jednak, zabierając głos i krytykując.

Mało tego, ustawa wręcz gwarantuje, że nie może być mniej niż było w roku poprzednim. Każdy samorząd jest przyzwyczajony do tego, żeby zawsze płakać. Zawsze im mało. Ja to rozumiem, bo każdy samorząd chciałby jak najwięcej pieniędzy, ale w tym przypadku wszystkie ubytki są pokryte. Samorządy różne rzeczy mówią. Nie warto powtarzać. Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do obu projektów ustaw poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie te projekty do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.